Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Bardzo proszę, pan poseł Borys Budka.

By stanął tutaj wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wytłumaczył się przed Polakami z tego bezprawnego użycia siły wobec protestujących kobiet, z tego, że naraża zdrowie i życie Polaków na niebezpieczeństwo [[Oklaski]] - a dzisiaj nawet nie ma odwagi przyjść do Sejmu. Ale chcę z tego miejsca zapowiedzieć, że pan, panie Kaczyński, nie schowa się przed Polakami, że tutaj będzie pan musiał przyjść i się wytłumaczyć.

Ooo! ...musiała Wysoka Izba rozpatrzyć. I wreszcie po tylu latach niszczenia Polski pan Kaczyński będzie musiał stanąć tu.

wszystkich państwa - także tutaj - o spokój, żebyśmy mogli zacząć procedować. Wniosek przeciw, proszę bardzo. Bardzo pana proszę.

Proszę bardzo. Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym. wydarzyła się rzecz niesłychana. Z mównicy Sejmu usłyszeliśmy, że jesteśmy godni tego, żeby skończyć w więzieniu. Ale w więzieniu skończą ci.

Domagamy się informacji, bo składamy również wniosek o wotum nieufności dla premiera Kaczyńskiego. Koniec odpowiedzialności za niebezpieczeństwo.

Proszę bardzo, pan poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od wczoraj mamy do czynienia jednak z kuriozalną sytuacją. Dzieją się rzeczy straszne.

Pani jest marszałkiem nie swoich, tylko polskiego Sejmu. Pani powinna reagować na to, jeżeli posłowie przychodzą tutaj i mówią, że są przepychani przez policję, niewpuszczani do Sejmu (Dzwonek), że policja ich legitymuje. Złożył pan wniosek formalny o przerwę, panie pośle. Przegłosujemy ten wniosek. Pani Marszałek! Pani powinna stać na straży polskiego Sejmu. Pani powinna otoczyć opieką każdego parlamentarzystę, [[Oklaski]] niezależnie od tego, z jakiego jest klubu. Jeżeli pani nie żąda wyjaśnień od policji, od pana posła Kaczyńskiego, od pana Wąsika, od pana Kamińskiego na temat tego, co zdarzyło się wczoraj, to naprawdę ogranicza pani swoją władzę. Pani marszałek, my tylko prosimy panią o to, żeby była pani marszałkiem polskiego Sejmu, a nie marszałkiem PiS-u.

Padł wniosek formalny o przerwę, w związku z tym ten wniosek poddam pod głosowanie.

W takim razie pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, wniosek formalny. Szanowna Pani Marszałek! Wczoraj mieliśmy do czynienia z rzeczą niesłychaną w tej Izbie, ponieważ pan poseł Gawłowski... Gawkowski.

Jak się okazuje, prawda jest zgoła inna. W związku z tym zwracam się do pani marszałek z prośbą o to, [[Oklaski]] aby do czasu wyjaśnienia tej sytuacji pan wicemarszałek Czarzasty nie prowadził obrad Wysokiej Izby, nie uczestniczył w posiedzeniach Wysokiej Izby.

Panie pośle, o tym, kto będzie prowadził obrady Sejmu, decyduje marszałek, w związku z tym proszę. Ale panie pośle, czy może pan w tej chwili nie dyskutować ze mną?

Proszę państwa, chciałam państwu udzielić informacji na temat tego, co się wczoraj wydarzyło. Ale państwo składacie wnioski formalne, więc zaczekam cierpliwie do wyczerpania wniosków formalnych i udzielę państwu informacji. W tej chwili te wnioski formalne nie są wnioskami formalnymi - na razie, póki co, z wyjątkiem jednego o przerwę. Najpierw. Panie pośle, do wniosków formalnych nie ma sprostowań, bo to były wnioski formalne. Wysoka Izbo! Wnoszę o odroczenie obrad do czasu, aż pan minister Kamiński i pan wicepremier Kaczyński przygotują informację na temat wczorajszego dnia. Bo wczorajszy dzień był szczególny. Wczorajszy dzień to był dzień przeglądania się trochę w lustrze. To znaczy najpierw pan wicepremier Kaczyński przeglądał się w lustrze i zobaczył tam ewidentnie twarz naszego posła Grzegorza Brauna bez maseczki, skoro wchodząc tutaj, na mównicę, ją zdjął.

Wyszła wasza hipokryzja, kiedy zamaskowani funkcjonariusze wchodzą do tłumu, kiedy prowokują, kiedy wyciągają pałki teleskopowe. Kiedy to dotyczy Marszu Niepodległości, to oczywiście wy klaszczecie, kiedy to dotyczy was, to oczywiście płaczecie.

Padł wniosek o odroczenie posiedzenia. Proszę bardzo. Panie pośle, mam nadzieję, że pan będzie miał wniosek formalny. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mam wniosek formalny o to, żeby pani marszałek ludzi, którzy składają wnioski, które nie są formalne, pod pretekstem formalnym, karała odbieraniem głosu. Proszę państwa, padły dwa wnioski formalne. Jeden - o przerwę, drugi - o odroczenie posiedzenia. W związku z tym głosujemy. Poddam ten wniosek pod. Proszę państwa, proszę o spokój. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść

Sejm wniosek odrzucił. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolicie, parę słów wyjaśnienia po tym, co się wydarzyło wczoraj. Dzisiaj te obrady są trochę późniejsze ze względu na to, że postanowiłam zapoznać z sytuacją przede wszystkim Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, ale też państwu chciałam przekazać informacje, przy czym od razu zaznaczam, że to nie podlega żadnej dyskusji, przechodzimy potem do realizacji porządku dziennego.

Ogłosiłam przerwę i natychmiast przystąpiłam do sprawdzenia tej informacji, bo ona jest bardzo ważna.

Proszę państwa, ja się nie odnoszę do tego, co było podczas całego zgromadzenia, tego, które było na ulicy, nielegalnego, nawiasem mówiąc, państwo o tym wiecie. Nie wiem, co było przez cały czas. Jeżeli państwo nie chcecie słuchać wyjaśnień, to proszę powiedzieć. Trzykrotnie rozmawiałam z komendantem, natychmiast wystosowałam pismo, żądając wyjaśnienia od komendanta głównego, powołując się na konstytucję i na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, mówiące o tym, że otrzymałam informację o zatrzymaniu i o fizycznym.

W tym piśmie od komendanta głównego była informacja o tym, że pan wicemarszałek Czarzasty razem z dwiema innymi osobami, jak się potem okazało, posłami, chciał się dostać na teren Sejmu. Policja wykonywała swoje zadania, proszę państwa, bo takie miała zadanie - ochraniać Sejm, zapewnić. Proszę państwa, naprawdę przerwę, jeżeli państwo nie chcecie słuchać. Albo pan wysłucha tego, co mam do powiedzenia, albo państwo nie chcecie tego słuchać. Proszę mi to powiedzieć.

To trochę trwało, trzeba to było zgrać, trochę oczyścić, żeby zobaczyć, jak to wyglądało, co się działo. Rzeczywiście na nagraniu, które też dzisiaj puściłam - to jest nagranie z tego momentu, jeszcze raz mówię, nie z całego przebiegu obecności państwa na tej manifestacji, bo niestety nie mam takiej możliwości, żeby obserwować, co się dzieje z posłami na tych manifestacjach - ewidentnie widać, że pan marszałek nie został przez nikogo pobity, nie został zatrzymany. Pani poseł Żukowska pokazała legitymację i widać na filmie, jak spokojnie przechodzi do Sejmu. Druga posłanka - czy poseł, już w tej chwili nie pamiętam, czy to była pani, czy pan - również okazała legitymację i też została przepuszczona.

Ale pan marszałek nie wszedł do Sejmu, tylko rozpoczął dyskusję, rozmowę z policjantami. Proszę państwa, z pisma, które otrzymałam od komendanta głównego, wynika, że w trakcie. Panie pośle Kaleta, bardzo pana proszę - żebym mogła kontynuować, dobrze? W tej informacji, którą otrzymałam na piśmie od pana komendanta głównego.

Nie oceniam tego, panie przewodniczący.

Proszę państwa, dzisiaj słuchałam wypowiedzi rzecznika prasowego komendy Policji, który wyjaśniał tę sytuację.

Chciałabym być o tym wtedy poinformowana.

Będziemy wyjaśniali ten incydent, bo to są rzeczy niedopuszczalne. Przedstawiciele władzy, szanowni państwo, muszą zachowywać się zgodnie z pewnymi procedurami i okazywać szacunek funkcjonariuszom państwa polskiego, jakimi są policjanci, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe w imieniu państwa polskiego. Chcę państwu jasno powiedzieć.

Ten wniosek jest źle skierowany. To ja od samego początku jako minister spraw wewnętrznych codziennie w pełni sprawuję realny nadzór nad formacjami mi podległymi, w tym nad polską Policją.

Panie ministrze, bardzo przepraszam, sekunda.

Moim celem nie jest podgrzewanie atmosfery ani na tej sali, ani w kraju. Jako minister spraw wewnętrznych mam swoje obowiązki państwowe, które wykonuję. To ja, jeszcze raz chcę to podkreślić, od momentu dużego wybuchu społecznego, jaki nastąpił po 22 października, czyli po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, na bieżąco nadzoruję działania podległych mi służb, w tym Policji. Ponoszę pełną odpowiedzialność, każdego typu, w tym polityczną, co oczywiste, za działania Policji. Uważam, że były to działania podjęte w interesie państwowym, w interesie wszystkich obywateli. To, że Policja jest dziś atakowana zarówno z lewej strony, zarówno przez was, jak i przez was, świadczy o jej bezstronności.

Po pierwsze, zabezpieczyć stabilność państwa, uniemożliwić destabilizację państwa, a tym samym.

Kiedy będziecie mieli głos, będziecie mogli komentować moje słowa i działania służb mi podległych. Pierwszym, podstawowym celem w sytuacji pandemii, kiedy mamy do czynienia z ogromnymi społecznymi protestami, jest zabezpieczenie w sposób korzenny bezpieczeństwa państwa, a tym samym swobody funkcjonowania wszystkich instytucji publicznych.

To był cel policji. Dlatego tu stała i dziś też tutaj stoi. Bo takie były zapowiedzi organizatorów - zablokować Sejm, uniemożliwić nam pracę, nam jako parlamentarzystom, wam jako parlamentarzystom. Szanowni państwo, drugim celem, jaki postawiłem policji w związku z tym, że emocje społeczne były ogromne, było niedopuszczenie do fizycznej agresji między poszczególnymi grupami demonstrantów. Często mieliśmy do czynienia ze zorganizowanymi grupami szkolonymi do walk ulicznych, związanymi ze skrajnie lewicowymi środowiskami. Przedstawię w odpowiednim momencie też precyzyjną informację co do szkoleń dotyczących walk ulicznych. Proszę państwa, niezależnie od tego, jakie poglądy były głoszone na ulicy, policja zawsze stosowała te same zasady. Niezależnie od haseł działania policji miały być i były stanowcze tam, gdzie trzeba działać stanowczo, i zdecydowane punktowo tam, gdzie trzeba było działać zdecydowanie, gdzie mogła polać się krew niewinnych ludzi, którzy wyszli na ulicę, by demonstrować swoje poglądy. W całej Europie Zachodniej dochodzi do różnego typu gwałtownych sytuacji ulicznych. Spójrzcie, co się dzieje w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech.

W Polsce doszedł nowy temat - temat aborcji. Ważny temat, który dzieli społeczeństwo. Przepraszam. który dzieli społeczeństwo. Szanowni państwo, chcę powiedzieć jasno: Rozumiem protestujących. Nie akceptuję jako polityk i jako człowiek formy tych protestów, jednak rozumiem, że wielu ludzi uznało, że musi zaprotestować i wyrazić swoje poglądy w tej sprawie. Ale oprócz wielu młodych ludzi, którzy byli na ulicach w tej sprawie, mieliśmy grupy skrajne, grupy, które wzywają wprost do obalania konstytucyjnych organów. W Polsce tylko w jeden sposób można zmienić władzę - tylko demokratyczne wybory o tym decydują. Jeden z elementów tych demokratycznych wyborów mieliśmy kilka miesięcy temu. Uszanujmy to wszyscy. Nie będzie w Polsce żadnej rewolucji, nie dopuścimy do tego. Rewolucji rozumianej nie w sensie politycznym i ideowym, bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Sejm, Senat, rząd i

I polska policja tego dopilnuje.

W trakcie tych gwałtownych wystąpień, z którymi mieliśmy do czynienia, policja ochraniała również protestujących - mimo fatalnej, nieakceptowalnej formy tych protestów - przed bandytami, którzy mogli spowodować, że krew niewinnych ludzi będzie przelewana na polskich ulicach. Tak, policja to uniemożliwiła, w tym funkcjonariusze po cywilnemu, którzy zawsze są, którzy mają obowiązek pilnować, żeby ci agresorzy - pojedyncze osoby, które są w tłumie i które myślą, że są anonimowe i bezkarne - nie przyczynili się do tragedii. Było tak i 11 listopada, i wczoraj, i na każdym większym zgromadzeniu - w czasach, kiedy rządziła Platforma, też.

Proszę zachować emocje na wodzy. Teraz chcę nawiązać do sprawy kościołów.

Dla wielu Polaków kościoły i msze to rzeczy niebywale ważne. Państwo polskie musi zagwarantować.

ale gdyby tak się złożyło, że jakaś grupa agresorów niszczyłaby cerkwie prawosławne czy żydowskie synagogi, z taką samą stanowczością będziemy egzekwowali prawo tych obywateli do swobodnego wyznawania swojej wiary i do nieobrażania ich uczuć religijnych.

Chcę do państwa zaapelować, do was, parlamentarzystów: Tu jest wasze miejsce pracy, nie na ulicy. Nie organizujcie swoich pseudointerwencji poselskich.

Szanowni Państwo! Mówicie, że policja wczoraj działała brutalnie. Na tym, że legitymowano osoby, które biorą udział w nielegalnych zgromadzeniu i dopuszczają się wykroczeń? Tak, dopuszczają się wykroczeń.

To wy prowokujecie, wy obrażacie godność polskich funkcjonariuszy, polskiej Policji. Do swoich małych gierek politycznych wprowadzacie element. ataku na innych funkcjonariuszy publicznych, jakimi są policjanci, którzy dobrze wykonują swoją pracę dla całego społeczeństwa, którzy są na pierwszej linii.

Wykazują się niezwykle wysokim morale i poczuciem służby dla wszystkich obywateli. że chronione są prywatne posesje ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiadam wam tak: jeżeli 30 tys. ludzi będzie szło pod wasz dom, wykrzykując nienawistne hasła. Powiem państwu, że w czasie 11 listopada w Internecie pojawiły się głosy, że pójdziemy pod dom Trzaskowskiego. Komenda stołeczna nawiązała kontakt z prezydentem i była tam ochrona policji na wszelki wypadek.

Chcę jasno powiedzieć, że wprowadzanie tak wielkich emocji jest nieodpowiedzialne.

Z tego tytułu policja podejmuje kroki porządkowe, często spotykając się z agresją ze strony osób legitymowanych. Często funkcjonariusze są obrażani, atakowani fizycznie. bo niektórzy mają fałszywe poczucie bezkarności właśnie z powodu tego parasola politycznego, jaki dajecie im swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami. Jeżeli ktoś decyduje się dopuszczać się wykroczeń, łamać przepisy sanitarne, ponosi konsekwencje w postaci mandatu. Nie ma agresji, nie ma tłumienia jakichkolwiek protestów politycznych z uwagi na ich charakter. Obowiązują ogólne, dotyczące wszystkich, niezależnie od tego, jakie poglądy są głoszone w trakcie zgromadzeń, obostrzenia wynikające z epidemii. To jest oczywiste. W wielu krajach Unii Europejskiej jest godzina policyjna, szanowni państwo, jest zakaz jakichkolwiek zgromadzeń, jest możliwość wychodzenia z domu tylko do pracy. Przestańcie manipulować emocjami młodych ludzi. Oni mają swoje poglądy, ja te poglądy szanuję, ale forma tych protestów, to, że się gromadzą, że narażają siebie, swoich najbliższych, swoich sąsiadów, swoich kolegów, jest nieakceptowalne państwowo. Będzie czas na dyskusję polityczną i na szukanie politycznych rozwiązań - nie policyjnych rozwiązań, ale politycznych rozwiązań - wszystkich ważnych problemów, które nurtują naszych wyborców. Dziękuję, panie ministrze.

To nie jest punkt porządku dziennego, żebyśmy prowadzili debatę, więc bardzo proszę, rozumiem, że chce się pan.

Proszę bardzo. Proszę państwa, jestem takim samym parlamentarzystą jak wy po tej stronie i po tej stronie. Mam takie same prawa jak wy i mam takie same prawa bronić tych praw, naszych praw. Panie Ministrze! Nie powiedział pan prawdy na temat tego wydarzenia, dlatego że sytuacja, proszę państwa, była taka. I muszę tę informację przed państwem złożyć. Chciałem wejść na teren Sejmu, ze mną były posłanki, byli ludzie, którzy mi towarzyszyli. Podszedłem do kordonu policji, przedstawiłem się, poinformowałem, że nazywam się Włodzimierz Czarzasty, poinformowałem, że jestem wicemarszałkiem Sejmu. Ponieważ nie miałem legitymacji, to pani posłanka Żukowska wyjęła swoją legitymację, pokazała tę legitymację, poinformowała, że jest posłanką, oraz zaświadczyła, pokazując ten dokument, złożyła oświadczenie, że jestem marszałkiem i jestem posłem.

Od tego momentu policjanci, nawet jeżeli mnie nie poznali, a nie jestem za bardzo zarozumiały - mogli mnie nie poznać. W międzyczasie nastąpiła taka sytuacja: po pierwsze, zostałem zatrzymany, po drugie, zostałem pchnięty na maskę samochodu, po trzecie, jak zostałem pchnięty na tę maskę samochodu, poczułem uderzenie z tyłu, w plecy. Zostałem unieruchomiony siłą. I zostałem pozbawiony wolności. Taka sytuacja nastąpiła. Film, który pokazała pani marszałek, jest od momentu, kiedy to się już wydarzyło. Po tym wydarzeniu podeszła ochrona sejmowa, strażnicy, i jak powiedzieli, że jestem posłem, dopiero zostałem puszczony.

Pani posłanka z Koalicji Obywatelskiej... Wielichowska. Wielichowska dała swoją legitymację, która została złamana. Proszę państwa, chcę wam powiedzieć, że to nie jest, panie ministrze, zachowanie godne policji. Wczoraj powiedziałem, że nie będę oskarżał tego policjanta, który mnie pchnął. Ale chciałem powiedzieć jasno, że wobec dzisiejszej sytuacji, wobec sytuacji, że dzisiaj rano dowiedziałem się, że pobiłem policjanta.

Nie było pokazane, chociaż pani mówiła: to jest ten moment, kiedy pan marszałek pchnął policjanta, Chciałem wam powiedzieć, że mam 60 lat. Jeżeli bym się dowiedział. Chciałem powiedzieć tak: wczoraj, panie ministrze, wielu policjantów biło ludzi pałkami teleskopowymi.

Musi pan być uczciwy w tych rzeczach, które pan mówi.

Chciałam państwu powiedzieć, że nie może tak być. Przystępujemy do realizacji normalnego, zaplanowanego porządku dziennego.

Projekty to odpowiednio druki nr 755, 749, 754 i 753. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu oraz w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 7-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 737. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, druk nr 742. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Dziękuję. Pani Marszałek! Mam zaszczyt zaprezentować projekt uchwały Sejmu w istocie wzmacniający mandat negocjacyjny dla premiera polskiego rządu i polskiego rządu w rozmowach o Wieloletnich Ramach Finansowych. Bardzo krótko zrelacjonuję zapisy tego projektu uchwały. W art. 1 są przedstawione podstawowe ramy prawne, które Sejm pragnie przypomnieć i podkreślić. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym i suwerennym państwem prawa, to jest odwołanie do art. 2 polskiej konstytucji, ale także odwołanie do zapisów preambuły polskiej konstytucji, mówiącej także o tym, że Rzeczpospolita Polska stanowi wspólnotę polityczną wszystkich obywateli. Zapis z pkt 2 odwołuje się do Traktatu akcesyjnego, do traktatu o Unii Europejskiej, podkreśla, że Rzeczpospolita Polska i jej obywatele mają prawo do poszanowania swoich praw i suwerenności na równi z wszystkimi innymi państwami i ich obywatelami zgodnie z art. 2 i 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

W pkt 4 wskazana jest zasada niedyskryminacji, która obowiązuje z jednej strony wobec obywateli, ale z drugiej strony niedopuszczalna jest także dyskryminacja wobec państw członkowskich, stosowanie wobec nich różnych standardów postępowania. W pkt 5 i 6 wskazane są przykłady, które budzą poważne wątpliwości z przeszłości działania Komisji Europejskiej.

Nigdy nie zgłaszano zastrzeżeń do funkcjonowania tego ciała. Taki upolityczniony system wybierania sędziów istnieje również we Francji, w Irlandii, w Hiszpanii, w Austrii. Do tych wszystkich rozwiązań ustrojowych nie zgłaszano w przeszłości żadnych zastrzeżeń ze strony instytucji europejskiej. Nie ma tu takich samych standardów. Ale proszę też, żeby nikt nie żądał tego, żeby nas karać za system ustrojowy wyboru sędziów. Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej to zasada przyznania mówiąca o tym, że jeżeli jakaś kompetencja nie została przyznana Wspólnocie Europejskiej, Unii Europejskiej, pozostaje ona w gestii państwa członkowskiego. Przypominam, że kompetencja co do decydowania o reformie wymiaru sprawiedliwości czy też o kształcie wymiaru sprawiedliwości nie została nigdy przekazana na poziom europejski, więc pozostaje w gestii państwa członkowskiego. W pkt 10 mówimy o tym, że liczne wypowiedzi polityków z wielu europejskich krajów nie pozostawiają wątpliwości, że to Polska ma się stać celem takich działań.

Trudno o bardziej trafne zdradzenie intencji, jaka stoi za tego rodzaju działaniami. I wreszcie, mając na uwadze te aspekty prawne, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej... tutaj chcieliśmy jedną rzecz wyjaśnić: będzie poprawka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości usuwająca pkt 1, ponieważ chcemy jasno wskazać, że weto nie jest celem samym w sobie, weto jest narzędziem do tego, żeby ostatecznie osiągnąć negocjacyjny sukces. My nie chcemy niczego blokować, ale nie możemy dopuścić, by to Komisja Europejska zablokowała dobry budżet dla Polski. Dlatego apelujemy do wszystkich sił politycznych, aby w tej sprawie była jedność. Szanowni Państwo! Odpowiedzcie sobie na pytanie: Czy wy chcecie wzmocnić mandat premiera Mateusza Morawieckiego w tych negocjacjach. czy chcecie wzmocnić mandat Komisji Europejskiej w tych negocjacjach? o wydawaniu środków decydowały instytucje europejskie? Czy państwo chcecie, żeby, tak jak powiedział pan premier Morawiecki, nasz los leżał w naszych rękach, czy też państwo chcecie, żeby było tak, jak powiedziała pani przewodnicząca Katarina Barley, chcecie państwo „zagłodzić” [[Dzwonek]] niektóre kraje w imię politycznych celów? Pani marszałek, ostatnie kilka zdań. Szanowni Państwo! Rok 2020 to rok szczególny. To rok z jednej strony pandemii, z drugiej strony rok 40-lecia „Solidarności” Polska, Polacy mają w sobie ten szczególny gen solidarności. Chcemy, by ten polski gen solidarności stał się genem solidarności europejskiej. Chcemy budowy takiej solidarnej, sprawiedliwej Unii Europejskiej, także w zakresie, w aspekcie jej finansów, jej budżetu, która będzie dobra dla Polski, będzie dobra dla innych państw Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę pana posła Borysa Budkę o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały zawartego w druku nr 749. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak naprawdę ta dzisiejsza debata dotyczy bezpieczeństwa Polek i Polaków. Ta dzisiejsza debata dotyczy tego, czy będziemy w stanie dalej budować wielki europejski projekt, który opiera się na solidarności, bezpieczeństwie, współpracy, poszanowaniu wartości i wzajemnym szacunku i tolerancji. I nie bez przyczyny od 5 lat ten rząd, krok po kroku, wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo Unia Europejska to zasady, to wartości, to przede wszystkim reguły, które są równe dla wszystkich. Niestety państwo udowodniliście, że wasz interes polityczny, wewnętrzne rozgrywki, walka o władzę i o pieniądze, które tak bardzo kochacie i które was tak bardzo łączą, są ważniejsze niż bezpieczeństwo Polaków. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, że opozycja, wspólnie, zarówno klub Koalicji Obywatelskiej, klub Lewicy, jak i klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej, chce zadeklarować wsparcie dla tego rządu, wsparcie dla rządu w sytuacji, w której mówimy o miliardach złotych dla Polski. Od samego początku podkreślaliśmy: fundusz odbudowy, na który zgodził się premier Morawiecki jeszcze w lipcu, to gwarancja, że jesteśmy w stanie wspólnie wyprowadzić Polskę z kryzysu gospodarczego - wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej. Odwołujecie się do solidarności, ale absolutnie nie rozumiecie tego słowa, dlatego że dla was solidarność oznacza solidarność wyciągania kasy z kieszeni polskich podatników. Wiecie, co oznacza praworządność? Praworządność oznacza, że nie będziecie mogli bezkarnie kraść, że kolejny kolega pana ministra nie wyciągnie z pieniędzy polskich podatników milionów złotych na lewe maseczki, respiratory czy lewe testy. Praworządność oznacza, że nie będziecie mogli w sposób bezkarny. Praworządność oznacza, że nie będziecie bezkarnie, w sposób systemowy, sięgać do kieszeni polskich podatników, kiedy obsadzacie kolejne spółki Skarbu Państwa. I wreszcie praworządność oznacza, że będziecie pod kontrolą. Przejęliście prokuraturę, żeby móc bezkarnie umarzać postępowania w sprawie dwóch wież, żeby chronić gangsterów, którzy próbowali przez KNF zagrabić polskie banki. Zbudowaliście system bezkarności i dzisiaj chcecie tę bezkarność kontynuować nawet pod groźbą utraty pieniędzy europejskich. Ale, szanowni państwo, dziś opozycja mówi jednym sło... jednym... tą samą myślą. Jesteśmy po stronie Polek i Polaków. Dziś wspólnie przedłożyliśmy trzy projekty uchwał, które wspierają polski rząd. I w tej Izbie, gdybyście tylko byli na tyle odważni, by odrzucić ekstremizmy tzw. Solidarnej Polski - ludzie, o których jeszcze niedawno mówiliście, że cóż, nie mają kompetencji, ale musieliście gdzieś ich upchnąć w tych ministerstwach - gdybyście odrzucili ekstremizmy, bylibyśmy w stanie zbudować dobre porozumienie. Bylibyśmy w stanie zbudować dobre porozumienie dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, dla polskich rolników, dla samorządowców, dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, dla przedsiębiorców, którzy dzisiaj cierpią z powodu skutków kryzysu gospodarczego. Chcemy uchwały, która będzie wspierać polski rząd, który pokaże, że tak jak kiedyś w tej Izbie potrafiliśmy wspólnie zaakceptować dobry traktat lizboński, tak jak wspólnie potrafiliśmy głosować w sprawach kluczowych dla Polski, tak i dzisiaj chcemy wsparcia dla dobrego budżetu europejskiego. I dzisiaj musicie odpowiedzieć sobie na proste pytanie: Co jest dla was ważniejsze, racja stanu, bezpieczeństwo Polek i Polaków czy bezkarność, której chce wasz pseudominister pseudosprawiedliwości? Dzisiaj, panie premierze, mógł pan uzyskać w tej Izbie szerokie poparcie, odrzucając skrajności, odrzucając ludzi, którzy mają takie pojęcie o praworządności jak Jarosław Kaczyński o demokracji i poszanowaniu praw człowieka. Ale pan, panie premierze, szantażowany przez własny obóz władzy, idzie pod prąd całej Unii Europejskiej. Dziś znowu idziecie na ścianę, dziś znowu wpadliście w ten korkociąg i ziemia jest tuż przed wami. Apeluję do was w imię interesu narodowego: zatrzymajcie się. Porozmawiajmy, jak ten dobry budżet wykorzystać dla Polek i Polaków. Nie straszcie Polaków Unią Europejską, nie wyprowadzajcie Polski z Unii Europejskiej. Po raz kolejny wzywam was do tego, by w sprawach kluczowych mówić jednym głosem. I daję gwarancję, że jeżeli pan, panie premierze, przedłoży w Wysokiej Izbie do ratyfikacji zwiększony budżet europejski o fundusz odbudowy, to będzie szerokie porozumienie, poparcie. Niech pan wreszcie będzie raz odważny. Niech pan to zrobi, nawet z konsekwencjami we własnym obozie władzy. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę pana posła Krzysztofa Gawkowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały.

Przepraszam państwa, ale taką dostaliśmy.

Bardzo proszę, pan Krzysztof Gawkowski, druk nr 754. Wysoka Izbo! Unia Europejska to nasza wspólna rodzina, w której mamy nie dzielić się tylko środkami finansowymi, ale również dzielić się wartościami. Unia Europejska, która ma nas łączyć w praworządności, demokracji, przestrzeganiu regulacji. Taką Unię wybraliśmy w roku 2004 i w takiej odnaleźliśmy się przez ostatnie 16 lat. Budowaliśmy wspólnotę, która miała nam dawać poczucie sprawiedliwości, i przez lata Unia to poczucie nam dawała. Dzisiaj Unia Europejska może czuć się zdradzona, ale nie przez Polki i Polaków, a przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który w ramach swoich interesów chce odmówić Polakom dostępu do środków finansowych, chce zaprowadzić nas w miejsce, w którym każda Polka i każdy Polak... ich portfele zostaną puste. To, co proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, to autostrada do katastrofy. 100 mld zł - tyle możemy stracić, jeżeli uchwała autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zostanie przyjęta. Ale to nie są pieniądze Prawa i Sprawiedliwości, to są pieniądze nas wszystkich, dlatego Lewica zaproponowała uchwałę Sejmu, w której mówimy jasno: polskim interesem stanu jest przyjęcie uchwały, w której będziemy walczyli o każdą złotówkę, nie zawetujemy budżetu, a postaramy się, żeby środki trafiły wszędzie tam, gdzie trzeba walczyć z pandemią, gdzie trzeba odbudowywać gospodarkę, gdzie trzeba jasno i czytelnie mówić, że trzeba więcej pieniędzy na infrastrukturę. Uchwała Lewicy ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa każdej obywatelki i każdego obywatela. Pieniądze, przez które wy się w Unii Europejskiej kłócicie, są dla nas standardem bezpieczeństwa, i o tym powinniście pamiętać. Panie Ministrze! Odpowiedzialność za to, czy chcecie wetować, czy nie, to nie jest odpowiedzialność PiS-u, to jest odpowiedzialność za Polskę, i dlatego Lewica zrobi wszystko, żeby te pieniądze dotarły do obywateli. Jeżeli wy Polaków i Polki okradniecie, my te pieniądze do budżetów samorządów ściągniemy. To będzie trudniejsza, bardziej okrągła droga, ale nikt nie zostanie z tych pieniędzy ograbiony. Samorządy gmin, powiatów, województw mają prawo do tego, żeby swoim obywatelom pomagać. Jeżeli wy tego nie załatwicie, to w Europie przez eurodeputowanych Lewicy przy współpracy z innymi grupami będziemy właśnie o taką procedurę lobbować. Co wy dzisiaj chcecie zrobić Polkom i Polakom? Chcecie im wmówić, że tutaj na sali walczycie o sprawiedliwość i samorządność. Chcecie im wmówić, że walczycie o solidarność, o korzenie Unii Europejskiej, tyle że te korzenie to nic innego jak brak waszego pomysłu na to, jak wybronić się z procesu praworządności, który został przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości wdrożony. Unia Europejska to ojczyzna nas wszystkich, a to znaczy, że odpowiedzialnie musimy walczyć o każdego obywatela.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie, nie, 5 minut jest jako prezentowanie, a w dyskusji klubowej 7 minut. Bardzo proszę pana posła Andrzeja Grzyba o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały zawartego w druku nr 753. Wysoka Izbo!

Ta wspólnota w ponad 80% jest przekonana o tym, że polska obecność w Unii Europejskiej jest wartością, której należy bronić. Elementem tej naszej obecności jest również to, co się dzieje w sprawach dotyczących podstawowych zasad jej funkcjonowania, w tym również kształtowania wieloletniego budżetu i wszystkiego tego, co jest związane z polityką gospodarczą, ekonomiczną, z regulacjami, które mają być tworzone we wspólnocie 27 państw członkowskich. Chciałbym powiedzieć, że w projekcie uchwały przedłożonym przez posłów Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego wzywamy prezesa Rady Ministrów do przyjęcia wieloletnich ram finansowych, bowiem uznajemy, że kwoty wynegocjowane w wieloletnim budżecie oraz w funduszu odbudowy są w obecnej sytuacji szansą na rozwój Polski i odbudowę polskiej gospodarki, która poniosła i jeszcze będzie ponosiła ogromne straty.

Ten spór jest żywy do dzisiaj. Myślę, że to powinna być główna argumentacja, że powinniśmy ratować byt ekonomiczny wielu przedsiębiorców, rolników, wspólnot samorządowych, szpitali - bo to leży w interesie Polaków. 21 lipca Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu oraz funduszu odbudowy, które zostało ogłoszone przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jako sukces negocjacyjny polskiego rządu. Integralną częścią porozumienia liderów, jak wtedy mówiono, była decyzja o wzmocnieniu kontroli nad środkami unijnymi. Zatem wyraziliśmy zgodę na warunkowość. Zapowiedź weta, którą słyszeliśmy ze strony pana premiera Morawieckiego, może zablokować powstanie funduszu odbudowy, który ma pochodzić z emisji długu na jego sfinansowanie, na co pan premier 21 lipca również w imieniu Polski, w imieniu polskiego rządu wyraził zgodę. Fundusz odbudowy jest oczekiwany przez państwa członkowskie, w tym przez Polskę. Nikt tego nie kwestionuje, również na tej sali.

Zarówno w wieloletnich ramach finansowych, jak i w funduszu odbudowy znajdują się środki na proces sprawiedliwej transformacji na obszarach pogórniczych. Podnoszono, że to jest szansa na odbudowę polskiego potencjału gospodarczego i energetycznego.

Są też środki na wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska i klimatu oraz finansowanie procesu modernizacji. Pan minister Szczepański w wypowiedzi na posiedzeniu Rady stwierdził: Dla Polski nie jest problemem warunkowość, dla Polski problemem nie jest praworządność. To co jest problemem dla Polski? Problemem dla Polski jest pewność prawna.

Rząd dysponuje informacją, że pozostałe 25 krajów członkowskich jest za przyjęciem wieloletnich ram. One nie mają problemu z pewnością prawną, tylko Polska i Węgry mają problem z pewnością prawną. Więc przełammy to, wysoki rządzie. Wysoka Izbo! W imieniu wnioskodawców tej uchwały chciałbym zaapelować: więcej wiary, panie premierze, więcej wiary, wysoki rządzie, nie gaście ducha w Polakach, nie mówcie, że 25 pozostałych państw członkowskich chce oszukać Polskę, chce podstępnie odebrać nam suwerenność czy narazić na szwank pomyślny rozwój ekonomiczny i gospodarczy Polski, polskich przedsiębiorców, rolników, bo tak nie jest, bo przecież zasada pomocniczości czy subsydiarności, chrześcijańska zasada stoi u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Elementem tej pomocniczości jest również jeden z najwyższych, jak powiedział pan premier, wynegocjowanych budżetów, łącznie z funduszem odbudowy, czego rządowi gratulujemy i oczekujemy, że się z tego nie wycofa, nie zrejteruje. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Otwieram dyskusję. Pierwsza - pani poseł Joanna Borowiak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec poselskich projektów uchwał zawartych w drukach nr 749, 753, 754 oraz 755. Jasne stanowisko w kwestii negocjacji budżetowych usłyszeliśmy wczoraj w Sejmie z ust premiera Mateusza Morawieckiego. Chcemy uchwalenia budżetu Unii Europejskiej w imię interesu Polski, a także pozostałych krajów członkowskich. Nie akceptujemy przy tym żadnych uznaniowych mechanizmów opartych na motywowanych politycznie kryteriach. Ich przyjęcie będzie prowadzić w konsekwencji do stosowania podwójnych standardów i nierównego traktowania państw Unii Europejskiej. Jak to jest, Wysoki Sejmie? Podobno opozycja jest za równością, ale gdy idzie o równe traktowanie państw Unii Europejskiej, próbuje zobowiązać własny rząd do zupełnie odmiennych działań. Unia, do której w 2004 r. wstępowała Polska, to unia wspierania pokoju i wartości - przypomnijmy, wartości chrześcijańskich - unia równości, także wobec prawa, unia zwiększania spójności gospodarczej i społecznej, unia solidarności między państwami członkowskimi, nie unia, w której jedni chcą uzyskać prymat nad drugimi. Przytoczę słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, które padły tutaj wczoraj: Rok 2020 to trudny czas i wyjście z niego będzie możliwe, jeśli będziemy solidarni i jeśli będziemy prowadzili politykę w interesie narodu polskiego. Tak, dziś interes naszego narodu wymaga tego, byśmy podjęli wspólne działania i nie pozwolili na wprowadzenie tylnymi drzwiami mechanizmów, które są szkodliwe dla Polski i przy okazji są szkodliwe dla całej Unii Europejskiej. Dlatego należałoby oczekiwać dziś od opozycji parlamentarnej wspólnego stanowiska popierającego działania polskiego rządu w imię obrony praworządności, równości i solidarności, w imię dobrze pojętego interesu własnej ojczyzny i jej suwerenności. Premier Mateusz Morawicki mówił jasno: Mówimy głośne „tak” dla Unii Europejskiej, ale głośne „nie” dla tych, którzy w nierówny sposób traktują Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. Praworządność jest dziś stosowana w Unii Europejskiej jako straszak w sposób odwrotny do wartości tego sformułowania. Dziś nie tylko Polska widzi zagrożenie w próbie stosowania mechanizmu naruszającego art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Przypomnę, że nie pozwala on na dyskryminacyjne działania wobec żadnego państwa członkowskiego ze strony instytucji unijnych i innych państw członkowskich. Widzą to Węgry, widzi to i mówi o tym głośno premier Słowenii. Jego słowa: Jeśli dojdzie do tego, że większość będzie decydowała o tym, co jest, a co nie jest zgodne z praworządnością, to będzie to koniec Unii Europejskiej. Premier Słowenii postuluje, aby wrócić do porozumienia z lipcowego szczytu Unii Europejskiej i, uwaga, nie forsować obecnego rozporządzenia. Opozycjo, wsłuchaj się w te odważne głosy. I jeszcze jeden cytat do opozycji, tak na smaczek: Nie byłoby dobrze, gdyby mieszać dwa porządki. Pieniądze, które w budżecie przeznaczamy na różne kwestie, nie powinny podlegać kryteriom czysto politycznym. Jak państwo posłowie myślą, czyje to są słowa?

Tacy jesteście światowi i europejscy, to przestańcie się bać. Czego się boicie? Dania, Szwecja, Holandia zagroziły wetem. Nie. Po prostu dopasowano budżet. Ale zaraz, te słowa też powinniście pamiętać, bo to za czasu waszych rządów wypowiedział je europoseł Janusz Lewandowski, w 2010 r. A więc odwagi, opozycjo. Polska potrzebuje dzisiaj waszej odwagi, nie tchórzostwa. Pani Marszałek! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości składam poprawkę do poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej, druk nr 755. o przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, bez odsyłania do komisji poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej, druk nr 755, a także wnoszę o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy, druk nr 749, o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej, druk nr 754. Ja tylko wnioski o odrzucenie przyjmę od pani. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Sławomir Nitras, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Panowie Ministrowie reprezentujący rząd! To jest niezmiernie ważna debata. Żałuję, że w czasie tej debaty nie ma tutaj ani pana prezesa Kaczyńskiego, ani pana premiera Morawieckiego, kolejność nieprzypadkowa. To jest ważna debata, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest debata o stanie negocjacji, o poziomie negocjacji, o tym, jaki chcemy osiągnąć skutek w negocjacjach budżetowych, również w negocjacjach nad funduszem odbudowy, odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-owym, gospodarki, która jest naprawdę w trudnej sytuacji. Ale to nie jest tylko debata o tym, to jest również debata o tym, czy Polska będzie w Unii Europejskiej za kilka lat, dlatego że takie procesy przechodzą w sposób dynamiczny.

Stawiam z tej mównicy twardą tezę: moim zdaniem zdolność pana Kaczyńskiego do realnej oceny polskiej pozycji w Unii Europejskiej, polskiej obecności w Unii Europejskiej jest zachwiana. Ona nie jest prawdziwa. Pan Kaczyńskie w stanie, w którym się znajduje, nie jest w stanie uczciwie ocenić, w jakiej jesteśmy sytuacji politycznej i jakie są skutki decyzji politycznej. którą wymusza na panu Morawieckim.

Przedstawiał się jako polski patriota, przedstawiał się jako człowiek, który broni polskiego interesu. Jakie były skutki i jakie były przyczyny takiego jego stanowiska, dzisiaj wiemy. To był człowiek, który był niesamodzielnym, to był człowiek, który działał na polecenie sił z Moskwy, i to był człowiek, który nie był polskim patriotą, tylko to był człowiek, który działał wbrew interesowi państwa. To był człowiek który. Oni mieli marne kadry.

To nie jest przypadek. Dzisiaj na poziomie ministra i wiceministrów w MSZ nie ma nikogo, kto przeszedł przez szkołę dyplomatyczną, jakiekolwiek szczeble kariery czy byłby na jakiejkolwiek placówce. Ci ludzie dzisiaj decydują o polskim stanowisku w Unii Europejskiej. To jest o panach, panowie, o panu Szynkowskim, o panu Kowalskim. Polacy! O polskiej polityce zagranicznej decydują dzisiaj tacy ludzie, którzy - powtórzę za panem Czaputowiczem - nie przeszli żadnej szkoły dyplomatycznej, nie przeszli żadnych szczebli dyplomatycznych, ba, nigdy nie byli na żadnej placówce. Ci ludzie dzisiaj decydują o tym, czy Polska weźmie udział w podziale funduszy na odbudowę gospodarki europejskiej po kryzysie. Decydują o tym, czy będziemy mieli europejskie pieniądze z budżetu, w imieniu samorządów i wszystkich innych, i ci ludzie dzisiaj decydują o tym, czy za kilka lat Polska będzie w Unii. Apeluję do wszystkich parlamentarzystów: będziecie rozliczani z tego głosowania dzisiaj, będziecie rozliczani.

Dyskutujmy na argumenty. Możemy się nie zgadzać, różnimy się tutaj w opiniach, natomiast jeżeli pan mówi o wicepremierze, wygłasza uwagi dotyczące jest stanu rozpoznania rzeczywistości, jego stanu zdrowia, wykracza to poza normalną debatę parlamentarną. Pan może mnie krytykować, ministra Kowalskiego. Byliśmy razem w jednym Stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści i wtedy się dobrze współpracowało, to było 20 lat temu. Od tego czasu pan postanowił zostać politycznym happenerem, a ja jestem wiceministrem polskiego rządu reprezentującym Polskę w polityce zagranicznej.

Dlaczego?

Problem polega na tym, że suwerenem w Polsce jest naród, obywatele, a nie pan Kaczyński. To jest problem. lub braku zdrowia psychicznego pana Kaczyńskiego, i nie mówiłem na ten temat ani słowa. Mówiłem o tym, że wczorajsze wystąpienie pana Kaczyńskiego tutaj, w Sejmie, wyraźnie pokazuje, że nie jest on w stanie realnie ocenić sytuacji, w jakiej znajduje się politycznie Polska w Unii Europejskiej, i podtrzymuję to twierdzenie. On nie jest w stanie racjonalnie tej sytuacji ocenić, i boję się, że pod wpływem człowieka, który [[Dzwonek]] nie jest w stanie racjonalnie tego ocenić. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Agnieszkę Pomaską. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Myślałam, że ta debata o suwerenności będzie przede wszystkim o tym, iż suwerenność przez PiS jest rozumiana jako obrona interesów kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości. Ale okazuje się, że jest jeszcze cel nadrzędny, czyli ochrona interesu pana Jarosława Kaczyńskiego. ale chodzi o obronę interesów koleżanek i kolegów pana Kaczyńskiego, a na końcu pana Kaczyńskiego. Po drugie, chodzi o zapewnienie ministrowi Ziobrze komfortowych warunków dalszego niszczenia niezależnego sądownictwa w Polsce.

Po czwarte, chodzi o możliwość niepublikowania wyroków, jeśli są niewygodne dla władzy, chodzi o niepublikowanie ustaw, jeśli nie podobają się panu prezesowi Kaczyńskiemu lub komuś innemu z Prawa i Sprawiedliwości. I chodzi o rzecz chyba najważniejszą. Mówimy o pieniądzach europejskich, ale dobrze wiemy, że chodzi o obronę interesów w spółkach Skarbu Państwa i wydawania publicznych pieniędzy nie tak, jak powinny być wydawane. Dzisiaj mówimy o pieniądzach unijnych. Chodzi o to, żeby unijne pieniądze mogły być przez Prawo i Sprawiedliwość wydawane tak, jak są wydawane dzisiaj publiczne pieniądze, polskie pieniądze, polskich podatników, ze spółek Skarbu Państwa. Takich przykładów na nadużywanie władzy, na nadmierne wykorzystywanie środków publicznych w Polsce mamy dzisiaj mnóstwo. Przypomnę kwestię respiratorów - bezużytecznych. Przypomnę kwestię testów - wadliwych testów za miliony złotych. Czy ktoś dzisiaj poniósł konsekwencje? Nie. Przypomnę chociażby kwestię słynnego portalu Puszcza.tv, założonego przez szefów „Gazety Polskiej” - 7 mln zł na portal, o którym pewnie niewielu z państwa słyszało - tylko po to żeby ktoś z koleżanek i kolegów pana prezesa Kaczyńskiego (Dzwonek) mógł zarobić. Czy ktoś za to został rozliczony? Nie. Nie będzie. Panie ministrze, niech pan wyjdzie i powie, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o ochronę interesów pana prezesa Kaczyńskiego i wszystkich pana kolegów. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szejna, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie chcę powiedzieć, że dosyć żałosna jest sytuacja, w której jeden człowiek, mam na myśli pana Zbigniewa Ziobrę, będzie wetował budżet. To Zbigniew Ziobro, bełkocząc coś o zniewoleniu, o utracie suwerenności, zmusił tych dwóch ludzi do tego, aby ustami ambasadora na posiedzeniu COREPER wyrazić wstępne weto wobec budżetu Unii Europejskiej, a więc wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy. Mógłbym dzisiaj dokonać bardzo konkretnej, bardzo głębokiej analizy - na to jest za mało czasu - co spotka Polskę i Polaków po tej waszej nie tylko karkołomnej, ale drastycznej decyzji. Ale chcę powiedzieć o jednej liczbie: 637. To jest liczba zgonów w Polsce dziś. Proszę się skupić. To 637, a może więcej, osób. A za chwilę mówimy też o przedsiębiorcach, o pielęgniarkach, o lekarzach, mówimy o samorządach, mówimy o wszystkich tych, którzy czekają właśnie na fundusz odbudowy gospodarczej skonstruowany w Unii Europejskiej. To jest 750 mld euro. Czekają na to wszyscy w Polsce. A wy dzisiaj odbieracie im nadzieję, tym wszystkim, o których wspomniałem, i przyczyniacie się do zwiększenia śmiertelności, do pogłębienia beznadziei, do unicestwienia oczekiwania na obronę miejsc pracy wielu Polek i Polaków. Bo wy unicestwiacie fundusz odbudowy gospodarczej. Może pani poseł się skupi, pan minister też i zrozumiecie jedną rzecz. Jesteście bezproduktywni, ponieważ wetując budżet, nie wpłyniecie na rozporządzenie Parlamentu i Rady dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. To są dwie różne rzeczy. Nawet jeżeli zawetujecie, Unia Europejska przyjmie to rozporządzenie, panie ministrze, przyjmie to rozporządzenie większością kwalifikowaną. Wy nie możecie postawić weta. Niech pan się nie śmieje. Chyba pan nie studiował prawa europejskiego. Przyjmie. Po pierwsze, nie dostaniemy funduszy związanych z wieloletnią perspektywą finansową. Po drugie, fundusz odbudowy gospodarczej odpadnie. A po trzecie, nawet jeżeli będzie prowizorium budżetowe, to będzie właśnie podlegać przepisom tego rozporządzenia.

Ale to uderzy we mnie i w innych Polaków. W opozycję, ale też w waszych wyborców. To chcę wam dzisiaj powiedzieć i to jest bardzo, bardzo ważne. Ponosicie ogromną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia Polek, przyszłe pokolenia Polaków. Za to was rozliczymy bez wątpienia. Za to was rozliczmy już wkrótce. Ale ja pani nie grożę, pani poseł. Ja pani przemawiam do rozumu.

Bardzo się cieszę, że w tej kwestii opozycja mówi jednym głosem. Chcę wam powiedzieć, że jest to jeden z bardzo ważnych momentów, w przypadku których Polki i Polacy będą się wokół opozycji jednoczyć przeciwko wam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan minister mówił o planie zagłodzenia Polski w imię politycznych interesów przez polityka. Chciałbym ujawnić tożsamość tego polityka, który ma dokładnie taki plan. Jest to minister Zbigniew Ziobro. To minister Zbigniew Ziobro w imię swoich politycznych interesów polegających na tym, że chce obsadzić polski wymiar sprawiedliwości swoimi kolegami, chce zagłodzić Polskę.

To są środki, które mają służyć odbiciu się polskiej gospodarki po kryzysie. I te środki nie znikną, bo Unia Europejska nie zrezygnuje z planu odbudowy przez jakąś niezbyt rozsądną szarżę Polski i Węgier. Oni się zorganizują, oni ten plan odbudowy zorganizują. Dlaczego osłabiacie Polskę i wzmacniacie Niemcy? Dlaczego, mówiąc dużo o suwerenności, dużo mówiąc o sile Polski, robicie coś dokładnie odwrotnego? Premier Morawiecki bardzo ładnie mówił wczoraj o tym, że te słabsze państwa Unii Europejskiej powinny się organizować przeciwko hegemonii tych najsilniejszych, powołując się m.in. na państwa południa Europy, które mają podobny interes. To dlaczego nie mamy sojuszu z państwami południa Europy? Dlaczego one za nami nie stoją? Może dlatego, że kiedy Polska miała okazję wykazać się solidarnością wobec krajów południa Europy, chociażby w przypadku kryzysu uchodźczego, to tej solidarności im odmówiła. Więc może mniej gadania, a więcej konkretów, bo wychodzi odwrotnie. Mówicie o sojuszu słabych, a macie słaby sojusz z Węgrami. Mówicie o silnej Polsce, a osłabiacie Polskę, pozbawiając ją niezbędnych środków do tego, żeby rosła w siłę. Polska nie będzie silna albo słaba tym czy innym rozporządzeniem Unii Europejskiej. Będzie silna swoją gospodarką, będzie silna swoją edukacją, będzie silna swoją służbą zdrowia, będzie silna swoimi relacjami z partnerami w Unii Europejskiej. Wy to wszystko niszczycie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Po pierwsze, czym powinna być polityka, szczególnie w takich ważnych momentach? Polityka powinna być roztropnym dbaniem o dobro wspólne. I miarą tej roztropności jest właśnie uczynienie wszystkiego, żeby Polska była prawdziwie suwerennym, bezpiecznym i demokratycznym państwem. Będzie bardziej suwerenna, jak będzie coraz bogatsza, gospodarczo rozwinięta, jak jej obywatele będą żyli w dostatku. Żeby to uczynić, trzeba szukać pieniędzy. Część pieniędzy wypracowujemy my, płacimy podatki, rozwijamy się, ale od kilkunastu jesteśmy we wspólnocie państw, które dzielą się swoimi pieniędzmi, składają się na wspólny budżet. Stoimy na straży, żeby Polska nie straciła ani jednego euro. Jeżeli władza zeszła z drogi roztropności, roztropnego dbania o dobro wspólne, to rolą świadomej opozycji, rolą konstruktywnej opozycji jest wzywać, po pierwsze, do opamiętania, a także obiecać, po drugie, że po przejęciu władzy przywrócimy każde zmarnowane przez was euro. Weto jest silną bronią, tylko jego siła jest większa nie w momencie użycia, tylko do momentu użycia. To tak jak z przyciskiem atomowym.

Nie robicie tego niestety na użytek dyplomacji, która powinna być środkiem do osiągania celów za granicą czy we wspólnocie Unii Europejskiej. Wy dyplomację sprowadziliście do rozstrzygania swoich sporów wewnątrz obozu władzy. Jest walka w obozie władzy. Ona jest od dawna. Jest walka pomiędzy radykałami i premierem Morawieckim.

Do czego doszło? W lipcu doszło do postawienia kroku w stronę federalizacji Unii Europejskiej. O tym w ogóle nie dyskutujecie. O wspólnym zadłużaniu, o wyemitowaniu obligacji.

Ohydnym jest używanie sformułowania: tzw. praworządność.

Bo nie ma suwerenności bez praworządności. Jeżeli nie macie sobie nic do zarzucenia, a często tak powtarzacie, że jesteście najlepsi, to czemu się tej praworządności boicie? To ją przestrzegacie czy jej nie przestrzegacie? To nie mają być regulacje dotyczące tylko i wyłącznie dwóch państw w Unii Europejskiej, tylko wszystkich. Jak orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dla was korzystne, to Trybunał Sprawiedliwości jest fajny i praworządność jest dobra. Jak się zdarzą niekorzystne, to się obrażacie nie na błędy - i nie wyciągacie wniosków z błędów popełnionych przez was - tylko obrażacie się na sprawiedliwość, na praworządność. Szukacie takich rozwiązań, które komplikują pozyskanie tych środków. Po pierwsze, przestrzegać praworządności - nie będzie żadnego problemu z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Po drugie, za błędy wasze, rządu PiS nie mogą zapłacić Polacy i będziemy tego strażnikiem, będziemy tego pilnować, żeby żadne euro nie zostało zmarnowane. Po trzecie, jeżeli rząd nie chce wydatkować tych środków, to one powinny trafić bezpośrednio do samorządów. I o to będziemy zabiegać w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, żeby skrócić ten transfer, żeby było bezpośrednio i jak najbliżej obywateli - to też jest, jak myślę, pomysł na ciekawe pójście do przodu, na ciekawą debatę dotyczącą w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie dopuścimy i zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić do utraty środków, które są dzisiaj Polsce bardzo potrzebne. Wyjście z kryzysu, rozbudowa naszej gospodarki i uzyskanie większej, a nie mniejszej przez to suwerenności. To jest spór o charakterze kierunków rozwojowych Polski. My chcemy Polskę silną, dostatnią i bezpieczną. Wy chcecie Polskę sprowadzoną na manowce, Polskę siedzącą w oślej ławce Unii Europejskiej i będącą czarną owcą - to już jest połączenie wszystkiego, co jest niestety esencją waszych rządów. Opamiętajcie się, wróćcie na drogę rozsądnego dbania o dobro wspólne, traktujcie dyplomację na użytek zewnętrzny, a nie na rzecz walki wewnętrznej. Niech premier Morawiecki dopełni tego, do czego się zobowiązał na szczycie. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! W „300Polityka” czytam, cytat: Proszę pamiętać, że corocznie bogate kraje Unii Europejskiej wyprowadzają z Polski dużo, dużo większe pieniądze niż te, które uzyskujemy z dopłat unijnych. Dopłaty unijne są mechanizmem rekompensującym. Kto to mówi? Minister sprawiedliwości w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Pytanie: Po co pan premier Morawiecki zachęca inwestorów z zewnątrz, żeby inwestowali w Polsce? Po co pan premier Morawiecki uznaje za sukces kolejne inwestycje w przemysł motoryzacyjny? Przecież to są elementy, które mają wzmacniać naszą gospodarkę. Jeżeli ktoś wyprowadza pieniądze, a władza publiczna o tym wie, to powinniśmy poszukać metod prawnych rozwiązania tej sytuacji. Natomiast nie łączmy tego, nie łączmy tego. Bo kontekst tej wypowiedzi jest jaki? Z uznaniem przyjmuje się fakt zablokowania przez przedstawicieli Polski dalszych prac nad budżetem, nad pakietem rozwiązań budżetowych. Myślę, że jeżeli chcemy być poważnym krajem, to powinniśmy użyć swojej dyplomacji i swoich umiejętności oraz swoich przewag po to, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. To jest sukces polskiego rządu, [[Dzwonek]] który my z ochotą przyjmiemy w tej Izbie. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Kiedy widzę działania rządu PiS w tej sprawie, to mam przed oczami scenkę sprzed 3 lat, kiedy wesoła gromadka pod przewodnictwem pana Jarosława Kaczyńskiego witała panią premier Szydło wracającą z Brukseli po łomocie, jaki dostała wtedy Polska w sprawie przewodniczącego Rady Europejskiej. Ano dlatego, że państwo z PiS-u kilka lat wcześniej, łącznie z panem prezydentem śp. Lechem Kaczyńskim, zgodzili się na traktat lizboński, zgodzili się na takie mechanizmy, które Polskę pozbawiły realnego wpływu na bieg zdarzeń. W lipcu Rada Europejska przyjęła zapisy o tym, że łączy się interesy finansowe Unii, że są chronione w związku z praworządnością. Koniec, kropka. Na to zgodził się premier Morawiecki w lipcu. Teraz obecne weto, o którym rozmawiamy, dotyczy tylko unijnego budżetu na lata 2021–2027. Wiele państw w historii Unii Europejskiej czy jeszcze wcześniej wspólnot europejskich wielokroć stosowało instrument weta jako normalny instrument nacisku politycznego, jako element negocjacji politycznych w Unii Europejskiej. Natomiast podkreślmy, Mateusz Morawiecki już oddał polską suwerenność w lipcu tego roku, zgadzając się na powiązanie mechanizmu praworządności z finansami. Taka jest prawda. Procedura nigdy nie była testowana. Ostatecznie wszystko będzie zależało od tego, czy będzie wola polityczna ukarania danego kraju, czy uda się dla takiej decyzji uzyskać większość. Tydzień temu, w czwartek, Komisja Europejska przedstawiła pierwszą strategię w historii Unii Europejskiej dotyczącą promocji LGBT, m.in. wzajemne uznawanie rodzicielstwa w sytuacjach transgranicznych, co legalizuje, co ma legalizować w całej Unii homoadopcje. Zaproponowana strategia jest niezgodna z traktatami, niezgodna z prawem państw członkowskich, w przyszłości stanie się podstawą do zastosowania mechanizmu praworządności - ku temu zmierzamy. Każdy, kto dzisiaj z PSL-u, z Lewicy, z Platformy jest za tym, żeby Polska powiązanie tego lipcowego mechanizmu szanowała, honorowała i nie przeciwstawiała się temu, jest za tym, żeby Unia m.in. egzekwowała od nas uznanie homoadopcji. Tak, państwo z Koalicji Obywatelskiej i z PSL-u, za tym dzisiaj jesteście. Rozszerzenie prawa rodzicielskiego na pary homoseksualne w krajach UE, w których takie prawo nie obowiązuje, wynikało z orędzia pani Ursuli von der Leyen o stanie Unii z 16 września 2020 r. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju Unii, to jesteś rodzicem w innym kraju - to jest tekst pani Ursuli von der Leyen.

Praworządność jest tylko pretekstem, chodzi o polityczny szantaż, prymat politycznych i arbitralnych decyzji nad merytoryczną oceną decyzji politycznych danego państwa członkowskiego. Będzie to forma presji politycznej na Polskę i Węgry. Dzisiaj, kiedy stoimy tutaj, w tym miejscu, musimy sobie jasno powiedzieć, że Polska powinna realnie przejść do ofensywy. W 2010 r., kiedy Viktor Orbán został premierem Węgier, wezwał Polskę do tego, żeby była liderem Europy Środkowej. W 2015 r., kiedy zmienił się rząd w Polsce, ponownie Orbán mówił takie słowa. Pojechał do Waszyngtonu i powiedział: przy tobie, najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. Otóż dzisiaj decyduje się to, czy Polska, współpracując m.in. z powstającym właśnie w Azji największym obszarem wolności gospodarczej, współpracy gospodarczej na świecie, będzie pomostem między Wschodem i Zachodem, czy będzie prowadziła politykę wielowektorową, czy będzie realnie odgrywała rolę na scenie politycznej i gospodarczej świata, wykorzystując swoje położenie, czy utrwalimy swoje peryferyjne położenie w strukturach euroatlantyckich wobec Zachodu, który nas kolonizuje politycznie, gospodarczo i kulturowo. To jest walka o realną suwerenność. Trzeba powiedzieć jasno: rząd Morawieckiego tę suwerenność oddał niestety już w lipcu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Nie da się spokojnie słuchać tych opowieści z mchu i paproci, które tu słyszymy z obu stron. Ale prawda jest po prostu taka, że tak działa Unia, tak działa gilotyna, w którą wsadziliśmy głowę dawno temu. Unia jest skonstruowana właśnie w ten sposób, żebyśmy nie mieli tam nic do gadania, żebyśmy byli prowincją, której zarządców, gubernatorów lokalnych przekupuje się paciorkami. Tak działa gilotyna. Liczenie na to, że jakoś to będzie, że jakoś tę głowę uchylimy, że może przejdzie bokiem, jest po prostu skrajnie naiwne. I tak, oczywiście że Unia Europejska stosuje podwójne standardy, ale skarżenie się teraz na to przez polityków PiS to jest jakaś polityczna piaskownica. Nie wiedzieliście, że tak będzie, jak podpisywaliście traktat z Lizbony? Przecież my to mówiliśmy już w 2003 r., w 2009 r., powtarzamy cały czas, że kupujemy sobie bilet w jedną stronę - do statusu kolonii brukselskiej. Przez cały ten swój krótki pobyt w Parlamencie Europejskim starałem się, żeby jedna prosta rzecz do wszystkich tutaj dotarła: Unia Europejska będzie się stawała jednym państwem, z jednym rządem, z jedną walutą, jedną armią i pod przewodnią rolą Niemiec. Nikt nas nie będzie pytał o to, czy się na to zgadzamy, czy nie. Albo się zapisujemy do tego projektu na takich zasadach, albo nie. Nikt nas nie będzie pytał. W tej sprawie lewa połowa sali jest nawet w pewnym sensie uczciwsza, bo oni nie próbują udawać, że walczą o niepodległość. W czasie exposé pytałem pana premiera, jak sobie wyobraża reformowanie Unii od środka, bo według mojej wiedzy to Unia nas zreformuje. Jak idzie reformowanie Unii od środka?

Ale PiS, grupa PiS-u głosowała przeciwko temu. To wy nie przekonaliście swoich kolegów i to wy nie uratowaliście Polski przed tym. Tak że nie ma żadnych złudzeń, Unia Europejska tak będzie działała. Jeśli trwamy w Unii na takich zasadach, na jakich się do niej zapisaliśmy, to nie jesteśmy w stanie nic więcej wynegocjować i poprawić swojej pozycji negocjacyjnej, zwłaszcza z taką klasą polityczną, która wzywa na pomoc obce siły na użytek walk wewnętrznych. Powiązanie praworządności z funduszami jest w oczywisty sposób mechanizmem, który służy do destabilizacji sytuacji w Polsce w realiach, kiedy oni chcą zmienić władzę.

Bardzo proszę, w trybie sprostowania pan poseł Dariusz Rosati. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Pan poseł Sośnierz był łaskaw mnie wywołać do głosu, więc chciałbym wyjaśnić nieporozumienie wynikające z tego, że rzeczywiście był dość krótko w Parlamencie Europejskim i do końca nie wie, jak przebiegają procedury.

Natomiast rząd PiS przegrał sprawę w Radzie, nie w Parlamencie. W Parlamencie zawsze większość była za tymi dyskryminacyjnymi rozwiązaniami. Chciałbym więc sprostować, że pozycja rządu polskiego osłabła tak dalece, że w Radzie rząd PiS nie był w stanie zgromadzić odpowiedniego sojuszu i odpowiedniej koalicji, żeby nie dopuścić do przyjęcia tych przepisów. Przechodzimy do pytań.

Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Suwerenność was bardzo uwiera, suwerenność polska was bardzo uwiera i dlatego zgłaszacie uchwały, które w istocie popierają nie stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej, ale stanowisko niemieckie. Szkoda, że krzykacze z Platformy Obywatelskiej wczoraj nie słyszeli znakomitego przemówienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział jasno - i takie było przesłanie - że polska suwerenność nie może być i nigdy nie będzie przedmiotem handlu. Gdybyście rządzili, tobyście przehandlowali polską suwerenność nie tylko za miliardy euro, których i tak byśmy nie otrzymali, ale też za złudne stanowiska. Dzisiaj, szanowni państwo, jest moment historyczny. Jeżeli rzeczywiście chcecie wspierać polski rząd i Rzeczpospolitą Polską w negocjacjach, poprzyjcie stanowisko zgłoszone przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Za panem premierem Mateuszem Morawieckim stoi 235 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią jasno: Suwerenność nie jest na sprzedaż. Chciałbym, żeby posłowie Platformy Obywatelskiej w końcu zaczęli myśleć po polsku, nie wypełniali rozkazów Berlina, Manfreda Webera i nie zgłaszali uchwał, które w istocie są poparciem Berlina. Dziękuję, panie pośle. Kolejne pytanie zada pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. Ale mam wielką prośbę do szanownych państwa. Wysłuchajmy się nawzajem. Bardzo proszę, pani marszałek. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Świat wokół nas jest niebezpieczny. W takim momencie bardzo dużo mówi się takich górnolotnych słów jak „patriotyzm” A czy patriotą jest ktoś, kto chce pozbawić Polskę funduszy? Czy patriotą jest ktoś, kto chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej? Czy patriotą jest ten, kto pozbawia nas praworządności, a co więcej, chce, żebyśmy byli osłabieni i nie mieli sojuszników? W tym czasie bardzo ważne jest podjęcie decyzji, czym naprawdę jest patriotyzm i co jest ważne dla naszego kraju. Nikt, kto mówi, że ważny jest interes jego ugrupowania, i stawia go nad interesem państwa, nie może o sobie mówić jako o patriocie. Mam wrażenie, że jeżeli nie przyjmiemy wspólnie, jako cały parlament, uchwały przeciwko wetu - chodzi o to, żebyśmy współpracowali z Unią, żebyśmy byli poważnym partnerem - to pokażemy, że nie jesteśmy nic warci, bo nie zależy nam na bezpieczeństwie naszego kraju. Chciałam jeszcze powiedzieć, że dla Europy Polska to nie tylko PiS. To także inni obywatele, którzy myślą o wartościach demokratycznych, o bezpieczeństwie, o współpracy. Dlatego to bardzo ważne, abyśmy dzisiaj wspólnie podjęli jedną uchwałę wspierającą uczestnictwo Polski w Unii, [[Dzwonek]] uczestnictwo w całym tym procesie. Kolejne pytanie zada pani poseł Beata Maciejewska, klub Lewica. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Jak to jest, że panu nie jest wstyd być takim słabym szefem rządu? Jak to jest, że pan się nadaje wyłącznie na prezesa banku, prezesa banku o nazwie PiS, w którym swoje akcje i interesy ulokowali politycy PiS-u, nieudolni ministrowie i przekrętacze?

Nie ma pan kręgosłupa. Pozwala pan na to, żeby harcownicy i fanatycy z Solidarnej Polski rozgrywali interes naszego kraju. Wyprowadza pan Polskę z Unii. Ma pan na to zgodę ludzi? Ze strachu przed Ziobrą i jego ludźmi wetuje pan budżet, który ma pozwolić odbić się od dna ludziom, którzy w odróżnieniu od pana i pańskich kolegów siedzących dzisiaj w tych ławach, zasiadających w spółkach Skarbu Państwa, siedzących na różnego rodzaju posadach niczego nie stracili. Dla Kaczyńskiego, dla Morawieckiego, dla Ziobry to są tylko słowa. Przez to, że zawetujecie budżet, szczególnie fundusz odbudowy gospodarczej, po pandemii możemy stracić 30% środków budżetowych wynegocjowanych przez pana w lipcu. Proszę kończyć. Pańskie motto, panie premierze Morawiecki, można określić krótko: po mnie choćby potop. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Posłowie! Panowie Ministrowie! Otóż zawsze w historii Polski, tej najnowszej i tej odleglejszej, bardzo źle kończyliśmy, kiedy partykularne interesy określonych grup, polityków zaczynały dominować nad racją stanu, nad interesem ogółu. Dzisiaj, drodzy państwo parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, przed nami też taki moment.

Spycha was na manowce, ale przez to ciągnie za sobą interes Polski. Być może sondaże, drodzy państwo, będą sprzyjać przez krótki czas.

Przestrzegamy przed tym. Myślę, że rozsądek u was też powinien wziąć górę, bo w interesie Polski leży dzisiaj to, [[Dzwonek]] aby korzystać z obecności w Unii Europejskiej, a nie to, żeby z niej wychodzić.

Ja nie wierzę, że państwo nie są w stanie zrozumieć, że takim właśnie rozgrywaniem konfliktu z Unią Europejską, takim przyklaskiwaniem szantażowi ze strony Unii Europejskiej pogarszacie sytuację negocjacyjną Polski, zmieniacie naszą i tak beznadziejną sytuację na jeszcze gorszą. Ale to jest zarzut do obu stron, bo zachowujecie się państwo wszyscy, jak byście szli do. Bo z drugiej strony też mieliśmy próby wpisywania do konstytucji i teraz mamy pomysł jakichś wiernopoddańczych laudacji na wstępie. Zachowujecie się jak człowiek, który idzie do szefa po podwyżkę i na dzień dobry mu mówi: Szefie, ja bez pana firmy to sobie nie dam rady, ja poza pana firmą nie dam sobie rady, ja zdechnę pod płotem, ja muszę tu pracować, poza tym jestem do niczego, tylko Białoruś, nędza i głód. A teraz będziemy twardo negocjować moją podwyżkę. Tak się zachowujecie. Musicie mieć z tyłu głowy możliwość twardego negocjowania również wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli chcecie się tam liczyć w ogóle w jakikolwiek sposób. I tak sytuacja jest beznadziejna, a wiernopoddańczymi laudacjami tylko ją jeszcze bardziej pogarszacie. Co chcecie w ten sposób osiągnąć?

rządzić się u siebie swobodnie? Pamięta pan, jak było? Nie powtórzyli wam tego głosowania, gdy zgrupowali tysiące waszych poprawek, żeby to przepchnąć przed końcem kadencji. Pamięta pan, jak było? I zrobią tak samo, żadnych złudzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W uchwale, którą dzisiaj prezentował pan minister Szymon Szynkowski vel Sęk, napisano, że zasada państwa prawnego sformułowana jest w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Ja jestem bardzo dumna, że we wczorajszym wystąpieniu pan premier Mateusz Morawiecki wypowiedział słowa, które właśnie zacytuję: Zrobimy wszystko, żeby przywrócić pewność prawa. A o tej pewności prawa w tych dwóch artykułach - jeszcze raz powtarzam, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Traktat o Unii Europejskiej - mamy wszystko jasno napisane. I o tę pewność prawa będzie walczył pan premier Mateusz Morawiecki, bo, cytuję dalej: Jesteśmy za silną, zasobną Europą i za silną Polską w silnej Europie. Bardzo serdecznie dziękuję za taką postawę i mam nadzieję, że Polska nie będzie w tej walce osamotniona. Chciałabym zapytać pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka, które państwa rozważają przyłączenie się do obrony europejskich wartości określonych w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską traktatach, bo wiemy, że to nie tylko Polska i Węgry. Bardzo proszę, pan poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że wszyscy pamiętamy taki film - a może książkę - „Kariera Nikodema Dyzmy” Tam jest taka scena, jak główny bohater powołany na zarządcę majątku w Koborowie mówi: Byle się jeszcze utrzymać, byle się jeszcze utrzymać, może miesiąc, może dwa, i liczy tak pieniądze. Wczorajsze wystąpienie pana Morawieckiego było właśnie takie: byleby się jeszcze utrzymać, może miesiąc, może dwa. Panie prezesie Kaczyński, proszę mnie nie odwoływać, ja zrobię wszystko, co chce pan minister Ziobro. W imię interesów pana Kaczyńskiego, w imię czy z racji waszych problemów koalicyjnych zabieracie, okradacie Polaków de facto z pieniędzy europejskich. Ta debata, która się dzisiaj toczyła, to nie jest debata tak naprawdę o praworządności, to jest debata o bezkarności. Wy chcecie sobie jeszcze na kilka miesięcy kupić bezkarność, ponieważ testu praworządnego... takiego testu praworządności nie przeszlibyście w żadnej procedurze, nawet jakbyście sami tę procedurę pisali. To, co widzimy na naszych ulicach, gazowanie i bicie pałkami kobiet, kordony policji, przekręty przy pandemii to jest przecież wasza codzienność, to jest wasza praworządność. Wy walczycie tylko i wyłącznie o waszą bezkarność. Naprawdę wiem, że was to boli, ale w imię jakiejś elementarnej przyzwoitości nie sprzedawajcie interesu Polski [[Dzwonek]] tylko dlatego, że jeszcze 2 czy 3 miesiące chcecie się utrzymać. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica.

Rozumiem, jeszcze dyskutujecie. Pan minister tutaj powiedział, że za panem premierem stoi 235 posłanek i posłów z PiS-u, a ja bym chciał, żeby stało 80% Polek i Polaków, bo tyle Polek i tylu Polaków popiera nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej. W związku z tym powinniście przede wszystkim [[Oklaski]] słuchać głosu Polaków, a nie siebie samych - siebie, by w imię swoich interesów podejmować decyzje w tej sprawie. Macie prawo oczywiście do weta, tak jak każdy kraj w Unii Europejskiej. Mówicie o tym, że kraje z tego korzystały. Tak, tylko proszę zobaczyć, z jakich powodów korzystały. Rzeczywiście walczyły o swoje interesy, a wy o co walczycie? O to, żeby nie było zapisów o tym, żeby była praworządność w Polsce. No, kompletne szaleństwo. Kompletne szaleństwo. Zwracam uwagę na to, że taką postawą powodujecie, że przynajmniej 25 innych krajów będzie, mówiąc krótko, przeciwko nam.

Druga rzecz.

Wysoka Izbo! Przez ostatnie 5 lat słyszeliśmy ze strony rządzących, że są praworządni, sprawiedliwi - mają z resztą w nazwie prawo i sprawiedliwość - że nigdy nie naruszają żadnych przepisów ani konstytucyjnych, ani krajowych, ani europejskich. Wczoraj z trybuny sejmowej nie kto inny, jak premier Kaczyński oznajmia: jeśli w Polsce będzie praworządność, będziecie siedzieć. W związku z tym wczoraj pan premier Kaczyński przyznał, że przez 5 lat w Polsce nie mieliśmy praworządności.

Chcę wam powiedzieć: nie bójcie się Ziobry.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Problemem opozycji jest dość poważny deficyt myślenia propolskiego. To po pierwsze. To, co mówicie, pokazuje, że macie bardzo nikłą wiedzę na temat procesów integracyjnych, jakie zachodzą w ramach wspólnot europejskich i Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu, od wielu lat Komisja Europejska w swoich działaniach prowadzi politykę podwójnych standardów. Jedne państwa karze, a drugie ewentualnie głaszcze.

Mam pytanie do pana posła sprawozdawcy.

Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo!

Panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Robert Kwiatkowski, Lewica. Bardzo dziękuję. Chciałem zaproponować trochę wbrew nastrojom panującym na sali taki eksperyment myślowy, który polega w skrócie na tym, że poważnie potraktujemy te pomysły, które rząd Prawa i Sprawiedliwości zgłasza, tzn. wymachiwanie szabelką i ogłaszanie możliwości zgłoszenia weta, co w znaczący sposób ograniczyłoby możliwości rozwoju Polski. Ta strona ław sejmowych, opozycja uważa to, mówiąc w skrócie, za szaleństwo, ale państwo najwyraźniej idziecie tą drogą. Dokąd chcecie nas zaprowadzić? Innymi słowy: Jaki jest plan B? I tu - wniosek do przedstawiciela rządu o pisemną informację na temat tego, jak rząd planuje cykl inwestycyjny, jakie punkty z krajowego planu odbudowy chce wyeliminować w sytuacji, w której będzie chciał bądź musiał zawetować wieloletnie plany finansowe, w której krajowy plan odbudowy zostanie zlikwidowany, bo drodzy państwo, Wysoka Izbo, to nie jest tak, że debata na temat środków europejskich odbywa się tylko tutaj. Pracują nad tym już od lata tego roku, tzn. od momentu, w którym premier Morawiecki ogłosił sukces, samorządy. W samym województwie kujawsko-pomorskim wstępne wnioski opiewały na ponad 400 mld zł i to nie jest żaden wyjątek. Poinformujcie naród, poinformujcie Polaków, że wszystkie te plany, wszystkie te wnioski inwestycyjne trzeba wyrzucić do kosza.

Mam nadzieję, że zostałem właściwie zrozumiany. Zapraszam panią poseł Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Wszelkie działania prawne muszą być oparte o jasne, jednakowe dla wszystkich, precyzyjne, określone z góry przepisy prawa.

Pacta sunt servanda - to jest stara prawnicza zasada.

Więc ja mam do was, droga opozycjo, pytanie: Dlaczego nie chcecie stanąć w prawdzie i zadać sobie najważniejszego, oczywistego pytania? Nie ma się co uśmiechać, bo prawo powielaczowe doskonale znamy ze słusznie minionego ustroju.

Bardzo proszę, pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! To jest debata o przyszłości Polski, o naszych żywotnych interesach, o wartościach. W żywotnym interesie Polski jest bycie w Unii Europejskiej i zajmowanie tam jak najsilniejszej pozycji, a w interesie każdego obywatela, każdego z nas, także w waszym interesie, jest przestrzeganie praworządności, jest to, żeby prawo było przestrzegane, żeby wszyscy byli równi wobec prawa i żeby władza nie mogła wykorzystywać swojej przewagi nad obywatelem.

Wiecie, czym jest ta uchwała? To jest akt zdrady narodowej. I każda osoba, która zagłosuje za tym dokumentem, podpisuje się pod aktem zdrady narodowej. Wy w imię waszych brudnych interesów jesteście w stanie zniszczyć nasze interesy narodowe. Naszą przyszłość. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Z kolei rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje sprawiedliwą, dostatnią Polskę. Ta sprawiedliwa Polska to również zdrowy system sądownictwa. I tutaj reforma sądownictwa, która jest prowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego, wzoruje się bardzo często na rozwiązaniach, które były wdrożone w innych krajach Unii Europejskiej.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cóż takiego się stało - to jest pytanie do koalicji rządzącej - że u dumnych Hiszpanów zanikło poczucie suwerenności? Co takiego się stało, że dzielni Litwini wyrzekają się suwerenności i swojej niepodległości? Jak to się dzieje, że tyle krajów europejskich nagle na naszych oczach wyrzekło się patriotyzmu i swojej ojczyzny i idą wprost na dyktat niemiecki? Przecież tak naprawdę jedynym waszym sojusznikiem jest człowiek, który dokonał takich działań korupcyjnych na pieniądzach unijnych, że Unia powiedziała, że nie będzie finansowała budowania węgierskiej oligarchii. On ma za sobą już naprawdę ścianę. To jest wasz sojusznik. A wy w tej sprawie zachowujecie się, szanowni państwo, jak szuler, który złapany za rękę mówi: Polska, Polska, ponieważ ma wrażenie, że kradzież tych drobnych w ten sposób ujdzie uwadze. Otóż najgorszą zbrodnią, jaką możecie zrobić, jest ośmieszenie patriotyzmu polskiego, [[Oklaski]] ośmieszenie rangi Polski jako państwa, które po prostu rozumie swoją suwerenność. Jesteście w tej sprawie szulerami posługującymi się słowami: ojczyzna, Polska i suwerenność tylko po to, żeby tak naprawdę. ochronić swoje drobne interesy, [[Oklaski]] tak jak właśnie robi to Orbán, tylko Orbán nie ma wyjścia, a wy macie wyjście. Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szefowie rządów 27 krajów Unii Europejskiej w lipcu tego roku zgodzili się na powiązanie przyszłych wydatków z budżetu Unii Europejskiej z praworządnością, ale ten mechanizm miał nawiązywać do traktatowych zapisów o ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej, a więc miał na celu walkę z zagrożeniem przy wydawaniu środków europejskich. Chodzi tutaj o korupcję, niegospodarność czy defraudację. Dlatego pragnę zadać pytania. Czy prawdą jest, że jesteśmy tutaj wzorcowym państwem, że właśnie w naszym kraju dokładnie i w sposób bardzo precyzyjny i zgodnie z prawem realizujemy ten traktat? Czy prawdą jest, że dzisiaj w Holandii można. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w poniedziałek wniosek prokuratury i odmówił przekazania małżeństwa, które zabrało cierpiącego na autyzm syna z niderlandzkiej placówki i przyjechało z nim z Holandii do Polski. Para jest ścigana europejskim nakazem aresztowania. Postępowanie władz holenderskich należy ocenić jako skrajnie nieludzkie i barbarzyńskie.

I czy prawdą jest, że dzisiaj w Unii Europejskiej obowiązuje takie prawo? Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po tych słowach, które powiedziała przedmówczyni, czas jest jednak na chwilę prawdy. To nie Unia się zmieniła, to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii. Robicie to dla obrony własnych interesów, dla ulegania rokoszowi Zbigniewa Ziobry, dla utrzymania władzy, która wymyka wam się z rąk. Inaczej przecież nie da się wytłumaczyć tych lunatycznych działań, tych gróźb, weta dla unijnego budżetu i dla Funduszu Odbudowy, dla wsparcia, które pomoże wyjść z pandemii, które jest szansą na zrewolucjonizowanie polskiej gospodarki, na postawienie jej na nowe tory, na modernizację, na transformację energetyczną, na walkę o klimat. W imię własnych interesów chcecie pozbawić Polki i Polaków szansy na bezpieczne jutro. A przypomnę, że praworządność, do której zobowiązała się Polska, wynika wprost z zasad traktatu. Poszanowanie prawa, ochrona sądownicza, zakaz dyskryminacji. Na to zgodziliśmy się w referendum w 2003 r. i wstępując do Unii Europejskiej w 2004 r. Dlaczego kompromitujecie Polskę [[Dzwonek]] na arenie międzynarodowej, szkodzicie Polsce? Dlaczego chcecie wciągnąć w to także Sejm? Bardzo proszę, pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość.

mówił tak podłe rzeczy o Polsce. Jeżeli on dzisiaj mówi o polskim patriotyzmie, to proszę wybaczyć, proszę państwa, ale ja mam po prostu odruch wymiotny. To jest po prostu coś obrzydliwego. Kolejna sprawa, proszę państwa, to jest rzecz dotycząca wizerunku Polski w Unii Europejskiej. Przecież to są bzdury. Ale dlaczego mówicie, że to, co my w tej chwili robimy, to jest kwestia PiS-u? nam zaufało i nam powiedziało, że droga, którą idzie Prawo i Sprawiedliwość, jest drogą właściwą dla interesów Polski. I czy się wam podoba, czy nie, będziemy dbać o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Nie zakrzyczycie.

Kolejna sprawa. Jeden z posłów Lewicy tutaj mówił, że oto bawimy się Unią Europejską, tak jak zrobili to rządzący w Wielkiej Brytanii, doprowadzili do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie oni, proszę państwa. Zrobiła to społeczność Wielkiej Brytanii.

I my o taką Unię Europejską będziemy walczyć.

Wysoka Izbo! Za kilka godzin pan premier będzie próbował przekonać unijnych liderów do tego, że polskiej praworządności nic nie grozi. Mam w związku z tym pytanie: Czy w praworządnym kraju prześladuje się sędziów z powodów politycznych? Przecież zaledwie wczoraj odebrano immunitet sędziemu Igorowi Tulei. Zrobiła to bezprawnie działająca Izba Dyscyplinarna wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tuleya jest prześladowany politycznie, bo ujawnił niewygodne dla was fakty [[Oklaski]] dotyczące nielegalnego głosowania na sali kolumnowej. Już wobec tysiąca sędziów toczą się postępowania dyscyplinarne za to, że są niezależni od polityków obecnej władzy. I pan premier będzie mówił o praworządności? Przecież to są znamiona dyktatury. Państwo nie bronicie polskiej suwerenności, państwo bronicie Zbigniewa Ziobry i jego szaleńczej polityki niszczenia polskiej praworządności. I naprawdę zamierzacie robić to dalej? Naprawdę będziecie bronić dalej Ziobry i jego chorej polityki i poświęcicie na to 150 mld euro, na które czekają Polacy, Polki i polska gospodarka? Wysoka Izbo! Tylko wariat albo zdrajca może dzisiaj powiedzieć, że z uznaniem przyjmuje zablokowanie prac nad unijnym budżetem. Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak, proszę państwa, to bardzo dobra, bardzo potrzebna uchwała przypominająca, że Polska to - dużymi literami, proszę państwa - suwerenny kraj, przypominająca najważniejsze ważności, m.in. solidarność międzyludzką, o której tak często zapomina opozycja, a wręcz ordynarnie ją wypacza. O tę solidarność między państwami zabiegał i zabiega pan premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, dziękujemy wszyscy, że, myśląc o przyszłości Polski, myśli również o przyszłości Unii Europejskiej. Dlatego, panie ministrze, proszę o przedstawienie przykładów, może z tego roku, wyjątkowego roku pandemii, kiedy polski rząd pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego wykazał się solidarnością z innymi krajami Unii Europejskiej. Po co? A mianowicie po to, żeby Polska zobaczyła, opozycja usłyszała, że nie jesteśmy pariasami Europy, nie jesteśmy żebrakami Europy, jak chcecie nam wmówić. Bo to nie o interes ekonomiczny chodzi, ale o sprawy ideologiczne.

Prawdę powiedział pan Kierwiński, prawdę powiedział pan Kierwiński.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Większość sejmowa chce dzisiaj przegłosować uchwałę, która ma m.in. takie słowa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem przyjmuje fakt zablokowania przez przedstawicieli Polski dalszych prac nad pakietem rozwiązań budżetowych. Mamy w Polsce kryzys zdrowotny, kryzys gospodarczy, kryzys społeczny i kryzys finansów publicznych.

Wy nie jesteście wariatami, na pewno nie wszyscy. Jesteście wrogami Polski. Chcecie dalej bezkarnie niszczyć praworządność i wolne sądy, bo musicie mieć partyjne sądy, musicie mieć partyjne sądy po to, żeby broniły waszych złodziejskich interesów. Żeby broniły Banasiów, Szumowskich, Biereckich. Ale mam dla was złą wiadomość: pieniądze Polaków niestety mogą przepaść, ale mechanizm powiązania finansów z praworządnością i tak wejdzie w życie, [[Dzwonek]] bo Parlament Europejski przegłosował go już w 2019 r. i większość kwalifikowana jest, a Morawiecki się na to zgodził w lipcu. Bardzo proszę, pan poseł Daniel Milewski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Drodzy Państwo! Wy nawet macie trochę racji. Europa potrzebuje debaty o praworządności. Wy dzisiaj zaczęliście dzień posiedzenia od opowiadania o jakichś rzekomych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu polskiej Policji.

Rozmawiajmy o tym, co się dzieje we Francji i jak się tam traktuje sędziów. Rozmawiajmy o tym, jakie są skutki kryzysu emigracyjnego wywołanego przez Niemcy na dzisiejszą sytuację, na dzisiejsze bezpieczeństwo obywateli w Europie. Ale my dzisiaj mówimy o budżecie, o budżecie, który ma być wolny od nacisków politycznych. Polska i Węgry sprzeciwiają się mechanizmowi arbitralności, uznaniowości i mówimy to w sposób otwarty. Są też inne państwa, które mają coraz więcej wątpliwości co do propozycji przyznania Komisji Europejskiej pozatraktatowych uprawnień, bo w obecnej formie ta propozycja to jest mechanizm niepraworządnego paradoksu. Panie Ministrze! Proszę przybliżyć Wysokiej Izbie, w jaki sposób ten mechanizm uznaniowości, arbitralności, warunkowości w takiej formie narusza zarówno traktaty, jak i [[Dzwonek]] polski porządek konstytucyjny. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Jeszcze w lipcu pan premier mówił, że weto byłoby jak strzelenie sobie w łeb, teraz słyszymy: weto, weto, weto albo śmierć. No rzeczywiście brak weta, powiązanie z praworządnością byłoby jak śmierć dla polityki rządu, który praworządność ma za nic. Natomiast dla mnie to krzyczenie: weto, weto to jest tak jak: amnestia, amnestia w zakładzie karnym. Oczywiście weto chcecie po to, żeby móc kraść, żeby móc łamać prawo i żeby traktować Polskę jako wielkie sukno, z którego możecie wyrwać jak najwięcej. Bardzo często powołujecie się na Wielką Brytanię. Wielka Brytania rzeczywiście groziła wetem. Tak, że na końcu wyprowadzili ją z Unii Europejskiej. Zwykle wetem groziły te kraje, które były płatnikami netto, które musiały dopłacić do budżetu Unii Europejskiej. My dostajemy więcej, niż wpłacamy. 100 mld rocznie to jest to, co otrzymamy w najbliższej perspektywie razem z Funduszem Odbudowy. Co to oznacza? 100 mld to jest nasz cały budżet na zdrowie, 100 mld to są wasze dwa programy 500+, 100 mld to są pieniądze, które decydują o życiu Polaków, o życiu ekonomicznym, o życiu edukacyjnym, o kulturze, o zdrowiu. Tego chcecie pozbawić Polaków.

Wysoka Izbo! Ta debata jest debatą o przyszłości Polski, o tym, czy będziemy decydować o naszych sprawach tu, w Warszawie, w parlamencie. czy też będą za nas o tym decydować jacyś brukselscy urzędnicy, których nikt nie wybierał i którym nikt nie dawał do tego prawa. Od lat opozycja chce likwidacji polskiej suwerenności. Brzydząc się polską przeszłością, Tusk mówił o tym, że Polska to taka nienormalność.

Szanowni Państwo!

Jaruzelski nawet wzywał na pomoc rosyjskie wojska. Teraz w Polsce mamy ludzi, nawet tych samych co wtedy, twierdzących, że służba Unii Europejskiej jest równoznaczna ze służbą ojczyźnie. Otóż, szanowni państwo, siła Polski bierze się z ducha przywództwa narodowego i dzisiaj polski parlament może dać narzędzie naszemu przywództwu narodowemu do twardej walki o polskie interesy, a pokora i uległość służą tylko (Dzwonek) wzmacnianiu i utrwalaniu niewoli, do jakiej chcecie doprowadzić sprzedażą polskich interesów, proponując nam niby złotą klatkę. Ta nasza, o której mówimy. Dziękuję bardzo. Proszę o spokój na sali.

Szanowni Państwo! Pan przewodniczący Budka na początku swojego wystąpienia klubowego, w zasadzie chyba w pierwszym zdaniu powiedział o tym, że my nie wiemy, czym jest solidarność. Solidarność polega właśnie na tym, że mamy pewien wspólny mianownik, wspólny obszar działań. Na tym polega solidarność, że potrafimy coś ustalić razem. Ta uchwała dawała państwu taką szansę.

A mówicie, że nie rozumiemy, czym jest solidarność. W tym szczególnym roku 40-lecia „Solidarności”, szanowni państwo, pokazujemy tę solidarność w obliczu pandemii w praktyce. Szanowni państwo, w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności pomogliśmy Białorusi, pomogliśmy Ukrainie, pomogliśmy 14 innym państwom w ramach pomocy dwustronnej, wysyłając maseczki, płyn dezynfekcyjny, środki ochrony medycznej. Wysyłaliśmy misje medyczne do kilku krajów, m.in. do Włoch, Słowenii, Stanów Zjednoczonych. W ramach NATO-wskiego mechanizmu pomocy jesteśmy trzecim największym donatorem po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. My nie wiemy, co to jest solidarność? To jest polski gen solidarności z innymi w tym trudnym czasie. Tak, skończyłem prawo europejskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeśli pana to interesuje, to moja praca magisterska obroniona w 2006 r. była na temat procedur stanowienia prawa unijnego. Praca nowatorska, oparta - co panu pewnie się spodoba - na niemieckich źródłach, ponieważ wtedy w Polsce nie było tego typu prac. W międzyczasie był traktat lizboński, trochę się zmieniło, ale proszę się nie bać, aktualizuję wiedzę i wiem, jak tworzone jest prawo w Unii Europejskiej, i chętnie panu wyjaśnię szczegóły tworzenia tego prawa. Chciałbym wyrazić wdzięczność przewodniczącemu Grzybowi, że przeczytał treść uchwały, jako że ją cytował. Pan poseł Paszyk zapytał, czy będziemy reprezentować interes własny, czy interes Polski. Pani poseł Milczanowska pytała, które państwa stają z nami ramię w ramię w obronie wartości.

Pani poseł Paluch zapytała, czy Polacy powinni decydować o tym, jak wydajemy pieniądze, czy urzędnicy brukselscy.

Komisja Europejska nigdy tymi kwestiami się nie interesowała, panie pośle. Pani poseł Gasiuk-Pihowicz pyta, czy w praworządnym kraju prześladuje się sędziów. Nie ma chyba pani poseł. Odpowiadam: Nie, w praworządnym kraju nie prześladuje się sędziów, w Polsce nie prześladuje się sędziów.

Mówiąc w skrócie (Dzwonek), traktaty nie przewidują możliwości takiej kontroli, nie przeniosły kompetencji w tym zakresie na instytucje unijne, a te kompetencje, które nie zostały przeniesione na instytucje unijne, przysługują państwom członkowskim zgodnie z art. 5 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, tzw. zasadą przyznania. Odsyłam do tego artykułu.

Oczekiwałem większej liczby pytań, ale tylko niektórzy zdecydowali się na zadanie pytania w ramach pytań, niektórzy ograniczyli się po prostu do własnych wystąpień politycznych, nie zawsze kulturalnych. Straciliście szansę, żeby służyć Polsce - po raz kolejny. Żałuję. Dziękuję bardzo.

Gratuluję świetnego wykształcenia i znajomości prawa europejskiego, ale wydaje mi się, że albo pan używa swojej wiedzy w złym celu, albo nieuważnie czytał pan pewne książki i nieuważnie je teraz interpretuje. Po drugie, w trybie sprostowania. Pan nie odpowiedział właśnie na moje pytania. Otóż niech pan odpowie dzisiaj uczciwie wyborcom, tu i teraz, przed majestatem Sejmu, czy prawdą jest, że jeżeli zawetujecie budżet Unii Europejskiej, fundusz, zdewastujecie przyszłość Polek i Polaków, to i tak procedura praworządności zgodnie z rozporządzeniem będzie obowiązywać.

Gratuluję. W trybie sprostowania jeszcze pan Dariusz Rosati, a potem pan minister. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Chciałbym, żeby odpowiedział mi pan na proste pytanie w takim razie: Czy jak zawetujecie ten budżet, to Polska będzie miała pieniądze czy nie? Tylko niech mi pan to udowodni. A jeśli powiecie, że nie, nie będzie miała pieniędzy, to ja chcę panu powiedzieć, że to jest sytuacja, w której pozbawiacie Polskę pieniędzy i pozbawiacie Polskę praworządności, a jednocześnie zmuszacie Polskę do tego, żeby robiła to, czego nie chcecie. Czyli będzie podlegała mechanizmowi kontroli.

Ja wszystkich dobrze traktuję na tej sali. Teraz zapraszam pana ministra Michała Wójcika. Jako minister rządu ma prawo zabrać głos w dowolnym miejscu. Dziękuję, pani marszałek. Szanowni Państwo! Jeszcze nie zacząłem mówić, a państwo już krzyczycie. Z racji tej, że pełnię funkcję ministra konstytucyjnego, mam prawo odnieść się do pewnych rzeczy. Pani marszałek, ubolewam, że jako marszałek polskiego. Bardzo proszę o spokój na sali, proszę pozwolić mówić panu ministrowi. Jeżeli mogę, pani marszałek. Uważam panią za osobę z wielką klasą i nie wstydzę się tego powiedzieć, natomiast ubolewam, że pani nie reaguje na przejawy absolutnego chamstwa, którego mieliśmy okazję doświadczyć z tej mównicy. Nazywacie nas fanatykami, zdrajcami, nazywacie nas idiotami, głupkami. Nie, my jesteśmy wielkimi patriotami. My patrzymy wiele lat do przodu. Taka jest prawda. Nie macie prawa do tego, żeby używać takich słów wobec nas. Wy nawet się nie zastanawiacie, bo to była okazja, żeby prowadzić dobrą debatę, bo my rozmawiamy o przyszłości Polski. Nie jesteśmy tylko tu i teraz, my patrzymy na przyszłość. Czy was to nie boli, że jest próba przeforsowania mechanizmu, który ma dotyczyć praworządności, ale nie jest oparta na żadnym prawie traktatowym? Wam się to podoba, że tylnymi drzwiami wprowadza się mechanizm, który mówi o praworządności, a nie ma takiego przepisu. Nikt nigdy nie przyjął takiego przepisu. To nie jest tylko nasze zdanie, to jest zdanie służb prawnych Unii Europejskiej. Wam to nie przeszkadza. Dlaczego mówię, że jesteśmy patriotami? Dlatego że niezależnie od tego, kto będzie w przyszłości rządził w Polsce, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tylnymi drzwiami wprowadzić mechanizm, żeby urzędnicy brukselscy decydowali o tym, jak Polska ma być zorganizowana.

Pan Mark Rutte na początku procesu legislacyjnego chciał złożyć weto, on groził wetem, tak samo jak Francuzi grozili wetem. To jest coś, na co my się zgadzaliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej. My nie jesteśmy salonowcami brukselskimi, nas nie interesują ciepłe posadki, pieniądze. Nie, szanowni państwo, to wy jesteście, to wy jesteście salonowcami, taka jest prawda. To nawet wasz lider Donald Tusk mówił w 2018 r., że nie wolno łączyć (Gwar na sali, dzwonek) w tym mechanizmie praworządności ze środkami unijnymi. Co powiecie na to? Co pan powie, panie przewodniczący Budka, bo tak mocno wczoraj pan się wypowiadał pod adresem premiera? Mówił pan o zdrajcy, o zdrajcach, co pan powie o panu Tusku. Zamilkliście nagle, prawda? Pytacie się o Holandię, szanowni państwo, przez 5 lat zajmowałem się dziećmi, jeździłem po całej Europie. Proszę pani, wiedzą to ministrowie, moi odpowiednicy w innych krajach, co zrobiłem dla dzieci, nie tylko w Polsce.

Pary, małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które z dzieckiem autystycznym wyjechało z tej praworządnej Holandii i przyjechało do niepraworządnej Polski, szukając tutaj azylu, schronienia. Co zrobił sąd w Warszawie? Odmówił wydania tych ludzi w ramach europejskiego nakazu aresztowania. A wiecie, na jakiej podstawie? Nie fakultatywnej - obligatoryjnej, że się łamie prawa człowieka w tym kraju i że tym ludziom grozi niebezpieczeństwo, jeżeli wrócą do Holandii, i dlatego zachował się tak, jak przyzwoity człowiek - odmówiono wykonania ENA. Jedna z pań posłanek, pani Gasiuk-Pihowicz mówiła o panu Tulei i pokazywała, że z powodu pana Tulei, z powodu tego, co zrobiła izba dyscyplinarna, która nie jest podobno sądem, że to jest skandal, że to nie jest praworządność. A dlaczego?

Otóż chcę powiedzieć, że rozumiem, że praworządnym jest kraj, w którym sędziów wybierają politycy, bo tak jest w Niemczech, a nie w Polsce, i nie ma rady sądownictwa, czyli kogoś, kto stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Było milczenie, wymowne milczenie. Pamiętajcie o tym. Bardzo proszę o spokój na sali. Szanowni państwo, oczekujemy jeszcze na wystąpienia przedstawicieli wnioskodawców. Bardzo proszę o spokój, bo mamy jeszcze wiele punktów do zrobienia. Jeszcze wniosek formalny pan Krzysztof Paszyk. Wysoki Sejmie! Chciałabym złożyć wniosek formalny, prosić o przerwę i zaproszenie do Wysokiej Izby ministra do spraw Unii Europejskiej pana Konrada Szymańskiego, żeby wyjaśnił Wysokiej Izbie, szczególnie prawej stronie. Bardzo proszę o spokój na sali, koledzy. żeby wyjaśnił Wysokiej Izbie, panu ministrowi Wójcikowi i panu premierowi Morawieckiemu, którzy wprowadzili Wysoką Izbę w błąd, mówiąc, że jakieś przepisy wprowadza się tylnymi drzwiami. Chcę, żeby minister Szymański powiedział, że rozporządzenie o powiązaniu finansowania z praworządnością przyjęła Komisja Europejska w 2018 r., Parlament Europejski - w 2019 r., Rada Europejska zgodziła się na ten mechanizm w lipcu 2020 r., jednomyślnie z premierem Morawieckim, i teraz ten mechanizm ma być przyjęty większością kwalifikowaną (Dzwonek) przez Radę Unii Europejskiej i przegłosowany przez parlament. Jakie to są tylne drzwi? Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Nitras w trybie sprostowania. Tak, dlatego że wtargnął tutaj na mównicę jakiś pan, który mówi, że jest ministrem konstytucyjnym, chociaż nikt nie wie, czym się zajmuje - może pan powie, czym się pan zajmuje jako minister konstytucyjny - i zaczął nas obrażać. mówiąc o tym, że bronią praworządności. Ja panu powiem, na czym polega problem.

Pan był wiceministrem sprawiedliwości, kiedy do Polaków po kilka razy.

To co zrobiliście?

Niszczycie ludzi, a jednocześnie takich ludzi jak Kaczyński czynicie bezkarnymi.

Panie pośle, bardzo pana przepraszam, ale miałam upoważnienia dla pana ministra i pan minister zgodnie z prawem zabrał głos w tej debacie. Bardzo proszę, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. Szanowni Państwo! Pan minister Wójcik twierdzi, że tzw. Izba Dyscyplinarna może... nie może orzekać tylko i wyłącznie w kwestiach związanych ze zdjęciem immunitetu. Orzekł o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdjęcie immunitetu sędziemu Tulei jest bezprawnym działaniem, jest wywieraniem niewłaściwej presji na sędziów i robicie to masowo. Chcę powiedzieć jedną rzecz, bardzo jasno: Naprawdę standardami praworządności nie jest wywieranie presji na sędziów i niszczenie niezależności sądów. My dzisiaj walczymy o suwerenność Polski. Bardzo proszę o uspokojenie atmosfery na sali. Z wnioskiem formalnym pan poseł Krzysztof Paszyk. Potem zabiorą głos wnioskodawcy, a potem pan poseł w trybie sprostowania. Bardzo proszę o spokój na sali. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Składam w trybie art. 184 regulaminu Sejmu wniosek o przerwę, żeby panowie ministrowie Szynkowski vel Sęk i Wójcik ochłonęli i nie opowiadali więcej Wysokiej Izbie takich bzdur, jakie opowiadali.

Gdybyście system powoływania sędziów ukształtowali w Polsce w ostatnim czasie zgodnie z konstytucją i z ustawami, nikt by wam nie miał prawa na cokolwiek zwracać uwagę. Ale wy pogwałciliście konstytucję, pogwałciliście ustawy. A to się nazywa [[Dzwonek]] praworządność w całym cywilizowanym świecie, drodzy państwo.

Bardzo proszę o spokój na sali.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, czyli ci wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda prawdziwa solidarność, współpraca i elementarne zasady rządów prawa. I z drugiej strony szaleńcy, którzy dla własnego interesu politycznego podpalają Polskę. którzy są w stanie zaryzykować nawet utratę pieniędzy, które mogą pomóc Polsce w rozwoju, tylko po to, by nie zgodzić się na jakąkolwiek kontrolę. Odpowiadając na pytania posłów, które tutaj padały - otóż to jest strach przed rozliczeniem. Przecież to ci ludzie, którzy dzisiaj upominają się o zasadę praworządności, od 5 lat tę zasadę łamią. Przecież to ci ludzie, którzy w nazwie swojego ugrupowania już nie tylko mają „prawo i sprawiedliwość”, tak jak wy macie „polskie” w nazwie ugrupowania, ale zachowują się, zachowujecie się, jakbyście instrukcje dostawali z Moskwy. Jakbyście instrukcje dostawali pisane cyrylicą.

I dzisiaj sądzicie swoją metodą. Dzisiaj próbujecie wmówić, że nagle wszyscy są przeciwko Polsce. Wiecie, za co? Za „Solidarność”, za naszą historię, za to, że potrafiliśmy obalić komunizm. I zdecydowana większość Polaków jest proeuropejska. Mamy tego pecha, że rządzą nami współcześni bolszewicy, ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest integracja. ludzie, którzy ryzykują pieniądze rolników, pieniądze przedsiębiorców, pieniądze samorządowców, ryzykują rozwój Polski i bezpieczeństwo tylko dlatego, żeby umacniać swoją pozycję.

I on śmie pouczać premiera polskiego rządu, co ma robić? Tylko że gdybyście wy mieli odrobinę rozsądku - mówię do posłów Prawa i Sprawiedliwości - tobyście swojego premiera bronili, a nie wystawiali go na pożarcie człowiekowi, który później was wsadzi do więzień. Czy wy nie rozumiecie, że ta gra nie toczy się o to, jaki będzie budżet? To jest gra o to, kto będzie następcą Kaczyńskiego. Jesteście chorzy z nienawiści do wszystkich, którzy rozumieją, czym jest solidarność i współpraca. Niestety, szanowni państwo, ta debata was niczego nie nauczyła. Ta debata pokazuje, że wy jesteście w stanie poświęcić wszystko tylko po to, by utrzymać się bezkarnie przy władzy. Wy mówicie o solidarności, wy mówicie o praworządności? No tak, boicie się, bo wówczas instruktorzy narciarstwa nie mogliby interesów robić. Wy mówicie o praworządności, kiedy prokuratura tego pana, który tam siedzi, umarza postępowanie w sprawie wieszania na szubienicach?

Bo dzisiaj każdy prawdziwy patriota chce współpracy europejskiej. Dziś każdy prawdziwy patriota chce bezpiecznej Polski. Dziś każdy prawdziwy patriota chce.

Ugrają swoje i was zostawią. Wy chcecie tu i teraz. Wy chcecie po prostu tej władzy. Rozmontujecie Polskę i polski system bezpieczeństwa tylko po to, by utrzymać się przy władzy. Straciliście większość. Straciliście większość w momencie, kiedy podpaliliście Polskę.

Mówiłam, że po wnioskodawcach. Jeszcze pan poseł Grzyb przed panem wystąpi. Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców pana posła Andrzeja Grzyba.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Te emocje oczywiście są naturalne w debacie parlamentarnej, ale zdajemy sobie też z tego sprawę, że one przyniosły tutaj wiele niedobrych efektów. Właściwie wzmocniły ten podział, który obserwujemy od wielu lat w Wysokiej Izbie i również w polskiej polityce. Niemniej nie chcę podejrzewać nikogo o złe intencje. Przedstawiając ten projekt uchwały, który tutaj zaprezentowałem w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, jestem przeświadczony, że działamy w dobrej intencji. Działamy w dobrej intencji, stąd to nasze wezwanie do prezesa Rady Ministrów, który 21 lipca 2020 r. stwierdził, że sukcesem negocjacyjnym Polski - również premiera, który reprezentował Polskę na tym szczycie - jest osiągnięcie dobrego wyniku, jeżeli chodzi o wieloletni budżet i również plan odbudowy. Dlatego nie rozumiemy w chwili obecnej tego, jak wiele się zmieniło w stanowisku rządu i również w stanowisku premiera polskiego rządu, który chce postawić weto wobec tego budżetu.

Natomiast wydaje mi się, że ten konflikt wewnętrzny, który jest pomiędzy różnymi frakcjami Zjednoczonej Prawicy, prowadzi do akurat takiego stanowiska premiera. Jednak ufam, że to, co powiedział pan minister Szymański, m.in. w Radzie. Stwierdził: Polska nie ma problemu z praworządnością, Polska nie ma problemu z warunkowością budżetu, Polska ma tylko jedno pytanie, dotyczące właśnie tej pewności prawnej. Rozstrzygnijcie to państwo, bo wszystkie instrumenty ma premier, ma rząd, wszyscy jego współpracownicy, w duchu porozumienia pomiędzy tymi wszystkimi, którzy reprezentują Polskę w tej Izbie i reprezentują najlepsze intencje, ze swej strony, aby Polska i Polacy rozwijali się pomyślnie w Europie, która jest nam potrzebna. Nie jesteśmy na żadnym marginesie politycznych wydarzeń Europy. Jesteśmy w jej centrum. Nie podejmujmy decyzji, które w sposób bezprecedensowy niszczą tę naszą pozycję. To nie jest zrozumiałe, jeżeli w finale negocjacji nagle próbuje się wszystko zmienić. Również z naszej strony.

To są ważne fakty, których nie powinniśmy pomijać. W chwili obecnej serwujemy polskiej opinii publicznej poprzez tę debatę takie oto wrażenie, że tu dokonuje się jakaś sprzedaż polskich interesów. Wtedy też polski premier zgodził się na emisję obligacji, na sfinansowanie długu. To jest pytanie otwarte: Czy to nie jest tzw. moment hamiltonowski?

I to zrobiliście państwo jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, zawsze podkreślając ten element budowy Europy ojczyzn. My się z tym zgadzamy, ale jeżeli takie decyzje zostały podjęte, to szanujemy decyzję również polskiego premiera i polskiego rządu w tej sprawie. Dlatego oczekujemy tego, żeby dokończyć to z takim finałem, który będzie służył pomyślności Polski, a nie będzie pokazywał nas w nie najlepszym świetle. W trybie sprostowania pan poseł Kaleta. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie taka refleksja. Nigdy nie sądziłem, że powiem to z tej mównicy i w takich okolicznościach, ale można by było to powiedzieć: Grzegorzu Schetyna, wróć, bo to, co reprezentuje sobą człowiek. Sprostowanie. Państwo mówicie, że Prawo i Sprawiedliwość pod rządami premiera Mateusza Morawieckiego przynosi wstyd Europie. Puśćmy wodze wyobraźni.

Przyjeżdża do Polski delegacja, obojętnie z jakiego kraju. Negocjacje by poszły nie po waszej myśli. Co im powiecie?

Traktuję tę sprawę poważnie. Nie jest to fair i na przyszłość będę miała dużo mniejsze zaufanie do państwa posłów. Bardzo proszę, przedstawiciel wnioskodawców pan poseł Krzysztof Gawkowski. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Debata, którą kończymy, potwierdziła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wepchnąć Polskę do drugiej ligi europejskiej. Chcecie pozbawić Polskę 103 mld zł, które pomogłyby polskim firmom, rodzinom, zapewniłyby lepszą ochronę zdrowia i walkę z pandemią. Polska pod waszymi rządami miała wstawać z kolan. Zamiast tego będziecie na kolanach gonić europejską czołówkę i prosić, żeby was nie wypchnęła poza nawet drugą ligę. Lewica nie będzie bezczynnie patrzyła na to, co robicie, jak pozbawiacie Polki i Polaków środków na lepszą przyszłość. Mamy swoje rozwiązania i pracujemy nad ich wprowadzeniem w Unii Europejskiej od dawna. To was może zaskoczyć, ale was z Unii Europejskiej wypychają, a Lewicę, PSL i Platformę zapraszają. Wam nie można dać pieniędzy do ręki, bo nie jesteście dość odpowiedzialni, by nimi zarządzać. Wydajecie je na swoje limuzyny albo niedziałające respiratory. Dziwicie się, że Unia Europejska nie chce współpracować z rządem PiS-u, który świadomie i z pełną premedytacją łamie wszystkie reguły i standardy demokratycznego państwa. Pozbawiacie Polki i Polaków uczciwego procesu i zamiast rozmawiać, używacie politycznej pałki. Może zamiast pałki zacznijcie używać rozumu. Wtedy w Europie ktoś was będzie słuchał. Polki i Polacy nie mogą jednak tracić na waszym cynizmie i nieudolności, dlatego na forum Unii Europejskiej wnioskujemy o mechanizm, który zapewni wypłaty z Unii Europejskiej z pominięciem waszego rządu.

Ale nie wy będziecie o nich decydować. Nie wy będziecie po cichu, gdzieś w gabinetach decydować, że taka i taka gmina dostanie, bo jest tam burmistrz albo prezydent z PiS-u. O nie, nie, panowie i panie z Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy w opozycji wspierać swoje projekty, które służą Polsce. Boicie się tego, że was w Unii Europejskiej traktują jak persona non grata. Bo polska racja stanu to jest dla was polska racja Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość to dla was slogany, które mają zaprowadzić was do władzy. A dla nas prawo i sprawiedliwość to Polska odpowiedzialności, suwerenności, współpracy, zgody i wspólnego domu, jakim jest Unia Europejska.

Smuci was to, co mówimy z tej mównicy, dlatego że wiecie, że wasz czas się kończy. Czerwoną kartkę pokazuje wam Unia Europejska. Ale za to chcecie, żeby płacili Polacy. Premier z mównicy wczoraj mówił o suwerenności, ale to wy ją odbieracie Polakom. Premier wczoraj mówił o solidarności, ale to wy tej solidarności Polakom odmawiacie. Jesteście dzisiaj smutni, bo wiecie, że wasz lider wczoraj powiedział to, czego wy się wstydzicie. Jesteście pełni obaw i nie dlatego, że wam sondaże spadają, bo kiedyś spadną tak, że nawet nie wejdziecie do tego parlamentu. Problem polega na tym, że za cenę budżetu unijnego chcecie sobie kupić więcej czasu. Chcecie, żeby prokuratura was do więzienia nie wsadzała, a premier Kaczyński, żeby nas tu straszył. Przyszłość leży tam, gdzie Europa, nasz wspólny dom. W odpowiedzialności i we współpracy. W idei, która przez kilkadziesiąt lat pokazała, że od tego, że ktoś będzie machał kijem, pałką albo baseballem, nic w Europie się nie zbuduje. Lewica odpowiedzialnie wzywa was do tego, żebyśmy razem przyjęli budżet, który będzie służył Polkom i Polakom. Ale nawet jeżeli pójdziecie inną drogą, to ominiemy was, bo najważniejsza jest Polska. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Dziękuję, pani marszałek. Szanowni Panowie Posłowie! Chciałem jeszcze uzupełnić odpowiedzi. Pan poseł Szejna dopytywał, żebym konkretnie odpowiedział, więc odpowiadam. Zdawało mi się, że to było bardzo konkretne, ale odpowiadam jeszcze raz. Prace w sprawie rozporządzenia w sprawie warunkowości zostały zatrzymane, ponieważ do przyjęcia całego pakietu budżetowego potrzebna jest jednomyślność. Nie ma przyjętego rozporządzenia w tej chwili w sprawie warunkowości, więc ono nie będzie obowiązywało. Mówię to jasno. Chciałbym, żeby to jasno padło i żeby zakończyć dyskusję w tym względzie. Pan poseł Rosati pytał, czy weto sprawi, że Polska nie otrzyma pieniędzy. Istnieje roczne prowizorium budżetowe, tak że oczywiście nie jest tak, że Polska nie otrzyma pieniędzy z budżetu unijnego, jeżeli wieloletnie ramy finansowe nie zostaną przyjęte. Jeżeli pani poseł chce, żeby to dodatkowo wyjaśnić, oczywiście też to dodatkowo zrobię. W pierwszej rundzie zapomniałem na nie odpowiedzieć. Taką miarę można przyjąć niewykonanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: czy jakieś państwo realizuje prawo europejskie, czy nie, bo trzeba spróbować jakąś miarę przyjąć. Polska ma w tej chwili jeden niezrealizowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Dla przykładu, inne kraje, Niemy - trzy, Hiszpania - sześć, Grecja, jeśli dobrze pamiętam - 11, Włochy - 10. Na tej podstawie państwo oceńcie, czy Polska dobrze wykonuje prawo europejskie, czy też je źle wykonuje. Pan poseł Wieczorek też jeszcze pytał, czy przygotowujemy Polskę do wyjścia z Unii Europejskiej. Panie pośle, nie przygotowujemy Polski do wyjścia z Unii Europejskiej, ponieważ Polska nie planuje wyjścia z Unii Europejskiej, mówię to bardzo jasno, tak jak nie planowały wyjścia z Unii Europejskiej Francja, która odrzuciła traktat konstytucyjny dla Europy - poważniejszą rzecz niż wieloletnie ramy finansowe, bo to był traktat, czyli rzecz dotycząca całokształtu funkcjonowania Unii. Holandia - w referendum odrzucony traktat konstytucyjny dla Europy. Po drodze wiele innych państw, które mówiły o wecie - Dania, Holandia przy różnego rodzaju negocjacjach. To nie jest jakiś mechanizm, którego, nie wiem, od 50 lat, od czasu powstania Unii Europejskiej nikt nigdy nie zastosował, nie zagroził nim. Nie ma się też czego przesadnie obawiać. No i jeszcze pan przewodniczący Gawkowski mówił o jakichś mechanizmach, nad którymi pracuje Lewica, że będzie bajpasowany, że będzie obchodzony rząd, że bezpośrednio pieniądze będą trafiać do samorządów. Panie przewodniczący, wiem, że teraz mieliśmy czas pandemii, wszyscy dużo siedzieliśmy w domach, rzeczywistość wirtualna była nam bliska.

I nie w rzeczywistości prawnej. W rzeczywistości prawnej, traktatowej nie ma miejsca dla takich rozwiązań. Naprawdę to jest rzecz niebywała, żeby opowiadać takie głodne kawałki chyba tylko dla tych, którzy nie mają kompletnie żadnego pojęcia o prawie europejskim, bo ci, którzy już chociaż trochę mają pojęcie, to już widzą, że coś tu nie gra, że miałaby być taka konstrukcja wprowadzona demokratyczna, wedle której pan poseł Gawkowski decyduje, jak będą wydawane pieniądze unijne, a rząd polski nie decyduje o tym, jak będą wydawane pieniądze unijne. Poseł opozycji o tym decyduje, a większość parlamentarna o tym nie decyduje. To każdemu rozsądnie myślącemu człowiekowi wydaje się trochę dziwne i wirtualne, jak powiedziałem. Szanowni Państwo! Myślałem, że będą jakieś pytania, bo przecież złożyliście państwo projekt uchwały, że pan będzie odpowiadał. Ale pan jest zupełnie czym innym zainteresowany, pan nie jest zainteresowany własnym projektem uchwały, pan nie jest zainteresowany traktatami, podstawami prawnymi, pan jest zainteresowany tym, żeby wyjąć pałkę propagandową na tej mównicy i w tę stronę tą pałką wygrażać. To jest postawa, która lidera opozycji na pewno nie powinna charakteryzować, ale pan ma to wszystko gdzieś, pan rozmawia przez telefon, więc nie ma co z panem dyskutować. Na koniec powiem tylko tyle: z państwa wypowiedzi, z wypowiedzi opozycji przebrzmiewało przekonanie, że trzeba szybko przyjąć to porozumienie, bo będą pieniądze, bo będą pieniądze dla Polski.

że mu dopisuje warunki, że nie będzie mógł tych pieniędzy wziąć, jeżeli nie zrobi tego, jeżeli nie zrobi jeszcze czegoś, jeżeli nie spełni absurdalnych warunków. Tylko po to, żeby wziąć te pieniądze, podpisuje, co mu podłożą do podpisu. Chcemy ten kontrakt z Unią Europejską, unią wszystkich państw, wieloletnie ramy finansowe zrealizować, ale na sprawiedliwych, jasnych i uczciwych zasadach.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Bardzo chciałbym prowadzić normalną, odpowiedzialną debatę w tym parlamencie, ale to wy od 5 lat blokujecie taką możliwość. Dzisiaj przedstawiacie Wysokiej Izbie fałszywą diagnozę, fałszywe argumenty i fałszywą receptę. Polska nie jest sama w Unii Europejskiej, to wy jesteście sami jako ten rząd. Wy będziecie ciągle przegrywać. Dlaczego? Dlatego że wy nie potraficie zrozumieć, czym jest Europa. Europa opiera się na wartościach, które dla was są obce: solidarność, praworządność. Tego nigdy nie zrozumiecie, bo wy budujecie PRL bis. Tak jak kiedyś w PRL-u odrzucono plan Marshalla, tak dzisiaj tym wetem wy chcecie odrzucić plan ratunkowy dla Europy. Dlaczego? Bo chcecie być bezkarni.

Wysoka Izbo! Na podstawie regulaminu Sejmu składam wniosek formalny o przerwę, podczas której pani marszałek wyciągnie konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe wobec posłów, którzy złamali zarządzenie, które pani marszałek sama przygotowała i wydała. Wczoraj podczas posiedzenia pan poseł Jarosław Kaczyński występował bez maski. Abstrahując od tego, co mówił w tym haniebnym wystąpieniu, złamał zarządzenie pani marszałek.

Po pierwsze, przerwy nie ogłoszę, a po drugie, proszę państwa, przy okazji powiem, skoro pan o tym mówi, że wszystkie kluby złamały drugie moje ważne zarządzenie, ponieważ na drzwiach od prawa do lewa wisi lista posłów zgłoszonych do obecności na sali plenarnej. Powinno być 50 osób, a jest 139 osób. W związku z tym wszystkich państwa informuję, że jeśli w piątek, w następnym tygodniu będzie podobna sytuacja jak teraz, będziemy wyciągać konsekwencje regulaminowe. Proszę państwa, wytłumaczę. Wiecie co, państwo, naprawdę widzę, że wy nie macie poważnych spraw. Przechodzimy do głosowań nad projektem uchwały z druku nr 755. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały zawartego w druku nr 755, zechce nacisnąć przycisk.

Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały z druku nr 749. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały zawartego w druku nr 749, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały z druku nr 754. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały zawartego druku nr 754, zechce nacisnąć przycisk.

Proszę państwa, bardzo proszę o spokój i o powagę.

Spokojnie, spokojnie. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały z druku nr 753. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały zawartego w druku nr 753, zechce nacisnąć przycisk.

Przypominam, że wobec projektu uchwały z druku nr 755 zgłoszono wniosek o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania bez odsyłania do komisji. Kto z pań i panów posłów jest za propozycją niezwłocznego przystąpienia do drugiego czytania projektu uchwały zawartego w druku nr 755 bez odsyłania do komisji, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął, a tym samym wyraził zgodę na przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania. Przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały z druku nr 755. W związku z tym otwieram dyskusję. Proponuję, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji nad tym punktem. Jeszcze nie zdążyłam. Słyszę sprzeciw. W związku z tym, proszę państwa, 5 minut. Rozumiem, że sprzeciwu nie ma. Dziękuję bardzo. W takim razie otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, jak państwo wiedzą, pozytywnie ocenia projekt ustawy wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej, druk nr 755. Dziś w obliczu toczących się negocjacji budżetowych Polsce wyjątkowo potrzebny jest silny i wspólnie brzmiący głos polskiego parlamentu. Głos wspierający działania rządu służące obronie, podyktowane obroną przed tworzeniem mechanizmów naruszających unijne traktaty, zagrażających de facto praworządności w Unii Europejskiej. Takiego działania Polacy i my wszyscy dziś oczekiwalibyśmy od polityków i posłów opozycji parlamentarnej. Tego głosu polskiej opozycji niestety dziś zabrakło. Politycy opozycji nie skorzystali, pomimo szansy, jaką mieli, z możliwości zachowania się, jak trzeba, z możliwości ochrony polskiej racji stanu. Macie jeszcze państwo szansę na to, by jednogłośnie poprzeć projekt przygotowany przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Rok 2020 to trudny czas i wyjście z niego będzie możliwe, jeśli będziemy solidarni i jeśli będziemy prowadzili politykę w interesie narodu polskiego. Zapamiętajcie, dziś interes naszego narodu wymaga tego, byśmy podjęli wspólne działania i nie pozwolili na wprowadzanie tylnymi drzwiami mechanizmów, które są szkodliwe dla Polski i szkodliwe dla Unii Europejskiej. Macie szansę na to, aby poprzeć ten projekt, aby pokazać, że polski parlament wspiera polski rząd w negocjacjach budżetowych i w ochronie suwerenności. Pani Marszałek! Zgodnie z zapowiedzą wcześniejszą, działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszam poprawkę do projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej, druk nr 755. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Sławomir Nitras. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To jest naprawdę szalenie istotna debata. To jest ostatni moment, by wezwać państwa do opamiętania się, by wezwać większość parlamentarną do tego, żeby przemyślała swoją opinię, dlatego że wy nie decydujecie tylko o tym, że Polska nie weźmie udziału w pracach i zrezygnuje z pieniędzy, z wielkiego planu odbudowy Europy po COVID, wielkiego planu odbudowy Europy podobnego do planu Marshalla, wy powodujecie swoją polityką, jakimiś obsesjami dziwnymi, że Polska naprawdę może nie wziąć w tym programie udziału, a konsekwencją wieloletnią może być to, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej.

Chodzi o to, żeby paru typów spod ciemnej gwiazdy mogło rządzić Polską i żeby mogło ukarać każdego. kto stanie im na drodze.

Chodzi o to, żeby postawić tamę temu szaleństwu. Bo stan, w jakim wy podejmujecie tę najważniejszą decyzję w tym parlamencie, to jest stan, który tu wczoraj widzieliśmy. Jaki był stan ich świadomości? Czy można w takim stanie, w takim szaleństwie, podejmować najważniejsze decyzje o przyszłości narodu? Nie, nie można. To jest ostatni moment, kiedy możecie się zatrzymać. Prawda jest taka, że Polacy, których przez 50 lat trzymano poza Europą... komuniści 50 lat trzymali nas poza Europą, Polacy na taczkach ich wywieźli. I dokładnie tak samo: jeżeli podniesiecie rękę na obecność Polski w Unii Europejskiej, na taczkach was wywieziemy. Tak was historia oceni jak Cyrankiewicza. Bardzo proszę.

Panie i Panowie Posłowie! Poza śmiesznością tej uchwały trzeba jeszcze powiedzieć o kłamstwach wygłoszonych przez premiera Morawieckiego z tej mównicy, a tych kłamstw było całkiem sporo. Po pierwsze, pragnę zwrócić uwagę, że w lipcu pan premier Morawiecki zgodził się na wprowadzenie mechanizmu praworządności. Tylko pod szantażem pana ministra Ziobry zmienił zdanie. Taka jest prawda. Pan premier Morawiecki już zgodził się na to, co dzisiaj wetuje. Kłamstwo drugie. Pan premier Morawiecki mówi, że decyzje w Unii Europejskiej podejmują jacyś oligarchowie. Decyzje w Unii Europejskiej podejmuje 27 państw - członków Unii Europejskiej, szefów rządów. My należymy do tej wspólnoty i jesteśmy jednym z dwóch krajów. Na tym polega problem. Decyzje podejmują nie oligarchowie, tylko przedstawiciele społeczeństw poszczególnych krajów. Kłamstwo trzecie. Pan premier Morawiecki mówił, że Dania, Szwecja, Holandia zgłaszały skuteczne weto i dzięki temu dostały rabaty. Nie było żadnych rabatów, a weto było elementem negocjacji. Po porozumieniu nie było żadnego weta do tej pory. Pan premier przystąpił do porozumienia, a później mówi o wecie. Kłamstwo czwarte - prowizorium budżetowe. Co ono oznacza?

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! To jest kolejna odsłona naszej dyskusji. Nie będę zwracał się oczywiście w stronę opozycji, ponieważ jesteśmy zgodni. Szanowni państwo, odwołuję się do waszego serca, bo rozum niestety porzuciliście gdzieś tam po drodze i porzuciliście swoje przekonania, swoje doktoraty, panie ministrze, i przekonania dotyczące wykładni prawa europejskiego. Powiem jedną bardzo ważną rzecz, bardzo, bardzo ważną. Zrozumcie: wasz opór wobec praworządności w Polsce, w Europie nie znajduje nigdzie zrozumienia. Wasz opór wobec praworządności będzie realną szkodą dla polskich gospodarstw domowych, przedsiębiorców, rolników, lekarzy, pielęgniarek. Ale co jest najważniejsze? Czym jest praworządność? Otóż praworządność jest określona w wielu dokumentach Unii Europejskiej, traktatach, Karcie Praw Podstawowych UE. To jest państwo prawa, to jest dostęp do niezależnego, niezawisłego sądu, to jest poszanowanie praw mniejszości, to są wolne media, to jest wreszcie poszanowanie praw kobiet, których oczywiście nie uznajecie, bo pan premier Kaczyński uznał, iż kobiety w Polsce mają rodzić nieodwracalnie chore, uszkodzone płody czy martwe płody. Ale to nie jest najistotniejsze. Wasza strategia nie ma sensu, bo na końcu tej strategii jest porażka, porażka polegająca na tym, panie ministrze, że nie mówił pan prawdy w odpowiedzi na moje pytanie. Otóż i tak Rada przyjmie wspólnie z Parlamentem rozporządzenie, które uzależni wydatkowanie środków Unii Europejskiej od praworządności, od tego, czym żyjemy na co dzień. Przecież każdy z nas, każdy obywatel chce żyć w państwie, w którym ma prawo do sądu, ma prawo do opieki, ma prawo do bezpieczeństwa. Dlatego dziś tu i teraz chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz: nie szkodźcie Polsce, nie czyńcie szkody Polkom i Polakom. Nie ma w tym waszym działaniu niczego więcej niż strach przed Zbigniewem Ziobrą, który to Zbigniew Ziobro jest dzisiaj w Polsce premierem, ministrem spraw zagranicznych, ministrem sprawiedliwości i szefem Zjednoczonej Prawicy. Boicie się przyznać, że bez niego nie macie większości. Chcę dzisiaj tu, w tym miejscu, powiedzieć: nie pozwolimy na to, żebyście uczynili taką szkodę Polsce i Unii Europejskiej. Co więcej, apeluję do was: zastanówcie się i tę uchwałę, którą chcecie przyjąć, odrzućcie. Bo jak ją przyjmiecie, Polacy wam tego nie zapomną. Pan poseł Krzysztof Śmiszek, Lewica. Wysoka Izbo! Ta rozmowa dotyczy tego, w jakim kierunku pójdziemy: czy na wschód, czy na zachód. Ja wybieram zachód, Lewica wybiera zachód. Wybiera zjednoczenie, solidarność, rozmowę z partnerami, czasami trudną rozmowę, ale rozmowę opartą na argumentach. Rozmawiamy o kwestii międzypaństwowej współpracy w ramach najlepszego projektu, jaki wydarzył się w historii Europy, czyli Unii Europejskiej. Praworządność to prawa mniejszości, prawa kobiet, wolne sądy, wolne media, prawo do zgromadzeń, wolność ekspresji, wolność słowa. To wszystko zostało uregulowane nie tylko na bazie traktatowej, ale także np. w europejskiej konwencji praw człowieka, bo przecież na europejską konwencję praw człowieka niejednokrotnie powołuje się europejski trybunał sprawiedliwości. Standardy wyznaczone przez europejski trybunał sprawiedliwości czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to są te standardy, które powinny obowiązywać w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Wy wszystkie te zasady: prawa mniejszości, prawa kobiet, prawa człowieka, wolności obywatelskie rozumiecie na opak. My mówimy „tak”, wy mówicie „nie” Unia Europejska mówi: prawa kobiet, wy mówicie: zakaz praw kobiet.

Wasi eksperci, wasi europosłowie z Parlamentu Europejskiego mówią: a co tam, nie przyjmiemy budżetu, zawetujemy, będzie prowizorium. No to niech Polacy i Polki usłyszą: prowizorium to jest tylko dokończenie umów, które obowiązują teraz, zero nowych projektów, zero nowej wizji, zero nowych planów na odbudowę Polski. To jest tylko podstawowe finansowanie instytucji europejskiej, Komisji, Parlamentu itd., itd. Prowizorium staje się jakimś fetyszem, próbujecie zamydlić oczy Polkom i Polakom.

Bardzo proszę. Dziękuję, pani marszałek. Panowie Posłowie! Za sprawą niedawnego głosowania i większości PiS-owskiej debatujemy już tylko i wyłącznie nad jedną uchwałą, która zawiera zobowiązanie rządu polskiego do zgłoszenia weta i zablokowania pakietu finansowego, z którego dwa najważniejsze fundusze, czyli wieloletnie ramy finansowe oraz fundusz odbudowy, niosą ze sobą tak wiele euro dla Polski, tak wiele dla polskich funduszy i tak wiele środków finansowych na odbudowę naszej gospodarki po skutkach pandemii. Ta uchwała, która została nam do przedyskutowania, jest fatalna i bardzo szkodliwa. Ale jest jedno zdanie w tej uchwale, które zasługuje na uwagę. To zdanie mówi o tym, że polski Sejm wzywa rządy państw Unii Europejskiej, ażeby wróciły do uzgodnionych konkluzji Rady Europejskiej z lipca tego roku, kiedy szefowie państw, w tym Mateusz Morawiecki, zapisali następujące zobowiązanie związane z finansami unijnymi na najbliższą siedmiolatkę, tu cytuję: Interesy finansowe Unii są chronione zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w traktatach, w szczególności zgodnie z wartościami zapisanymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. A co ten traktat mówi? Ano ten traktat mówi, i warto to przypomnieć, że Unia opiera się na poszanowaniu godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym osób należących do mniejszości, i że wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji i tolerancji. Wiele z tych wartości w Polsce pod waszymi rządami zwyczajnie nie jest respektowanych. I to jest największy problem, z którym się dzisiaj mierzycie. Nie respektując tych wartości, chcecie brać pieniądze z Unii Europejskiej, a tych pieniędzy nie będzie. Ale, co gorsza, nie będzie ich nie tylko dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie ich dla Polaków. Mówienie o tym, że będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, jest oczywiście prawdą, tyle tylko, że pomija się jeden ważny aspekt: prowizorium budżetowe, jak każde rozwiązanie jednoroczne, nie może być użyte do finansowania inwestycji wieloletnich. A takie są również te, które w kampaniach wyborczych, w tym w kampanii parlamentarnej czy samorządowej, obiecywaliście. Jeden z moich kolegów klubowych ostatnio zapytał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy wreszcie powstaną te obiecane obwodnice na terenie województwa łódzkiego.

Kto wam podpowiada weto?

Wówczas też słyszeliśmy: Weto albo śmierć. Są w Parlamencie Europejskim, są w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wracamy do tekstu uchwały: Mając to na uwadze, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - proponujecie - z uznaniem przyjmuje fakt zablokowania przez przedstawicieli Polski dalszych prac nad pakietem rozwiązań budżetowych. To zdanie jest albo dowodem zdrady interesów Polaków, państwa polskiego i narodu polskiego, albo wyrazem politycznej głupoty. Zresztą tę polityczną głupotę potwierdza fakt, że za waszą propozycją weta stanęło zaledwie dwóch premierów, dwa państwa z budowanego od lat porozumienia, jakim jest Grupa Wyszehradzka, czy promowanego od niedawna tzw. porozumienia Trójmorza. A więc jedyne, co mi przychodzi teraz z tego miejsca wygłosić pod waszym apelem.

W ostatniej chwili przestał słuchać tych niedouczonych, tych szkodników i zatrzymał kurs Polski na ścianę. Tak i wy możecie przejść do historii Rzeczypospolitej Polskiej dobrym rozwiązaniem, wycofaniem się z weta, przyjęciem ram finansowych [[Dzwonek]] i poszanowaniem praworządności w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacja. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tutaj słyszymy, że z Unii mówią nam o praworządności. Praworządność to myśmy mieli czasami w Polsce, z Unii idzie nam leworządność, czyli przestrzeganie reguł opartych na wartościach lewicowych. Natomiast PiS nie chce mieć ani praworządności, ani leworządności, tylko po prostu robić, co chce, nie oglądając się na żadne przepisy, i to jest ta różnica. Co do weta to chciałem zauważyć, że po to jest prawo weta, żeby je czasami stosować, więc nie ma się co dziwić. Tylko oczywiście opozycja lewicowa, przekonując wszystkich, że premier Morawiecki to weto zastosuje, wzmacnia jego pozycję - bo będą się bali w tej Unii, że to zastosuje. Ale zdradzę tajemnicę państwową: on tego nie zastosuje, z całą pewnością. My nie wierzymy, że weto zostanie zastosowane. Dlaczego? Dlatego że przy okrągłym stole, właściwie w Magdalence, została zawarta taka umowa, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy, a niezależnie od tego wchodzimy do Unii i budujemy eurosocjalizm. Tylko po to, żeby udawać, że się opiera Unii, i dzięki temu dostać elektorat. Przypominam, co było już podnoszone wielokrotnie, że ta decyzja została podjęta już w lipcu. W tej chwili weto niczego już nie zmieni. To jest tylko i wyłącznie, powtarzam, po to, żeby elektorat PiS-u myślał, że tu jest ten dobry policjant, a tam jest ten zły policjant, z tej lewicy, i chce nas tutaj sprzedać. Natomiast jako ostatnią rzecz podniosę to, że wszyscy tu wierzą w te duże pieniądze z Unii. Jest taki mit na lewicy, że pieniądze dają nam szczęście i potęgę. To ja się pytam: Jeżeli dzisiaj - tutaj padł taki głos z tych ław - jesteśmy połączeni w czterech wielkich kryzysach, to dlaczego ten kryzys nie jest w Chinach, które nie dostały ani centa z Unii, tylko w kraju, który dostał ogromne pieniądze z Unii? A teraz mówię do strony, która nazywa się prawą, a prawą nie jest. Wierzycie, że Unia chce nam zrobić źle, że Niemcy chcą nam robić źle.

Parlament Europejski, Komisja Europejska czy jakiekolwiek inne organizacje międzynarodowe nie są od tego, żeby mówić nam, Polakom, co jest praworządne, a co nie jest praworządne. To jest nasza dewiza, to jest nasza suwerenność i powinniśmy o nią dbać.

Tak właśnie jest. Dziękuję, panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Szanowni Panowie Posłowie! Premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszego wystąpienia powiedział: to moment decyzji, czy nasz los ma być w naszych rękach. I to bardzo krótkie, esencjonalne, dobre ujęcie wagi tego momentu, w którym się znajdujemy. Opozycja miała szansę zrozumieć tę wagę i podjąć wyzwanie, miała szansę wzmocnić mandat negocjacyjny polskiego premiera, polskiego rządu do walki, do realizacji polskich interesów. Konieczna jest odpowiedź na to zasadnicze pytanie, a także na wynikające z niego dalsze pytanie:

Kiedy o to pytałem, państwo tutaj krzyczeliście: nie, premier Morawiecki nie zasługuje na nasze wsparcie. To jest ta odpowiedź. A więc jeżeli nie premier Morawiecki, to kto zasługuje na to wsparcie? Czy może pani wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley ze swoją tezą o zagłodzeniu niektórych krajów członkowskich?

Państwo wprost mówicie, że chcecie zrobić bajpas, żeby rząd nie miał udziału w wydawaniu środków, tylko żeby one bezpośrednio trafiały do samorządów.

To, że w ogóle pada taki pomysł, pokazuje, jakie są wasze intencje. I wy czasami też o tym mówicie. W szerokim katalogu tych wartości wymieniona jest również solidarność.

Ludzie pomagają sobie nawzajem, ale też Polacy na całym świecie organizują akcje pomocowe w 160 miejscach. Jest wiele akcji skierowanych do innych krajów, 14 krajów, którym pomogliśmy dwustronnie. Jesteśmy trzecim donatorem mechanizmu pomocowego NATO po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności nieśliśmy pomoc na Ukrainie, na Białorusi. Wiemy, czym jest solidarność, bo mamy w sobie polski gen solidarności, ale też my oczekujemy solidarności ze strony Unii Europejskiej, ze strony innych partnerów, innych państw i poszanowania różnorodności, a jednocześnie zachowania zasady jednomyślności, która powinna obowiązywać w kluczowych dziedzinach, bo z solidarności właśnie wynika zasada jednomyślności. A więc wymagany jest konsensus co do kluczowych spraw wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do tego się odwołujemy, to jest bardzo ważna zasada, chcemy, żeby polski gen solidarności stał się też europejskim genem solidarności. Może państwa zaskoczę tym, co powiem, bo państwo uważacie, że praworządność to jest taka idealna pałka propagandowa, jak to wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki, do okładania tych niepokornych. Tymczasem zasada praworządności jest bardzo ważna, przywiązujemy do niej dużą wagę. Zasada praworządności jest zapisana w art. 7 polskiej konstytucji. Proszę o wskazanie mi podstawy prawnej, na której został zaproponowany tzw. mechanizm warunkowości w traktatach europejskich. Bardzo proszę o wskazanie tej podstawy prawnej, gdzie ona jest. Nikt o niej dzisiaj nie powiedział. Bo ona nie istnieje. Taka podstawa prawna dla tego mechanizmu nie istnieje. Proszę o wskazanie mi w takim razie tej podstawy prawnej w polskiej konstytucji. Art. 90 polskiej konstytucji mówi bardzo jasno: możliwe jest przekazanie pewnych kompetencji kraju do organizacji międzynarodowej, ale tylko na podstawie umowy międzynarodowej, a więc na podstawie traktatu, nie na podstawie rozporządzenia. To jest niemożliwe, to jest rozwiązanie niezgodne z polską [[Dzwonek]] konstytucją. Praworządność to poszanowanie prawa, jeszcze raz podkreślam, działanie na podstawie i w granicach prawa. Te wszystkie elementy wskazuje ta propozycja uchwały. Ona wzmocni mandat negocjacyjny polskiego premiera. Ta moc mogła być jeszcze większa, ale państwo nie skorzystaliście z tej okazji. Pozostaje żałować. Proszę Wysoki Sejm o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie oraz poprawkę do projektu uchwały z druku nr 755, proponuję, aby Sejm przystąpił do głosowania nad tym projektem po doręczeniu paniom i panom posłom tekstu poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. 15 minut.

obrady. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. W trakcie drugiego czytania do projektu uchwały zgłoszono poprawkę oraz wniosek o odrzucenie w całości. Sejm podjął decyzję o nieodsyłaniu projektu uchwały do komisji i przystąpieniu do głosowania nad tym projektem po doręczeniu paniom i panom posłom tekstu propozycji. Zestawienie zostało paniom i panom posłom doręczone do druku nr 755. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu uchwały. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 755, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę wspierającą działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

Proszę pana posła Konrada Frysztaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Kto nie chce słuchać, proszę wyjść w kuluary, żeby pan poseł mógł zabrać głos. Proszę bardzo, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po wniosku o odrzucenie, tak jak referowałem wczoraj, ustawa ta wróciła na salę plenarną, jednak Wysoka Izba zdecydowała, że powrócimy do jej opracowywania. To tylko wskazuje, szanowni państwo, na fakt, że niestety ta ustawa nie jest dobrze przygotowana, a na pewno pod kątem procedowania nie było współpracy z rządem. Apelowaliśmy o to wielokrotnie, aby zabrać tę ustawę, poprawić ją, aby wrócić z ustawą, która będzie akceptowalna. Niestety takiego wniosku pan minister Dworczyk nie chciał przyjąć. Ustawa ta przede wszystkim podnosi wynagrodzenia podsekretarzy stanu, którzy mają zostać wcieleni do korpusu służby cywilnej. Podsekretarze, którzy znajdą się w korpusie służby cywilnej, będą zarabiać ponad 21 tys. zł. Jeśli chodzi o Radę Legislacyjną, o to też komisja pytała, dyskutowaliśmy dosyć długo na ten temat. Rada Legislacyjna - również zostaną im podniesione wynagrodzenia do sześciokrotności kwoty bazowej, czyli 12 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo członkowie Rady Legislacyjnej będą mogli za opinie i analizy pobierać dwukrotność kwoty bazowej, czyli dodatkowe 4 tys. zł. I również ważna zmiana, która znalazła się w tej ustawie, a o której powinniście państwo wiedzieć, to to, że zlikwidowano zapis o maksymalnej ilości członków Rady Legislacyjnej, która dotychczas wynosiła 20 osób. Bardzo wnikliwie podchodził do tej sprawy chyba przyszły szef komisji sportu pan poseł Szopiński, który bardzo wnikliwie pytał o sprawy dotyczące Narodowego Centrum Sportu. To, co do zasady, skopiowanie wszelkich obowiązków, które na dzień dzisiejszy wykonuje Ministerstwo Sportu, a które wręcz, trzeba powiedzieć jasno, zostaje zlikwidowane, a wszystkie kompetencje przejmie instytucja zewnętrzna, czyli Narodowe Centrum Sportu. Zwracaliśmy również uwagę Wysokiej Komisji na fakt, że cały czas istnieje w obiegu prawnym ustawa dotycząca Euro 2012 i nie wiem, czy państwo wiecie, ale Stadionem Narodowym zarządza spółka Euro 2012. Przecież można byłoby to zmienić, kto inny mógłby zarządzać, mogłaby zarządzać chociażby nowa instytucja, jaką będzie Narodowe Centrum Sportu. Ale warte podkreślenia jest, że większość rządowa w komisji nie uzyskała większości i poprawką opozycji Narodowe Centrum Sportu zostało skreślone z tej ustawy. To również, tak jak powiedziałem, warte podkreślenia.

Nie było rozstrzygnięte przyjęcie sprawozdania, nie było przyjęte odrzucenie tego sprawozdania, dlatego ogłoszona została przerwa do dziś rano. Trwały intensywne próby budzenia w nocy, które nie przynosiły rezultatu. Bardzo dziękuję.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, 1 minuta. Chwileczkę, panie pośle, jeszcze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Nigdzie nie aspiruję i nigdzie nie chcę z tego stanowiska, na którym jestem w ramach Sejmu, awansować. Natomiast interesuje mnie sam stopień tworzenia w Polsce prawa. I jeżeli mamy ustawę, która mówi o działach, a w ramach tej ustawy o godz. 3 nad ranem zmieniamy cały system związany z jednej strony z finansowaniem polskiego sportu, z drugiej strony z nadzorem nad polskimi związkami sportu, z trzecim elementem, z systemem kontroli, to musi to budzić mój niepokój. A jeżeli jeszcze zadaję pytanie, z jakimi polskimi związkami sportowymi było to konsultowane i otrzymuję odpowiedź, że z żadnymi, to pytam, dla kogo w Polsce tworzone jest prawo. Dziękuję bardzo. I teraz pan poseł Piotr Kaleta, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Nie chciałbym wchodzić w polemikę z panem posłem sprawozdawcą i z panem posłem z Lewicy. Wprawdzie sprawa była też trochę zgoła inna, niewątpliwie posiedzenie komisji doprowadziło do swego rodzaju klinczu, co wywołało naszą dzisiejszą debatę, ponieważ komisja nie była zgodna co do przyjęcia stanowiska, czy proponowany projekt ustawy przyjąć, czy też go odrzucić. W związku z tym spotykamy się dzisiaj na debacie plenarnej, aby do tego tematu powrócić po raz kolejny. W istocie przy wprowadzaniu, przy dyskusji nad poszczególnymi punktami były bardzo duże rozbieżności w stanowiskach poszczególnych klubów parlamentarnych, posłów i one skutkowały zgłaszaniem poprawek lub też ich negowaniem, negowaniem poszczególnych artykułów w projekcie ustawy. W związku z tym, proszę państwa, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podtrzymuje swoją deklarację, że ten projekt rządowy jest projektem dobrym i projektem potrzebnym. Ale jak to bywa na posiedzeniach poszczególnych komisji, pojawiają się również wątpliwości, które trzeba rozwiać, które trzeba doprecyzować, bo przecież po to są właśnie posiedzenia komisji, aby nad projektami poszczególnych ustaw debatować, dyskutować. I niewątpliwie, mimo że było to posiedzenie długie, nie można było tutaj odrzucić jak gdyby stwierdzenia, że nie było ono merytoryczne. Mogliśmy się oczywiście z poszczególnymi sprawami zgadzać bądź też nie. Ale w związku z tym, że niektóre artykuły zostały wykreślone, w związku z tym, korzystając z okazji, że w kolejnym czytaniu można tę ustawę uzupełnić, polepszyć, sprawić, żeby ona była jeszcze bardziej Bo przecież o to tutaj chodzi, żeby rząd miał. takie mechanizmy, które mogłyby być mechanizmami skutecznymi, dobrymi, właściwymi, również - co było też podkreślane - w sytuacji, w jakiej w tej chwili znalazła się nasza ojczyzna, a więc w sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Proszę państwa, żeby nie przedłużać, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałem złożyć poprawki do proponowanej ustawy, do przedmiotowej ustawy.

Panie marszałku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Tomasz Szymański, klub Koalicja Obywatelska.

I ta ustawa również dotyczy, szanowni państwo, pieniędzy, z tym że nie dla was, drodzy Polacy, drodzy rodacy, tylko kasy dla swoich. Celem, który przyświecał tej ustawie, zdaniem pana ministra Dworczyka jest oczywiście przygotowanie pewnych ram do zapewnienia właściwego funkcjonowania rządu, wprowadzenia nowych działów, ale nie zapomniał wspomnieć, że tutaj kluczową sprawą jest jednak podniesienie apanaży, jest upolitycznienie członków korpusu. służby cywilnej, co spowoduje jej bardzo mocne ograniczenie merytoryczne. Szanowni państwo, to, co powiedział pan poseł Frysztak jako sprawozdawca komisji, ma absolutnie kluczowe znaczenie, ponieważ podniesienie wynagrodzeń dla podsekretarzy stanu o niebagatelną kwotę przewyższającą 10 tys. zł miesięcznie i umożliwienie, szanowni państwo, dodatkowego zarabiania pieniędzy, a także konieczność albo brak konieczności ujawniania swoich źródeł dochodu poprzez nieujawnianie tzw. oświadczenia majątkowego powodują to, że mamy do czynienia z bardzo dużym ograniczeniem i upolitycznieniem członków korpusu służby cywilnej. Szanowni państwo, mamy również pozorne zmiany, które w sposób jednoznaczny, tak jak powiedziałem, pozornie np. likwidują Ministerstwo Sportu i Turystyki, zastępując je ulubionym przez państwa tworem narodowym, kolejnym, Narodowym Centrum Sportu. Oczywiście nic się nie zmienia, kasa zostaje ta sama, hierarchia, funkcjonowanie, aparat jest ten sam. Szanowni państwo, ponieważ wrzuciliście tę ustawę, klasycznie przyzwyczajając nas do tego, na 2 dni przed, stawiając nas pod ścianą, ze zmianą dotyczącą kilkudziesięciu ustaw, ze 112 artykułami, które odnoszą się do kilkudziesięciu ustaw, z wieloma zmianami, musieliśmy się skoncentrować na tym, co uszyliście, specjalnie zaszywając głęboko w tę ustawę - to kasa, kasa dla swoich. Jeszcze raz, szanowni państwo, musimy o tym powiedzieć w sposób jednoznaczny. W dobie kryzysu, w dobie pandemii, w dobie niepewności bytu dnia codziennego dla Polek i Polaków, szanowni państwo, po raz kolejny robicie to, co dla was jest najcenniejsze - wpychacie do kieszeni publiczne pieniądze przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli, do swoich kieszeni. Próbujecie powiedzieć, że od dzisiaj ci ludzie, będąc waszymi aparatczykami partyjnymi zainstalowanymi w ministerstwach, od razu, z dnia na dzień, staną się bezpartyjnymi, merytorycznymi członkami korpusu służby cywilnej. To jest przecież parodia. Tylko pytanie: Czego? Czy tego, co państwo proponujecie w tej ustawie, czy po prostu korpusu służby cywilnej, z wieloma porządnymi apolitycznymi, merytorycznymi urzędnikami? Będzie to swoisty most pomiędzy polityką a korpusem służby cywilnej. Szanowni państwo, absolutnie nie ma naszej zgody na tego typu reformowanie, na tego typu przygotowywanie ustaw, kiedy ma się kilkadziesiąt godzin, proceduje się po nocach, jest wiele pytań, wiele niejasności, pomieszanie z poplątaniem.

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ w dobie epidemii, zamiast pomagać branżom, które zamykacie, takim jak gastronomia, piloci wycieczek, przewoźnicy, wy podnosicie wynagrodzenia dla swoich, w KPRM biurek wam zabraknie, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panowie Posłowie! Po pierwsze, chciałbym bardzo podziękować wszystkim państwu za te ponad 5 godzin pracy, ale nie musielibyśmy, panie ministrze, spotykać się trzykrotnie, bo przypominam, że przecież w sprawie tej ustawy spotkaliśmy się trzykrotnie. Pierwszy raz, kiedy komisja odrzuciła ustawę w całości, a potem dwukrotnie, aby nad nią procedować. Gdybyśmy mieli ekspertyzy, analizy i opinie. I tu, panie marszałku, również do pana apel, żeby w sytuacji, kiedy rzeczywiście rozpatrujemy projekty, Biuro Analiz Sejmowych przygotowało nam opinię, bo do tego projektu takiej opinii po prostu nie było, chodziło o szybkie procedowanie. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, panie ministrze, bo o reszcie będzie mówił mój kolega, poseł Szopiński. Inne wynagrodzenia będą mieli podsekretarze stanu w ministerstwie i kancelarii premiera, a inne wynagrodzenie, o połowę mniejsze, w kancelarii prezydenta i o połowę mniejsze podsekretarze stanu w Sejmie. A więc mamy dwie grupy podsekretarzy: tych lepiej uposażonych w ministerstwach i tych mniej w kancelarii prezydenta i w kancelarii Sejmu. Mówię tu o ciężkiej pracy osób, które dzisiaj funkcjonują w sanepidzie. Zgłosiliśmy poprawkę, aby oni również znaleźli się w tej kadrze służby cywilnej, na co nie było państwa zgody. Może po przemyśleniu podejmiecie jednak państwo decyzję, aby te dwa zawody - nie jest to duża grupa - również uwzględnić w zakresie stanowisk służby cywilnej. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sport z natury to rywalizacja, ale ta rywalizacja nigdy Polaków nie dzieliła.

Była też taka sytuacja, że nigdy nie dzieliło Polaków procedowanie nad ustawami, które obowiązują w zakresie funkcjonowania polskiego sportu. Ale do czasu, do czasu.

Ta ustawa zawiera aż 60 różnego typu zmian, zmian podstawowych w wielu ustawach: w ustawie o służbie cywilnej, w ustawie o bezpieczeństwie imprez, w ustawie dotyczącej służby zagranicznej. Ta ustawa to ustawa, która kryje właśnie w sobie zmianę dotyczącą funkcjonowania polskiego sportu. Szanowny Panie Marszałku! W uzasadnieniu tej ustawy czytamy: Celem zmian obejmujących przepisy dotyczące działu: Kultura fizyczna jest wprowadzenie sprawniejszego i nowoczesnego modelu zarządzania zadaniami z zakresu sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji poprzez organizacyjne i funkcjonalne wyodrębnienie zadań polegających na kształtowaniu polityki państwa w istotnej dziedzinie życia społecznego, jaką jest sport. Mianowicie na pytanie, z jakimi związkami sportowymi była ta ustawa konsultowana, odpowiem, że z żadnymi. Kiedy pytaliśmy pana ministra, z jakimi wybitnymi polskimi teoretykami w zakresie zarządzania sportem były konsultowane te zmiany, to otrzymaliśmy odpowiedź, że z żadnymi. Chciałbym zapytać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny przesuwa w kąt sprawę polskiego sportu i polskich sportowców, dlaczego nie potrafi usiąść przy wspólnym stole ze związkami sportowymi i uzgodnić, co dla polskiego sportu jest najlepsze. Wtedy, kiedy będzie sukces, będziecie razem na wspólnych zdjęciach ze sportowcami i z tymi związkami sportowymi. Będziecie fetować wtedy sukcesy. Ale wtedy, kiedy by trzeba opisać to, jak to w Polsce powinno wyglądać, to niestety was nie ma. Ja bym chciał pracownikom Ministerstwa Sportu z tego miejsca powiedzieć: Panie i panowie, przeczytajcie dokładnie tę ustawę, albowiem w tej ustawie dość niejasno jest powiedziane, czy będziecie pracować w (Dzwonek) Narodowym Centrum Sportu, czy w tym Narodowym Centrum Sportu pracować nie będziecie. Panie pośle, dziękuję. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po raz kolejny z tego miejsca mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koalicji Polskiej - PSL - Kukiz15 w odniesieniu do druku sejmowego nr 738 w sprawie rządowego projektu ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Tutaj przed moim wystąpieniem wybrzmiało dość mocno i głośno, że ustawa rzeczywiście budzi wiele wątpliwości i emocji, i nie tylko wybrzmiało to na trzech posiedzeniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, ale również na posiedzeniach Sejmu, również przed chwilą. Wiele tych niejasności i niedomówień wynika z niedoprecyzowania zapisów. Chciałabym powiedzieć, że na posiedzeniu komisji padło wiele pytań, padło wiele opinii, przedstawiono różne stanowiska. Trzeba uczciwie powiedzieć, że wiele z tych wątpliwości zostało wyjaśnionych i wiele merytorycznych dyskusji na posiedzeniu tej komisji zostało przeprowadzonych. Jednak trzeba też powiedzieć, że ustawa rzeczywiście przeprowadzona jest w trybie ekspresowym, w trybie szybkiego, bardzo szybkiego procedowania i bez opinii, bez opracowanych ekspertyz i konsultacji.

Generalnie sama ustawa w swoim zakresie obejmuje też wiele innych ustaw i dotyczy spraw przyporządkowanych do działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko. Obejmuje również zakresy i tematykę związaną z powstaniem działu: centrum administracyjne rządu.

Oczywiście w takim stanie rzeczy podsekretarze z uwagi na wymogi formalne będą musieli zrezygnować z przynależności politycznej. Problemem jest znaczne podniesienie wynagrodzeń. W dobie koronawirusa, w dobie wielu problemów związanych z walką z COVID-em, z pandemią, w dobie licznych problemów w systemie zdrowia, w systemie gospodarki naszego kraju wydaje się, że jest to działanie, które jest nie na miejscu i na pewno nie w tym czasie. Dlatego, używając bardzo, powiedziałabym, kulturalnych słów, chciałam bardzo serdecznie poprosić o to, aby podejść do tej kwestii w sposób racjonalny, wyważony, żeby wyciągnąć pewne wnioski. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Natomiast pozostają też pytania, czy procesy decyzyjne związane z przekształceniem czy też utworzeniem nowych ministerstw i nowych działów administracji będą rzeczywiście prowadzone szybko i sprawnie, czy nie będzie dochodziło do swoistego chaosu, jeśli chodzi o wydawanie decyzji administracyjnych czy też wcześniej ustalanie, do kogo te decyzje idą, do kogo poszczególne pytania w konkretnych zakresach będą kierowane. I rzeczywiście pytanie, czy zmniejszą się koszty funkcjonowania administracji rządowej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy tej ustawie przychodzi na myśl powiedzenie, że po to są działy i podziały, i rozdziały, żeby posły nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały.

Kiedy to mówię, to trzeba stwierdzić z takim smutkiem o charakterze państwowym, że 15 lat po tym, kiedy PiS szedł do władzy, wówczas z hasłem IV Rzeczypospolitej, czyli gruntownej, zasadniczej przebudowy struktur państwa na każdym poziomie funkcjonowania urzędów, mamy wielką kontynuację. To jest najbardziej miarodajny opis wbrew temu, co lewa strona sali lubi często wykrzykiwać, co wy w PiS-ie często lubicie podkreślać, że budujecie całkiem nowe państwo. Otóż państwo Prawa i Sprawiedliwości, otóż państwo Jarosława Kaczyńskiego jest w fundamentalny sposób kontynuatorem wszystkich złych naleciałości, patologii, zwłaszcza w tym sensie biurokratycznym, administracyjnym, III Rzeczypospolitej rządów Platformy, wcześniej SLD i poprzedników. To jest wielka kontynuacja niesprawności, wielka kontynuacja marnotrawstwa, wielka kontynuacja biurokratycznych absurdów i wielka kontynuacja tego, co najczęściej obywatele doświadczają w swoim życiu codziennym: państwa silnego wobec słabych, silnego wobec szarego obywatela i państwa słabego wobec rozmaitych sitw, układów, wielkich korporacji, państwa, które przez 5 lat nie potrafi zapewnić elementarnej swobody wypowiedzi i wolności słowa na platformach internetowych, ponieważ jest słabe wobec silnych, jest słabe wobec gigantów internetowych, państwa, które ściga sklepikarza, ściga handlarza, ściga właśnie szarego człowieka za byle bzdurę albo nakłada kilkanaście tysięcy mandatu za to, że się pojawił w parku bez maseczki, jak w tym roku, ale państwa, które nie potrafi realnie rozprawić się z mafiami, które sprawiają, że płoną śmietniska w całym kraju. Tego obrazu niestety dopełnia brak zdecydowanego centrum koordynacyjnego. Przypomnę, że za pierwszego PiS-u, w 2006 r., zlikwidowano Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, co zresztą było kontynuacją praktyki SLD-owskiej, i właściwie od tego momentu mamy do czynienia przez kolejne rządy i Platformy, i właśnie znowu PiS-u z jednym wielkim doraźnym działaniem, gaszeniem pożarów, działaniami pozorowanymi, działaniami PR-owskimi, jeśli chodzi o całokształt polityki państwowej.

Problem polega na tym, że szefem Centrum Analiz Strategicznych jest dzisiaj prof. Norbert Maliszewski. Jest specjalistą od marketingu politycznego.

Polska swoimi działaniami powoduje chaos. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, poseł niezależna. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zwierzęta to nie są rzeczy, a lasy to nie są pola ziemniaków. Polska przyroda to skarb, a nie zasób do zbójeckiej eksploatacji. Zabrakło na limuzyny? Oddaje je pod opiekę ministrowi rolnictwa, co prawdopodobnie oznacza erę masowych wycinek polskich lasów oraz odstrzału dzikich zwierząt na niespotykaną dotąd skalę. To ostatnie, czego potrzebuje nasza przyroda w obliczu kryzysu klimatycznego. Na pewno wymagają reformy, ale nie wycięcia w pień. Pamiętacie państwo taką piosenkę: był kiedyś maj, szumiał gaj? Jeśli przyjmiecie zapisy tej ustawy, to jedyne, co będzie słychać na terenach leśnych, to warczenie harwesterów. Czy naprawdę chcemy, żeby Polska stała się dugą Amazonią? Ochrona przyrody świadczy o odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i o patriotyzmie. To nasz konstytucyjny obowiązek. Polskie lasy należą do wszystkich obywateli. Ich wycinka nie może stanowić sposobu na łatanie dziur w budżecie.

To PiS barbarzyńsko najechał Puszczę Białowieską, a mówiąc o szkodnikach, niestety, nie myślał o sobie.

Dziękujmy niebiosom, że nie został ministrem zdrowia podczas epidemii.

Dzisiaj proszę was, Wysoką Izbę o uratowanie ich przed zaoraniem. Do pytań zgłosili się posłowie.

Wysoka Izbo!

Proszę państwa, włączenie podsekretarzy stanu do służby cywilnej to znowu de facto upolitycznienie tej służby.

Panie Ministrze! Rozmawiamy o działach administracji rządowej, ale zanim będziemy projektować kolejne zmiany, warto również zwrócić uwagę na to, jak obecnie funkcjonują działy administracji rządowej, szczególnie dział: sprawy wewnętrzne.

Te działania były szczególne, ponieważ funkcjonariusze nie byli umundurowani, nie byli oznakowani, a co najgorsze, używali siły fizycznej, używali pałek wobec pokojowo nastawionych manifestantów. W związku z powyższym mam pytanie do przedstawiciela premiera. Czy w tej sytuacji nie powinniście państwo popracować nad zmianami prawnymi. Pan poseł Jakub Rutnicki, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt tej ustawy to jest wyjątkowa bezczelność i cynizm władzy PiS. Dzisiaj, panie ministrze, 637 zgonów, a wy cynicznie nie publikujecie ustawy, która miała pomóc medykom, personelowi, jeżeli chodzi o podwyżki. Na to pieniędzy nie ma. Zamykacie gospodarkę, pozbawiacie ludzi pracy, szkoły są pozamykane. Szanowni państwo, ten projekt ustawy powinien się nazywać: podwyżki dla swoich.

Czy wam po prostu nie jest wstyd przed ludźmi? Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, klub Koalicji Obywatelskiej. Jest pani poseł? Pani poseł Anita Sowińska, klub Lewicy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgodnie z konstytucją pracownicy służby cywilnej powinni być apolityczni. Czy naprawdę sądzicie, że czynny polityk stanie się nagle neutralnym urzędnikiem? Zastanawia mnie, co chcecie uzyskać tym sztucznym zabiegiem. Zwracam się z pytaniem do pana ministra: Jaki jest prawdziwy cel tego zapisu o przeniesieniu podsekretarzy stanu do korpusu służby cywilnej? Czy chodzi o to, by móc pochwalić się pozornym odchudzeniem administracji rządowej i fikcyjnym zmniejszeniem kosztów funkcjonowania rządu? Przecież to jest tylko przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. A może jest to początek całkowitego upolitycznienia służby cywilnej i wstawiania tam swoich kolesi? Czy jeszcze wam mało stanowisk? Zachłanność PiS-u nie zna granic.

Wysoka Izbo!

I mam do pana pytanie: Czy prawdą jest, że podsekretarz stanu będzie zarabiał więcej niż każda nauczycielka w Polsce, każdy lekarz, znaczna większość lekarzy w Polsce, szczególnie lekarze rezydenci, pielęgniarki i te wszystkie razem wzięte osoby, które są zaangażowane w pomoc wszystkim tym, którzy tej pomocy od nas realnie potrzebują w walce z COVID-em? Poseł Artur Łącki, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wczoraj kolega Frysztak nazwał tę ustawę gniotem. Dzisiaj sobie pozwolę: gniot, bubel, byle co, bzdura, chała, słabizna i szmira. Ze względu na to mam dwa pytania. Dlaczego w dobie pandemii, czyli w dobie narodowego zaciskania pasa, pozwalacie swoim pracownikom, swoim członkom zarabiać ponad 20 tys. zł w randze podsekretarza stanu, a prawie 20 tys. zł członkom Rady Legislacyjnej? To jest jedna strona medalu. Dlaczego w art. 39 zmieniającym art. 52 ustawy o służbie cywilnej nie chcecie dopisać do katalogu wyższych stanowisk w służbie cywilnej wojewódzkiego inspektora sanitarnego i powiatowego inspektora sanitarnego, chociaż jest w tej ustawie wojewódzki i powiatowy lekarz weterynarii lub wojewódzki inspektor jakości handlowej?

Jakiś czas temu pan premier zapowiedział, że zmniejszy liczbę ministerstw. Miała być to taka zabawa w gorące krzesła, taka zabawa weselna. Ale przyszła ustawa o działach. Nie ma już zabawy w gorące krzesła, bo każdy, kto nie znajdzie pracy w ministerstwie, znajdzie ją w jakiejś spółce. Pytanie: Czy będziemy mieć mniej urzędników? Odpowiedź: nie, nie będzie mniej urzędników. Czy będą miękkie lądowania? Pan minister na to wcześniej nie odpowiadał. Czy podsekretarze stanu będą zarabiali więcej? Tak, będą zarabiali dwa razy więcej. Nikt nie mówi o publikacji ustawy COVID-owej, o dodatkach dla pracowników ochrony zdrowia. Pytanie do pana ministra: Dlaczego pan premier śpi?

Pan jest specjalistą do spraw tworzenia Szpitala Narodowego. 4 lata pracowałem w szpitalu. W związku z tym rozmawiam jak specjalista ze specjalistą. Pan wypowiadał się, dlaczego z jednej strony medycy, pielęgniarki, laboranci, ci, którzy są salowymi, nie mogą otrzymać podwyżki, bo pan premier nie publikuje ustawy, która została przez prezydenta podpisana 3 listopada. Niech pan dzisiaj z tego miejsca polskim służbom medycznym to powie. Prosiłbym, żeby pan owe oklaski przeobraził w decyzje.

A może przede wszystkim: Panie Ministrze!

Tej ustawy nie publikujecie, ale chcecie jak najszybciej, na nocnych posiedzeniach, przepchnąć ustawę, w której kolesiom dajecie po 10 tys. podwyżki. Ludzie, którzy w czasie epidemii na froncie narażają życie w szpitalach tymczasowych, ale również w tych prawdziwych szpitalach, a może przede wszystkim w tych prawdziwych szpitalach, w karetkach, salowe, pielęgniarki, lekarze - to są ludzie, którzy walczą o życie Polaków. Co pan powie salowym, pielęgniarkom i lekarzom?

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ten projekt to nic innego niż upartyjnienie kolejnych urzędów. Dążycie do tego, aby każdą kolejną ustawą zrobić z państwa polskiego swój folwark, folwark swojej władzy. Nie dość, że zarobki podsekretarzy będą astronomiczne, to jeszcze chcecie, żeby rozbudowana gałąź rad, doradców, szefów gabinetów była ponownie obsadzana i namaszczana przez wasz aparat partyjny. Jeżeli to jest działanie mające na celu odchudzenie rządu, to dajcie sobie spokój i przestańcie kłamać. Powiedzcie, ile jeszcze będziecie tworzyć tych stanowisk. To wszystko pokazuje, w jakiej desperacji jesteście, żeby zapewnić stołki swoim ludziom i żeby wasza chwiejna koalicja nie rozpadła się jak domek z kart. Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niszczycie oczywiście służbę cywilną. Konstytucja jasno reguluje w art. 153, że służba cywilna działa w celu zapewnienia rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań w państwie. Żadna z tych osób nie będzie robiła tego na pewno z naciskiem na: bezstronnie i politycznie neutralnie.

A wy proponujecie 10 tys. więcej dla swoich. Oprócz niszczenia służby cywilnej jeszcze robicie to. Co powiecie ludziom ze służby cywilnej, którym daliście po 100 zł?

Bardzo dziękuję. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przepycha przez Sejm kolejną nowelizację ustawy o działach administracji, to od razu wiadomo, że chodzi nie o poprawę państwa, nie o poprawę funkcjonowania państwa, nie o lepszą organizację, tylko o niszczenie i kolejne stołki dla swoich. Pod tym względem nic się nie zmieniło.

Kiedy dzisiaj przedsiębiorcy walczą o utrzymanie swoich firm, kiedy ludzie walczą o utrzymanie miejsc pracy, kiedy ludzie w szpitalach i ludzie wykonujący zawody medyczne ostatkiem sił ratują nas przed całkowitym załamaniem, wy zajmujecie się kolejnymi apanażami i kolejnymi stołkami dla swoich.

Panie Ministrze! Dzisiaj wszyscy wiemy, że wicepremier Gliński zajmuje się resortowo sportem, chcemy na mocy tej ustawy utworzyć Narodowe Centrum Sportu. Ale nie tak dawno, 13 listopada, pełnomocnikiem rządu ds. organizacji mistrzostw, igrzysk europejskich w Małopolsce w Krakowie został minister aktywów państwowych. Czy państwo nie boicie się, że te igrzyska padną? Czy to pełnomocnictwo zostanie przekazane później prezesowi centrum sportu, czy nie? Czy dalej pozostaje to u ministra Sasina? Jeszcze jedno pytanie.

Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska i Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę zadać pytanie. Czy zmiany wynikające z tej ustawy, która tylko pozornie likwiduje część etatów, a tak naprawdę przesuwa zadania i stanowiska, usprawnią pracę rządu? Czy przyniosą oszczędności? Czy stanie się wręcz przeciwnie - najpierw będą ogromne koszty związane z przystosowaniem nazewnictwa i całej administracji? Czy są policzone koszty dostosowawcze i koszty osobowe? Czy nie będzie tak, że te zmiany będą kosztowały nas, Polaków, o wiele, wiele więcej? Czy te koszty zostały policzone?

Wysoka Izbo! Przez ostatnich 5 lat PiS nie robi nic innego jak tylko likwiduje ministerstwa, tworzy nowe, kasuje stanowiska sekretarzy, podsekretarzy po to, żeby zrobić miejsce nowym aparatczykom PiS-owskim, żeby Zjednoczona Prawica się nie rozsypała do końca. Trzeba im dołożyć pieniędzy, dać limuzyny, wtedy zostaną, bo jak nie, to może będą szukać fruktów gdzie indziej. Niestety na tej reformie chyba najwięcej zarabiają drukarnie, bo oprócz tego, że drukujecie dużo pieniędzy, to jeszcze trzeba wydrukować tabliczki z nazwami ministerstw, z nazwami kolejnych funkcji, zajmowanych stanowisk. Tak to dzisiaj wygląda.

Dziękuję. Głos zabierze minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Rozumiem emocje, ja to wszystko rozumiem, ale pamiętajcie państwo o jednym: celem tej ustawy jest usprawnienie i zwiększenie efektywności działania administracji. Natomiast niestety w przypadku większości wypowiedzi, o czym powiem za chwilę, usłyszałem zupełnie coś innego. Oczywiście były takie wypowiedzi - z którymi mogę się zgadzać albo nie zgadzać - które były merytoryczne, odnosiły się do konkretnych faktów czy do konkretnych decyzji, propozycji zapisów, takie jak wypowiedzi pani poseł Gill-Piątek czy pana posła Szopińskiego. Ja się mogę nie zgadzać co do rozwiązań dotyczących sportu czy rozwiązań związanych z gospodarką leśną, ale to były wypowiedzi dotyczące meritum. Natomiast większość tych wypowiedzi, które tutaj padły, budzi po prostu niesmak i zażenowanie, bo proszę państwa, w przypadku większości wypowiedzi jest jeden cel, takie można odnieść wrażenie: budzenie nienawiści, populizm w najgorszym wydaniu, oskarżanie innych i szczucie na przeciwników politycznych. Proszę państwa, o ile wcześniej, wczoraj jeszcze, jak rozmawialiśmy, myślałem, że niektóre wasze wypowiedzi wynikają po prostu z niekompetencji, z tego, że nie przeczytaliście tej ustawy i OSR-u - a większość odpowiedzi na pytania, które się pojawiały, jest w OSR - o tyle dzisiaj wiem, że to jest właśnie inny cel, to jest cel wyłącznie polityczny. Nie wiem, może gdzieś przeczytaliście państwo, że wielokrotnie powtórzone kłamstwo w końcu staje się faktem, ale tak nie jest. Kłamstwa dotyczące np. zarobków Rady Legislacyjnej, które się nie zmieniają, i to wykazałem panu, panie pośle, wczoraj, pokazując projekt rozporządzenia na posiedzeniu komisji. Naprawdę czasami wstydzę się, bo przecież też jestem posłem, że taki poziom dyskusji na tej sali sobie fundujemy wzajemnie. Dziękuję bardzo. Głos ma sprawozdawca komisji pan poseł Konrad Frysztak. Dziękuję. Panie Ministrze! Powinien się pan wstydzić tego, że przyniósł pan do Wysokiej Izby takiego gniota. Powinien się pan wstydzić tego, że jest masa błędów, głupstw zapisanych w tej ustawie.

W KPRM-ie, tak jak powiedziałem, zabraknie wam biurek. Pytanie pani poseł Skowrońskiej, czy ta ustawa nadaje się do kosza. To jest podstawowy argument, pierwszy i podstawowy: podnosicie wynagrodzenia kolegom. Pan poseł Szymański pytał mnie o Radę Legislacyjną. Pan mówi, że to jest kłamstwo, że pan coś wyjaśnił. To gdzie znalazł się ten zapis dotyczący 20 członków z obecnie obowiązującego przepisu? Po prostu zdjęliście maksymalną liczbę członków. To, że dziś pokazuje pan jakieś rozporządzenie. Przecież wasze rozporządzenia, jak mówił wczoraj jeden z posłów, pojawiają się tak naprawdę w każdej chwili i ta ustawa jest na swój sposób usankcjonowaniem innych rozporządzeń. To są słowa pańskiego kolegi, za którego też pewnie powinien się pan wstydzić, ale czy się pan za niego wstydzi, nie wiem.

Tak, niesie za sobą taki wzrost wynagrodzeń. Tak, to będzie taki wzrost wynagrodzeń. Szanowni Państwo! Nie może być tak, że państwo w kilkanaście godzin chcecie przepchnąć ustawę zwiększającą wynagrodzenie w dobie kryzysu, w dobie pandemii.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki. proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Chciałbym raz jeszcze zwrócić się do pana z gorącym apelem.

Raz jeszcze zwracam się z uprzejmą prośbą do pana ministra o taką decyzję rządu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 734 i 737) Proszę panią poseł Agatę Wojtyszek o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 734. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 10 listopada 2020 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przeprowadzenia pierwszego czytania. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. wnoszą, aby Wysoki Sejm przyjął załączony projekt ustawy. Komisja pracowała zgodnie i po spokojnej, merytorycznej dyskusji znaczną większością głosów projekt przyjęta.

Celem projektowanych zmian jest przede wszystkim stworzenie nowych kategorii zadań, które będą dofinansowywane z tego funduszu, obejmujących zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które są w zarządzie prezydenta miasta, w którym znajduje się siedziba urzędu wojewódzkiego czy też sejmiku województwa. Do tej pory takich rozwiązań nie było, ta ustawa je zawiera.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwsza pani poseł Anna Milczanowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono mechanizm skutecznego rozwoju inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury drogowej. Zadaniem proponowanej ustawy, będącej dziś przedmiotem obrad Wysokiej Izby, jest wprowadzenie zmian mających na celu rozszerzenie katalogu zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane z wykorzystaniem środków tego funduszu. W projekcie ustawy przewiduje się wprowadzenie możliwości inwestowania tych środków z przeznaczeniem na zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tzw. zadania obwodnicowe, oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub marszałka sejmiku województwa, tzw. zadania miejskie. Ponadto ustawa ma wprowadzić mechanizmy promujące działania służące zwiększeniu liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i gminnych. Proponuje się wprowadzenie dodatkowej kategorii zadań dofinansowanych z funduszu mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Piesi są grupą uczestników ruchu drogowego szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo zdarzeń w ruchu drogowym. Statystyki wypadków z udziałem pieszych wskazują, że wskaźnik wypadków jest wyższy niż średnia unijna i wskaźniki większości krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z obecną praktyką inwestycyjną zarządców dróg traktuje się inwestycje w infrastrukturę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych jako element większych inwestycji. Natomiast niewiele jest mechanizmów umożliwiających finansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych bez konieczności przeprowadzenia dużych inwestycji drogowych.

W projekcie zakłada się także modyfikację sposobu określania źródeł finansowania funduszu z części budżetu państwa, których dysponentami są odpowiednio minister obrony narodowej oraz minister właściwy do spraw transportu. W miejsce dotychczasowej dotacji celowej proponuje się wprowadzenie wpłat na fundusz. Powyższe umożliwi uelastycznienie zasad przekazywania i rozliczania środków uzyskanych z budżetu państwa. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie zadań większych, które w większości wypadków mają charakter zadań wieloletnich. Wprowadzone zmiany nie wyłączą wydatkowania środków publicznych, którymi dysponuje fundusz, z właściwej kontroli. Dysponent funduszu nadal będzie zobowiązany do sporządzania rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego funduszu. Oprócz tego minister właściwy do spraw transportu będzie zobowiązany każdego roku przedstawić prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań funduszu. Poza tym zmiany w procedowanej teraz ustawie zapewniają dodatkowe inwestycje, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które również w wyniku pandemii mogły ponieść pewne straty, jak też jest to realna pomoc finansowa dla jednostek samorządu, samorządów przeróżnych, od gmin poprzez powiaty, urzędy marszałkowskie. Aby móc dokonywać drogich inwestycji drogowych, będzie możliwość ich finansowania. Wprowadzenie powyższych zmian w korzystny sposób wpłynie na dostosowanie zasad uzyskania dofinansowania z funduszu do rzeczywistego zapotrzebowania. Klub Prawo i Sprawiedliwość popiera uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie i proponuje wniesienie dwóch poprawek. Jedna, bardzo istotna, a mianowicie żeby zwiększyć listę rezerwową. Do tej pory, zgodnie z zapisami, które obowiązują dzisiaj, 50% listy rezerwowej to były te jednostki samorządu terytorialnego... 50% z listy podstawowej. A teraz chcemy listę rezerwową zwiększyć do puli 75% listy podstawowej, ponieważ mamy to doświadczenie, że w wyniku przetargów pozostają pieniądze, oczywiście na terenie danego województwa, i chcemy, żeby jak najwięcej beneficjentów [[Dzwonek]] z tego funduszu mogło skorzystać. Dziękuję. Panie Marszałku! Szanowni państwo, to jest też bardzo dobra okazja, żeby sprostować często powtarzane przez premiera Morawieckiego słowa, jakoby po rządach poprzednich, Platformy Obywatelskiej i PSL-u, zastał polskie drogi w ruinie i dopiero teraz, cytuję pana premiera, będzie budował na potęgę drogi. Oczywiście to jest kłamstwo.

Warto o tym powiedzieć, dlatego że dopiero pomysł pana ministra Schetyny - zresztą ta potoczna nazwa programu nie wzięła się przecież z kosmosu - dał nowe tchnienie polskim drogom lokalnym. Chcę powiedzieć, że dla Prawa i Sprawiedliwości drogi do tej pory nie były priorytetem.

Warto o tym również wspominać. Ale przechodzimy teraz do programu Funduszu Dróg Samorządowych, który rząd ogłosił jeszcze przed wyborami samorządowymi. Popatrzmy, jak były przekazywane pieniądze. Wystarczy posłuchać samorządowców. Zacytuję jednego z nich: To najmniej przejrzysty mechanizm dystrybucji środków publicznych, jaki poznałem w ostatnich latach, premier może bez konkretnego uzasadnienia dać komuś pieniądze publiczne, a komuś je zabrać. Jest mnóstwo przykładów, czytamy, jak są te pieniądze zabierane. Przykład: 6 mln zł dotacji dostał jeden z wójtów na remont drogi, okazało się, że nawet dostał pamiątkowy voucher, ale później pan premier wymazał. 11 innych samorządów z tego samego województwa - dokładnie to samo. Podpisali, zrobiono konferencję, a później się okazało, że premier wymazał. I to jest główny zarzut wszystkich samorządów, że de facto jest to bardzo uznaniowe. Jeden z profesorów, pan prof. Paweł Swianiewicz, w raporcie „Wspólnoty”, pisma bardzo ważnego dla samorządowców, tak oto opisuje ten program, który działa kilkanaście miesięcy: Przewaga dotacji otrzymywanych przez gminy, których władze powiązane są z PiS, jest bardzo wyraźna. Najmniejsze wsparcie otrzymują gminy rządzone przez ugrupowania opozycyjne. Więcej niż połowa tych gmin nie otrzymała żadnej dotacji. Tak właśnie wygląda dzielenie tych środków finansowych. I dodatkowo oczywiście jest problem, jeśli chodzi o przekazywanie tych środków i czas przekazywania tych środków, a więc nie tylko brak transparentności, ale również tempo uruchamiania tych środków. Sam program, oczywiście wzorowany na programie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jest bardzo dobry. Tym razem, pomimo że będzie to dotyczyło dróg samorządowych, rząd wpadł na pomysł, że wykreśli słowo: samorządowe, żeby był tylko rządowy fundusz. Proszę państwa, to jest po prostu taka czysta zagrywka tylko i wyłącznie PR-owa, żeby pokazać, że to rząd, chociaż przecież rząd tylko dofinansowuje, samorządy muszą przekazać część pieniędzy, żeby te inwestycje zostały zrealizowane. W związku z tym w imieniu Koalicji Obywatelskiej będę składał trzy poprawki. Druga poprawka dotyczy uniknięcia sytuacji, w której w bardzo krótkim okresie obwodnica staje się de facto drogą miejską, niepełniącą w żaden sposób swoich pierwotnych funkcji - chodzi o dokładne uszczegółowienie. I kolejna poprawka - chodzi o to, aby w jasny i klarowny sposób określić środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [[Dzwonek]] w kontekście przepisu art. 17. I takie trzy poprawki przedstawiam.

Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Fundusz Dróg Samorządowych to chyba takie ciche marzenie każdego samorządowca i każdego posła. Już oczami wyobraźni widzę, jak w dość szybkim tempie są budowane obwodnice Lipna, obwodnica Golubia-Dobrzynia, obwodnica Brodnicy, Rypina, jak powstanie trasa średnicowa w Grudziądzu, jak wreszcie, bo i tego obecnie ma dotyczyć ten fundusz, powstaje most zachodni w Toruniu - trzeci most drogowy, jak powstaje nowe połączenie drogowe z trzecim mostem we Włocławku. No marzenie. Marzenie oczywiście ograniczone, po pierwsze, skromnymi środkami budżetowymi, bo właściwie ja już w tej chwili wyczerpałem tę kwotę 3 mld zł, o jaką planuje się powiększenie tego Funduszu Dróg Samorządowych. I oczywiście ten projekt nie przejdzie, choćby znalazł swoje uzasadnienie w decyzjach komisji, ponieważ ten fundusz jest chyba najbardziej uznaniowym funduszem ze wszystkich funduszy celowych, które w Polsce funkcjonują. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Będziemy mianowicie rekomendować, by rezerwa pozostająca w dyspozycji prezesa Rady Ministrów została zredukowana z obecnych 5% do 1%. Druga uwaga, druga poprawka, którą klub Lewicy będzie zgłaszał, dotyczy samej nazwy. Rzecz nie jest bagatelna wbrew pozorom. Nazwa, którą się obecnie proponuje, jest ewidentnie myląca. Ten fundusz jest funduszem samorządowym, a nie tylko rządowym. Dotyczy zresztą, jeśli dobrze rozumiem, nie tylko rozwoju tych dróg, mostów i obwodnic, ale także ich remontu. Jeśli coś działa, naprawdę nie kombinujmy. Proponujemy, żeby zostawić dotychczasową nazwę. Być może i słusznie. Tu odwołam się do dorobku poprzedniej koalicji PO-PSL. To, co kiedyś zwane było schetynówkami, działało. Rozumiem, że ten fundusz jest jakby wzorowany na tym pomyśle. Trzeba chwalić poprzedników, a nawet konkurencję wtedy, kiedy te pomysły miała dobre i skuteczne. Żałuję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy tego typu kultury politycznej uprawiać nie chce, nawet na tak pozornie neutralnym gruncie, jakim jest infrastruktura, jakim są drogi. Wysoka Izbo! Cieszę się także, i to warte jest także podkreślenia, że nacisk kładzie się na to, co jest osiągalne, co jest realne, bo jeśli ja byłem w stanie przed chwilą wymienić tyle projektów infrastrukturalnych z dziedziny dróg, to jestem przekonany, że każdy z obecnych tu posłów jest w stanie przedstawić swoją listę życzeń czy listę marzeń, a to oznacza, że powoli żegnamy się z kosmicznymi planami rządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącymi Centralnego Portu Komunikacyjnego zwanego w tej części lotniczej Centralnym Portem Lotniczym Baranów. Życie niestety, także za sprawą pandemii, zweryfikowało te plany. Być może moduł kolejowy zostanie, i fajnie, a być może te wszystkie środki, które były planowane, a przynajmniej ich znaczna część była planowana, na port lotniczy, zostaną przekazane w ten czy inny sposób na Fundusz Dróg Samorządowych. Jestem przekonany, że one zostaną wykorzystane i szybciej, i sprawniej, i z większym pożytkiem dla obywateli, dla naszych wyborców. Jeszcze jedna uwaga, całkiem na marginesie. Tłumaczono mi oczywiście, że Krajowy Fundusz Drogowy i ten fundusz, o którym my w tej chwili debatujemy, czyli Fundusz Dróg Samorządowych, to są jakby fundusze celowe z różnych światów i różnych bajek. Zauważam jednak, że przede wszystkim łączą je użytkownicy, beneficjenci, łączy pewna logika, o którą warto dbać nie tylko na poziomie ministra właściwego do spraw transportu czy Ministerstwa Infrastruktury. Być może ta koordynacja, której brakuje, mogła być tutaj lepiej przeprowadzona.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska dotyczące sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Może zacznę trochę od historii, bo pomysłodawcą tego był mój sympatyczny kolega z klubu Jan Łopata, który zaproponował ówczesnemu premierowi takie rozwiązanie, później od nazwiska ministra Schetyny - schetynówki.

Wszystko musi być rządowe. Wszystko musi być narodowe. Są samorządy, które budowały drogi i budują ciągle. My jako przedstawiciele samorządów, ale też wcześniej działający w rządzie, uważaliśmy, że drogi nie są polityczne. Drogi PiS-ie, samorządowcy od was też dostawali pieniądze, jeżeli mieli projekt, jeżeli chcieli zbudować drogę, bo to ma służyć wszystkim Polkom i Polakom.

To nie dajmy mu pieniędzy - tak w ostatnim czasie robiliście. Co do zasady to są potrzebne zmiany. Trzeba budować obwodnice na drogach wojewódzkich. Jeśli zaangażujecie w to samorządy, może wam się uda.

Oczywiście jak samorządy to zrobią i te pieniądze przekażecie, uda się. Miało być dofinansowanie do przewozów autobusowych, a dzisiaj pieniądze idą na drogi. Nie chcecie dofinansować przewozów autobusowych. Ludzie nie chcą korzystać z waszego programu. Coś jest nie tak. Dalej szukamy. Oczywiście gospodarstwo leśne Lasy Państwowe. Jak my proponowaliśmy te pieniądze, to PiS oskarżał, że chcemy ograbić lasy, że chcemy prywatyzować te lasy. Dzisiaj sięgacie po te pieniądze, żeby te drogi, obwodnice budować. Wiadomo, te pieniądze można przeznaczyć na wszystko, tak jak w przypadku Funduszu Sprawiedliwości, który powołaliście. Dzisiaj też te pieniądze będą przesypywane z jednej kieszeni do drugiej. Chcemy przebudowywać drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Chodzi oczywiście o zwiększanie bezpieczeństwa pieszych. Ogólnie zwiększanie bezpieczeństwa na drogach powinno nas wszystkich łączyć. Dlatego też oczywiście poprzemy ten projekt, zagłosujemy za tymi wszystkimi też poprawkami zgłoszonymi podczas komisji, bo one są potrzebne. Chcecie się wykazać dobrą wolą w przypadku współpracy z samorządami, ale jeszcze raz przypomnę to, o czym mówiłem na początku: nie tylko ze swoimi samorządami, ale ze wszystkimi. Współpraca rządu i samorządu być powinna. Związek Gmin Wiejskich, tak jak związek powiatów, związek miast, mówi, że dobrze, że te zmiany się pojawiają. Więcej będzie można zrobić, wybudować, wyremontować tych dróg. Ale od samej zmiany ustawy nic się nie zmieni.

Jeśli będziecie się upierać, tym samym pokażecie, że opozycji w żadnej, nawet najprostszej rzeczy nie słuchacie. A później mówicie, że to my nie chcemy z wami współpracować. Pan poseł Dobromir Sośnierz, koło Konfederacji. Budowa dróg to jedna z tych dziedzin, którymi państwo zajmować się niestety musi, co nawet najwięksi wolnościowcy raczej w większości przyznają. Tutaj macie szansę się wykazać w praktyce. Jednak państwo, które próbuje się zajmować wszystkim, niczym nie zajmuje się w końcu dobrze.

Mamy beznadziejne drogi, słaby sport, umierająca sztukę, a biurokracja przeszkadza wszystkim po kolei: lekarzom, rolnikom i piekarzom w pracy. Ale też nie twórzmy wokół tego iluzji czy złudzeń, że to nam rozrusza gospodarkę w kryzysie. Pieniądze na drogi to pieniądze zabrane obywatelom w podatkach, jak wszystkie pieniądze, które ma rząd. Gdyby nie zostały zabrane, też by zostały wydane przez obywateli tylko na coś innego, akurat nie na drogi.

Ale tu i teraz to gospodarki nie rozrusza, tylko zamieni jedne wydatki, których dokonaliby obywatele, na inne, te, których dokona rząd, czyli w tym przypadku na drogi. Nie jest to oczywiście argument przeciwko tym wydatkom, przeciwko drogom, oczywiście drogi to dobre inwestycje na przyszłość, ale przestańmy powtarzać ten fałszywy argument, który tu się w kółko pojawia w różnych rządowych uzasadnieniach, w tym pojawia się również, że to jest rozruszanie gospodarki.

To nie pan minister, nie posłowie na to zarobią, tylko obywatele, którym się w tym przeszkadza. Mamy coraz mniej pieniędzy ze słabnącej gospodarki, a nie słyszałem w żadnym przypadku o tym, że zamierzamy z czegoś w takim razie zrezygnować w tych trudnych czasach, coś ograniczyć. Co do samej ustawy, to jedna rzecz budzi ogromne zastrzeżenia. Pieniądze, które mają iść na drogi, na rozbudowę dróg, zgodnie z tą ustawą, będą też przeznaczane na ich dewastację, czyli na zakładanie progów zwalniających.

Progi zwalniające to jest karanie wszystkich za to, że niektórzy jeżdżą źle. Wszyscy musimy oblewać się kawą na tych wertepach, niszczyć zawieszenie, bezsensownie wytracać prędkość do 10 km/h, bo większość tych progów jest tak skonstruowana, że de facto wymusza prędkość znacznie poniżej dopuszczalnego na tym odcinku limitu, tylko dlatego, że samorządy i rząd źle projektują przejścia, źle, bez wyobraźni regulują ruch, a potem zrzucają zawsze winę na kierowców. To jest droga donikąd. Po niektórych miastach już teraz jeździ się jak na pewno na safari w Kenii, bo co chwilę próg, zwężenie, szykana, remont. Jeśli chcecie naprawdę zadbać o pieszych, to proszę wziąć pod uwagę kilka rzeczy, np. może trzeba zrezygnować z głupiego pomysłu jazdy na światłach w dzień, bo Austria wycofała się m.in. z tego powodu z tego nieszczęśliwego pomysłu, że zauważono, że wprawdzie tam nieznacznie spadła ilość wypadków na drogach, ale zwiększyła się ilość potrąceń pieszych, bo piesi nie świecą na drodze. Kierowcy przyzwyczajają się do obserwowania świecących przedmiotów, obiektów. Jeśli naprawdę chcecie zadbać o pieszych, to może trzeba wziąć pod uwagę zmianę systemu działania OC, bo w tej chwili OC zdejmuje ze sprawcy właściwie cały ciężar odpowiedzialności. Jeśli w ogóle ma to pozostać obowiązkowe, to może dobrym pomysłem byłoby zmienić zasady w tej sposób, żeby roszczenia wobec sprawcy, przynajmniej ciężkiego wypadku, gdzie wina nie budzi wątpliwości, były najpierw zaspokajane z jego majątku, a dopiero po wyczerpaniu jego możliwości finansowych, po sprzedaniu już ostatniej pary butów, z polisy OC. Oczywiście polisa powinna być wtedy tańsza, ale to już inny temat. Gdybyśmy mogli się ubezpieczyć od pójścia do więzienia, to byłoby pewnie więcej przestępstw, a nie mniej. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do zadawania pytań. Proszę państwa, z racji tego, że obrady dzisiaj nam się kroją do godz. 3 mniej więcej. 20 osób się zgłosiło do zadawania pytań i mam pytanie, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby się zgłosić? To jak państwo pozwolicie, zamykam listę, ze względu na godzinę. Tak, bardzo proszę, 21 osób.

Proszę państwa, 21 osób. Bardzo proszę, żebyście nie mieli pretensji. Pan poseł Krzysztof Gadowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Ustalam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przez te lata, kiedy rządzicie już 5 lat, pokazujecie, że program był dobry. Oczywiście trzeba go zmieniać i dobrze, że to robicie, że dokładacie więcej pieniędzy, które dzisiaj można na te cele przeznaczyć.

Czy państwo nie myślicie o tym, żeby podejść jakoś bardziej normalnie w tym czasie kryzysu do tematu tych dróg? Chciałem pana zapytać, czy dobrą metodą jest to, że państwo dopiero decyzję podejmiecie w przyszłym roku. Przecież samorządy budują, budżety uchwalają jeszcze w tym roku, do 15 listopada muszą zawrzeć. Czy ten temat decyzyjny podjęcia ewentualnie ostatecznej decyzji państwo będziecie się starać podejmować jeszcze w okresie tym budżetowym, kiedy gminy mogą uchwalać budżet, czy nie, bo, tak jak powiedziałem, złożone zostały jeszcze sierpień, wrzesień bodajże, do dzisiaj nie ma informacji. Pozdrawiamy starostwo. Pani posłanka Katarzyna Kretkowska, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Powiększenie tego funduszu, a także powiększenie tego funduszu o takie zadanie jak obwodnice, mosty, wiadukty jest bardzo celowe. Także powiększenie tego funduszu o miasta na prawach powiatu będące siedzibą województw jest bardzo celowe i było oczekiwane przez samorządy.

Budowa trzeciej i czwartej ramy, czyli obwodnicy miasta Poznania jest mało realna w kontekście przyszłego roku. Każda z tych obwodnic kosztowałaby 3 mld.

I ostatnie pytanie: Co z rozbudową drogi wojewódzkiej 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo, Mosina?

Proszę państwa, ja mam serdeczną prośbę, bo dwa pierwsze pytania były po półtorej minuty. Ze względu na posłów i posłanki, którzy będą siedzieć do godz. 3, po prostu będę grzecznie, ale stanowczo przerywał po minucie. Pan poseł Andrzej Szewiński, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ta inwestycja doprowadzi do wyprowadzenia tranzytu z centrum miasta.

Dzięki właściwym decyzjom decydentów marzenia te mogą się spełnić. Proszę. Wysoka Izbo! Zabraliście pieniądze na budowę dróg miastom na prawach powiatu takim jak Lublin, o czym wielokrotnie mówiłam. Ale macie także szansę naprawić to, co ostatnio zepsuliście w Lublinie i na Lubelszczyźnie, bo pozbawiliście pomocy i wsparcia Port Lotniczy Lublin w związku z kryzysem wywołanym epidemią, mimo że jeszcze w czerwcu w odpowiedzi na moją interpelację ministerstwo zapewniało o tej pomocy. Dlaczego tak kłamiecie? Dlaczego miała być pomoc, a teraz nie ma pomocy? Lubelszczyzna, najbiedniejszy region w Polsce i w Unii Europejskiej, nie otrzyma pomocy, bo według ministerstwa strata wykazana przez port lotniczy nie mieści się w definicji straty. To po prostu absurd. Panie Premierze! Panie Ministrze! Panowie Ministrowie z Lubelszczyzny!

Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Myśmy zastali po was Polskę drewnianą, a zostawiliśmy Polskę, która ma normalną komunikację na poziomie europejskim.

2 lata opóźnień w budowie drogi S3, którą wam zostawiliśmy, na odcinku Polkowice-Lubin. Giną tam ludzie. 2 lata opóźnień i nie możecie tej drogi skończyć.

Zgłoszę stosowną poprawkę, aby to miejsce było bezpieczne dla mieszkańców Lubina i Dolnego Śląska. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Dziś pracujemy nad zmianami w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy coraz lepsze drogi gminne i powiatowe. Naprawdę jest czym się pochwalić, wystarczy pojechać w Polskę. Mam też do pana ministra bardzo konkretne pytanie. Pan minister właściwy, minister infrastruktury, może określić maksymalną liczbę wniosków składanych przez poszczególne samorządy województw dotyczących dróg w ciągu dróg wojewódzkich i obwodnic.

Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Ryszarda Wilczyńskiego, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! To się teraz dzieje. Nie w całym zakresie, ale w pewnym zakresie.

Zmieści się to w limicie 100 mln zł, natomiast prezydent Opola musi wydać 60%, a marszałek - 40%.

Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeszcze w tym roku Fundusz Dróg Samorządowych, a parę lat temu tzw. schetynówki. Były one pomyślane w ten sposób, żeby dać pieniądze tym samorządom, które nie mają środków własnych, a mają najwięcej dróg do wyremontowania, czyli były pomyślane po to, żeby pomóc w remontach tych dróg szczególnie powiatom, ale też gminom.

Myślę, że chodzi o miasta duże, wojewódzkie i na prawach powiatu.

Nie możemy porównywać powiatu z województwem, dlatego że województwo ma inne środki, inny przychód, inne pieniądze, ma choćby pieniądze unijne na remonty dróg. Powiat nie ma żadnych pieniędzy. Ja się martwię o powiaty ziemskie i o gminy. Mam pytanie: Czy nie uszczupli to pieniędzy na remont dróg powiatowych i gminnych? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście przepisy idą w dobrym kierunku i myślę, że co do tego się zgadzamy. To dobrze, że ministerstwo podążyło tym tokiem myślenia, bo - jak myślę - to dobrze dla funduszu i dla rozwoju dróg. Chciałem pana ministra zapytać o to, jak będzie z przejściami dla pieszych, bo uważam, że kwestie budowania przejść dla pieszych, infrastruktury. Może prosiłbym o zatrzymanie czasu. panie ministrze? Nie wiem, dlaczego pan minister rozmawia teraz przez telefon. Chodzi o przejścia dla pieszych, o to, czy będą wydane jakieś nowe wytyczne dotyczące budowy dróg, bo to jest oczywiście lepszy kierunek niż jakieś (Dzwonek) określenie tego przepisami. Dwie uwagi, jeżeli pan marszałek z uwagi na ten incydent pozwoli. Ja jednak, panie ministrze, uważam, że to jest taki wyraz małostkowości, bo tak naprawdę, gdybyśmy przeszli do sedna, to to powinien być społeczny fundusz, bo jest z naszych podatków i z podatków osób pracujących. Natomiast art. 5, dotyczący rozwoju przewozów autobusowych i tych środków, uważam za dosyć mocną porażkę rządu. Szkoda, że ministerstwo nie usiadło z nami i z samorządami. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd zamierza zmienić Fundusz Dróg Samorządowych w Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Już sama zmiana nazwy pokazuje sposób myślenia obecnej władzy, która krok po kroku demontuje samorządność, pozbawiając ją autonomii i decyzyjności. Do funduszu włączone zostaną miasta na prawach powiatu, a premier będzie miał prawo usuwać i dodawać projekty z listy, a także rozdysponować 5% środków z funduszu rezerwy. Samorządowcy zwracają uwagę, że wątpliwości budzi także proces wyboru projektów. Dlatego mam pytanie: Czy i w jaki sposób zmiany ujęte w projekcie były konsultowane z samorządami? Niestety znamy odpowiedź: nie były. Przestańcie twierdzić, że wszystko wiecie lepiej od samorządów. O remoncie drogi, skrzyżowania czy przejścia dla pieszych powinny decydować lokalne władze, a nie minister czy premier gdzieś tam w oddalonym urzędzie. Już kończę. Panie Ministrze! W tym tygodniu w całej Polsce odbyły się protesty, podczas których przewoźnicy prosili o jakiekolwiek wsparcie. Dziesiątki tysięcy kierowców mogą stracić pracę. Dlaczego tak łatwo rezygnujecie ze wsparcia transportu zbiorowego, który mierzy się z największym od lat kryzysem? Dziękuję. Przepraszam posłankę i posła, których nie dopisałem, ale umówiłem się z salą, że już nie dopiszę, pamiętacie państwo. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! PiS postanowił bohatersko rozszerzyć swoje kompetencje o możliwość budowania obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tak jakby dotychczas nie było to możliwe na dużo prostszych zasadach. No ale PR to jest to, co najlepiej temu rządowi wychodzi. A ja bym radził, żeby PiS zaczął wywiązywać się z obietnic, chociażby z ostatnich wyborów, np. ze 100 obwodnic. Niedawno zapytałem dyrektora krajowej dyrekcji w Łodzi o budowę obwodnic w województwie łódzkim.

Mogliście równie dobrze obiecać, że to opozycja wybuduje tę obwodnicę, jak dojdzie do władzy. Podczas ostatnich wyborów obiecaliście, że wszystko już jest gotowe. A obwodnica Tomaszowa Mazowieckiego?

Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Konkretne pytanie: Czy w przypadku realizacji obwodnic w etapach ze względu na koszty możliwe będzie dofinansowanie kolejnego etapu, niekoniecznie całości tego zadania?

Nie likwidujcie stoczni w Świnoujściu. Tam nadal pracuje 200 osób. Ci ludzie chcą nadal pracować i remontować te statki. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Konrad Frysztak, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę serdecznie. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jestem z Radomia. Jako były wiceprezydent miasta Radomia chciałem panu powiedzieć, że nakładami wynikającymi z decyzji rządu Platformy Obywatelskiej w Radomiu wybudowaliśmy nową siedzibę sanepidu. Jako wiceprezydent wnioskowałem do Funduszu Dróg Samorządowych utworzonego przez państwa, przez wasz rząd, tak naprawdę przekształcony z dobrego programu schetynówek, o budowę ul. Zgodnej i ul. Piwnej. Nie dostaliśmy, szanowni państwo, dlatego że PiS te pieniądze daje swoim. Daje swoim samorządom i taki zarzut był wobec was wielokrotnie kierowany przez Związek Miast Polskich, którego również Radom jest członkiem, a ja pracowałem w jego zarządzie.

Pani posłanka Mirosława Nykiel, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Lepiej późno niż wcale - głosi porzekadło. Panie ministrze, mam pytanie o trzy kluczowe inwestycje z mojego okręgu wyborczego. Węzeł drogowy w Pszczynie łączący drogę krajową znajduje się w programie dla województwa śląskiego i w strategicznym planie odpowiedzialnego rozwoju, jest częścią.

No i Szczyrk, proszę państwa, poszerzenie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, ul. Beskidzkiej, z powiatową. Czy te trzy inwestycje, panie ministrze. Jest ich o wiele więcej, ale z uwagi na czas nie zdążyłam zadać wszystkich pytań. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Słuchamy was, bo tyle razy zwracaliście uwagę, żeby drogi wojewódzkie były tu ujęte, żeby w miastach, gdzie ma siedzibę wojewoda, marszałek, też można było remontować drogi, i te zapisy zostały wprowadzone, dodatkowe pieniądze zostały wprowadzone. Sukces ma wielu ojców, drodzy państwo, ale to rząd Prawa i Sprawiedliwości odważył się wprowadzić taki fundusz z ogromnymi pieniędzmi. To nie jest 800 mln w skali roku.

Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie marszałku. Panie Ministrze!

Jakie kwoty były przeznaczone na wsparcie dla samorządów na realizację tych inwestycji? Jak to się po prostu ma do kwot w poprzednich latach, w poprzednich programach realizowanych, zanim powstał ten program, o którym dzisiaj mówimy? Pani poseł Lidia Burzyńska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Ja wiem, że dyskusja, debata powinna być na argumenty, a nie na przerzucanie się nieprawdami, półprawdami albo nawet kłamstwami. Posłom z mównicy, szczególnie z opozycji, tak łatwo przechodzi przez usta to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego dzieli i daje tylko pisowskim samorządom, daje tylko swoim. Daję przykład: jestem mieszkanką powiatu częstochowskiego i szanowny panie, mój powiat jest zarządzany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, [[Oklaski]] i wie pan, ile otrzymał właśnie teraz na zadania z Funduszu Dróg Samorządowych? 27 mln na trzy inwestycje, które będą realizowane w przeciągu 3 lat. Niecałe 3 mln. Gdzie teraz brawa bijecie, nie bijecie braw? Pan poseł Dariusz Joński, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiązując do licznych wypowiedzi odnośnie do przekazywania środków i decydowania przez premiera, chcę powiedzieć, że wójtowie przesyłali to do wojewody, wojewoda zazwyczaj zgłaszał inwestycję drogową, ale jak już to lądowało w ministerstwie i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to premier brał długopis i tym długopisem wymazywał.

Natomiast chciałbym państwu zacytować pana Krzysztofa Sobolewskiego, który mówił: Jeśli zatem któryś z senatorów opozycji obiecał np. budowę hali sportowej, to gdy zgłosi się teraz do PiS, to rząd znajdzie na to pieniądze, taki senator będzie miał dużo większe szanse, że projekt będzie zrealizowany, będąc w obozie rządzącym, a nie w opozycji. Jak nie będziecie u nas, to wam nie damy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, panie pośle. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Bożenę Żelazowską z klubu parlamentarnego PSL-Kukiz15. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Trudno jest znaleźć powód, dla którego ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych ma teraz nagle nosić nazwę: o funduszu dróg rządowych. Możemy się go tylko domyślać. Mam pytanie. Na jaki cel będzie przeznaczone 5% rezerwy, która ma pozostać w dyspozycji prezesa Rady Ministrów? Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć tę kwotę na budowę dróg? Wiemy, że samorządy w dzisiejszym trudnym czasie są wyjątkowo obciążone - ciągle nowe zadania, ciągle nowe podatki. Myślę, że wszystkie 16 województw dostanie dofinansowanie na budowę dróg. Chciałaby, żeby tak się stało, i właśnie o to wnioskuję. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Rafała Webera. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 5 minut to naprawdę zbyt mało czasu, aby odnieść się do wszystkich zagadnień i pytań, które padły w tej gorącej dyskusji. W pierwszej części swojej wypowiedzi pozostanę w konwencji historycznej, bo warto przypomnieć, co się działo w przeszłości i w jakim stanie rząd Prawa i Sprawiedliwości zastał lokalne drogi. Argument nr 1, szanowni państwo - raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2014. Wtedy prezesem NIK był już były poseł, były minister Platformy Obywatelskiej, pan Kwiatkowski.

To jest raport Najwyższej Izby Kontroli przygotowany przez prezesa Kwiatkowskiego, to jest raport wstydu waszej władzy, raport wstydu pokazujący wszystkie działania, których nie prowadziliście na polskich drogach samorządowych.

Tylko w ciągu roku przeznaczyliśmy na drogi gminne i powiatowe więcej [[Oklaski]] niż wy w ciągu 8 lat.

To są, szanowni państwo, fakty, to są liczby.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych w chwili obecnej to 36 mld zł.

Jeszcze jeden temat, jeszcze jedno hasło.

My tą ustawą chcemy przekierować na Fundusz Dróg Samorządowych to, co zostanie, żeby środki, które zostały ciężko wypracowane, zostały przeznaczone na inwestycje drogowe, a nie wróciły do źródeł, z których pochodzą. Tak że myślę, że to bardzo pozytywne rozwiązanie. Szanowni Państwo! Teraz przedstawię, jeżeli moi koledzy będą w stanie mi pomóc, listę sukcesów.

To jest 30-metrowa płachta.

Porozmawiajcie z tymi samorządowcami, porozmawiajcie z wójtami, ze starostami, porozmawiajcie z radnymi, sołtysami.

chcemy wygenerować środki finansowe, dzięki temu, że potrafimy to zrobić, i dzięki temu, że jesteśmy wiarygodni.

Bardzo gorąco dziękuję.

Jeszcze raz powtarzam: będziemy pisać tę historię nadal, będziemy wspierać polskie samorządy, gminy i powiaty.

To są drogi, którymi codziennie dociera się do szkoły, do pracy, do sklepu, do kościoła, do ośrodka kultury, do ośrodka zdrowia.

Ten proces pomimo epidemii koronawirusa, pomimo. Zobaczcie państwo, w jakim jesteśmy momencie.

Dziękuję serdecznie.

Proszę uprzejmie, grzecznie. Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o obwodnice, chociażby w dniu wczorajszym został ogłoszony przetarg na obwodnicę Wąchocka, którą Platforma Obywatelska i PSL wykreślały z listy dofinansowania. Jeśli chodzi o dofinansowanie dróg lokalnych, gminnych, powiatowych, to w moim województwie świętokrzyskim wszystkie samorządy, które złożyły wnioski, otrzymały dofinansowanie. Zrobiliśmy trzy nabory po to, aby wszyscy, którzy są przygotowani, mogli z tych środków skorzystać. Niestety niektóre samorządy zarządzane przez PSL nie były w ogóle przygotowane. Dopiero po przejęciu władzy w 2018 r. w tym roku po raz pierwszy po przygotowaniu inwestycji mogły być złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Jakie będą efekty naboru, to zobaczymy.

Ten Fundusz Dróg Samorządowych to ogromne środki i ogromne wsparcie dla naszych mieszkańców, zwiększające bezpieczeństwo zarówno tych mieszkających w małych ojczyznach, jak i tych, którzy poruszają się i przejeżdżają przez nasze miasteczka i gminy. Jeśli mamy stać w prawdzie, to, panie ministrze, podam jeden przykład, jak funkcjonujecie i jak działacie.

Państwo przyszliście, wymazaliście ten węzeł, później dopisaliście. Problem polega na tym, że z węzła można będzie zjechać nie do miasta Łodzi, tylko w kierunku zachodnim, do mniejszych miejscowości, tylko dlatego, że w Łodzi nie rządzicie. To jest przykład trzeciego co do wielkości miasta, które jest przygotowane na tę inwestycję. Mieszkańcy na to czekają, a państwo na złość nie robicie zjazdu z tego ważnego węzła dla mieszkańców Łodzi w kierunku miasta, tylko w przeciwnym kierunku. To jest przykład, jeden z wielu, bo czasu pewnie brakuje. Dziękuję.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i 742) Bardzo proszę pana posła Zbigniewa Dolatę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie pośle, zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawartym w drukach nr 733 i 742. Projekt wpłynął do Sejmu 4 listopada, a w dniu 18 listopada połączone komisje rozpatrzyły przedmiotowy projekt ustawy zawarty w druku nr 733. Projekt ten ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/958.

Z uznaniem wypowiadali się oni o wysokiej jakości projektu rządowego.

Dyrektywa ustanawia zasady przeprowadzania przez państwa unijne ocen przed wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących przepisów regulujących zawody.

Został w niej zawarty obowiązek oceny ww. wymogów, ale nie określono w niej kryteriów tych ocen. Stąd nastąpiła konieczność nowelizacji ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdrażała dyrektywę z 2005 r. Do najważniejszych zagadnień zawartych w ustawie z druku nr 733 należą: po pierwsze, wskazanie zasad, z którymi przepisy muszą być zgodne, w szczególności zasad proporcjonalnego, uzasadnionego i niedyskryminacyjnego charakteru; po drugie, wskazanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych z powyższymi zasadami. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie ocen projektowanych przepisów regulacyjnych oraz monitorowanie ich zgodności. Ponadto określono kryteria, które należy brać pod uwagę przy przeprowadzaniu ocen zgodności wprowadzanych przepisów z ustalonymi zasadami. Wprowadza się również obowiązek konsultacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

W przypadku pracowników ochrony zdrowia szczególnie ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej zasady swobody państw członkowskich w kwestii podejmowania decyzji co do zasadności i sposobu regulacji danego zawodu związanego z ochroną zdrowia. Wysoka Izbo! Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyły ten projekt ustawy i przyjęły jedną poprawkę do art. 6, która stanowi, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Komisje wnoszą o uchwalenie przez Wysoką Izbę rządowego projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu z druku nr 742. Zapraszam panią poseł. Wysoka Izbo!

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Zasada proporcjonalności jest jedną z ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z tą zasadą oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisy krajowe, które mogą ograniczać lub czynić mniej atrakcyjnym korzystanie z podstawowych wolności zagwarantowanych przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinny spełniać cztery przesłanki, tj. być dostosowane w sposób niedyskryminujący, uzasadnione celami leżącymi w interesie publicznym, odpowiednie dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu oraz nie wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. W dyrektywie 2005 nie określono wspólnych kryteriów, które byłyby stosowane przez państwa członkowskie do oceny proporcjonalności wymogów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów. W wyniku wzajemnej oceny między państwami członkowskimi stwierdzono brak jasności co do kryteriów stosowanych podczas oceny proporcjonalności tych wymogów, a także niejednolity poziom kontroli takich wymogów na wszystkich poziomach regulacji. Tak więc dyrektywa z 2018 r. wychodzi naprzeciw wszystkim państwom członkowskim w zakresie zasad przeprowadzania oceny proporcjonalności przed wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących przepisów zawierających wymogi ograniczające dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeprowadzenia obiektywnej analizy szczególnych okoliczności charakteryzujących to państwo członkowskie, które wykaże, że osiągnięcie celów interesu publicznego jest rzeczywiście zagrożone, w związku z czym wymagane jest uregulowanie dostępu do danego zawodu. Zakres oceny powinien być proporcjonalny do charakteru, treści i skutków projektowanych przepisów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych. Ma to być stosowane bez uszczerbku dla innych przepisów zwartych w aktach unijnych dotyczących dostępu do danego zawodu. Zmiany proponowane w projekcie ustawy mają na celu wdrożenie zasadniczych celów dyrektywy z 2018 r. W związku z tym, że przepisy regulacyjne muszą być zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i dyskryminującego charakteru, projekt ustawy przewiduje konieczność zapewnienia ich zgodności z proponowanymi zasadami, a następnie określa mechanizmy służące zapewnieniu tej zgodności, tj. przeprowadzenie ocen projektowanych przepisów regulacyjnych oraz monitorowanie zgodności przepisów regulacyjnych z tymi zasadami - przeprowadzając oceny określone dla projektowanych przepisów regulacyjnych. Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Ustawa nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Projekt nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. Nie wpływa też na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Klub Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt ustawy. Dziękuję serdecznie. Zaskoczenia nie ma, powiem szczerze, ale fajny głos, dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Borys, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/958 z 2018 r. W momencie, kiedy przychodzi moment wdrożenia dyrektywy, nagle okazuje się, że można zachować wszelkie przewidziane normami zasady, które pozwalają na to, aby ustawa mogła być przygotowana zgodnie z zasadami, niepisana na kolanie, niewprowadzona w ciągu jednej doby - po prostu można. I to są te kryteria, które należy uznać, bo ustawa została właściwie skonsultowana, dobrze przygotowana. Poza tym to, co należy docenić, to fakt, że mieścimy się w tym korytarzu dotyczącym terminu, związanym z przyjęciem dyrektywy, a więc roku 2020, uwzględniając COVID - to należy uznać za sprawę ważną, zasadniczą. Państwa członkowskie zobowiązane są do tego, aby dokonać określonych ocen proporcjonalności wymogów, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych i ich wykonywanie, muszą również informować Komisję Europejską. Określony został szereg przesłanek dotyczących niedyskryminacji, uzyskania celów, które leżą w interesie publicznym, wyznaczenia tych celów. Te wszystkie elementy, o których mówi dyrektywa, zostały uwzględnione w projekcie ustawy. Faktycznie jest tak, że państwa członkowskie muszą mieć zakres regulacji, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, szczególnie w wymiarze aspektów zdrowotnych. Ale to, co należy docenić w tej ustawie, a tak naprawdę w intencji tej dyrektywy, to to, że w momencie, kiedy dochodzi do regulacji i ograniczeń wynikających właśnie z określonych zawodów, to wszystkie państwa członkowskie muszą zastosować określoną, tę samą metodologię porównawczą. A więc to jest element istotny, że w momencie, kiedy Komisja Europejska porównuje określone zawody, porównuje je według tej samej metodologii, co zostało uwzględnione w projekcie ustawy. Co jest istotne, można oczywiście od każdej decyzji się odwołać, więc kwestie dotyczące środka odwoławczego zostały również przewidziane - możliwość odwołania do polskich sądów, czy sądów administracyjnych, czy sądów powszechnych. Ale na nas, posłów, obecnie ta dyrektywa i ta ustawa nakładają nowe obowiązki, de facto zmuszą do zmiany regulaminu Sejmu, zmiany regulaminu Senatu, niejednokrotnie zmiany wewnętrznych przepisów różnych korporacji, które mają uprawnienia ustawowe do tego, aby określone zawody regulować, dlatego że każdy, kto będzie składał nowy projekt ustawy, będzie musiał spełnić te same kryteria. A jednym z tych kryteriów jest m.in. kwestia konsultacji. W związku z tym niewątpliwym atutem tej ustawy jest fakt, że dokonamy tak naprawdę uwzględnienia wszystkich reżimów wynikających z przepisów prawa, szczególnie tak naprawdę elementów konsultacji społecznych, poinformowania wszystkich stron.

Poprzemy stosowną ustawę. Podkreślam raz jeszcze, że ta ustawa została dobrze przygotowana na podstawie dyrektywy, i obyśmy mogli pracować nad podobnymi aktami prawnymi według podobnych schematów. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Bogusława Wontora, klub parlamentarny Lewicy. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy pragnę przedstawić stanowisko naszego klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, druki nr 733 i 742. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiany projekt ustawy jest niezbędny do wdrożenia do polskiego porządku prawnego z dwóch powodów.

Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do oceny proporcjonalności wymogów, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów oraz do informowania Komisji Europejskiej o wynikach tej oceny. Po drugie, zmienione prawo w tym zakresie będzie stosowane w sposób niedyskryminujący, będzie uzasadnione celami leżącymi w interesie publicznym, będzie odpowiednie do wymogu zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu i nie będzie wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, a w efekcie obejmie przepisy prawa polskiego określające formy kwalifikacji niezbędne do wykonywania zawodów regulowanych lub wymagania kwalifikacyjne, od których spełnienia jest uzależnione podejmowanie lub wykonywanie działalności regulowanej. Wysoki Sejmie!

Wskazano ministra odpowiedzialnego za materię tej ustawy. Można powiedzieć, że projekt ustawy został przyzwoicie przygotowany. Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie!

Panie Marszałku! Panie Ministrze! W związku z tym, co przedstawiłem, posłanki i posłowie Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy poprą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, druki nr 733 i 742. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zapraszam pana posła Dariusza Klimczaka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Projekt zmiany ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że do tej pory istniał problem braku wspólnych kryteriów, które byłyby stosowane w tym celu przez wszystkie kraje, dlatego od tej pory projektodawcy przepisów będą musieli - będziemy musieli - oceniać ich zgodność z unijną zasadą proporcjonalności, ale także weryfikować, czy mają uzasadniony charakter oraz czy są niedyskryminujące. Uregulowane zostały także wszelkie procedury mające zapewnić zgodność naszych przepisów z unijnymi zasadami, takimi jak obligatoryjność przeprowadzania oceny projektowanych przepisów przed ich wejściem w życie oraz, co jest niezwykle ważne, monitorowania ich zgodności w czasie ich obowiązywania. Nasz klub poprze projektowaną zmianę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, przechodzimy do zadawania pytań. Proszę bardzo, panie pośle. Nie, wiedziałem, że jestem pierwszy. Wiem, że rząd posiada informacje i ciekawe statystyki, dlatego postanowiłem zapytać. A mianowicie chodzi mi o zawody regulowane. Ilu przedstawicieli zawodów regulowanych opuściło Polskę w 2019 r. i jak to się ma do lat ubiegłych? Jakie reprezentowali zawody i do jakich krajów się udali? I odwrotnie, skąd do Polski przyjeżdżają pracować specjaliści, przedstawiciele zawodów regulowanych i przede wszystkim, jakie zawody reprezentują? Bodajże w lipcu pojawiła się informacja, że Komisja Europejska wezwała Polskę i Czechy przed TSUE właśnie w sprawie niestosowania tych regulacji. Czy więcej jest tego typu postępowań, o których wie rząd? Dziękuję bardzo. Pani poseł Mirosława Nykiel, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! To dobrze, że wdrażamy te dyrektywy do polskiego porządku prawnego. To na pewno przyczyni się do realizacji tych wszystkich wartości, wolności, na których w całej Unii wszystkim obywatelom unijnym zależy tak bardzo, a jestem przekonana, że również Polkom i Polakom.

Jak ocenia pan minister przygotowanie polskiego rządu do monitorowania, nadzorowania? Czy spodziewacie się, że tutaj mogą być jakieś przeszkody? Czy uważacie, że wszystko będzie pięknie i gładko. Jakie macie na ten temat zdanie? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana ministra Włodzimierza Bernackiego. Ale ma pan łatwe zadanie, panie ministrze, bo wszyscy pana chwalą, to rzadkie na tej sali. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Urząd piastuję od 4 listopada, tak że jest nadzieja na to. że w dalszej perspektywie czasowej będę zasługiwał na jeszcze lepszą ocenę ze strony również opozycji. Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o bardzo szczegółowe pytanie pana posła Dariusza Klimczaka, to pozwolę sobie przesłać na pana ręce pełną informację dotyczącą właśnie tych liczb odnoszących się do transferu, że tak powiem, osób wykonujących zawody regulowane z naszej przestrzeni w przestrzeń europejską, ale poza granice Polski.

I ten koordynator to jest pani naczelnik jednego z departamentów, w Departamencie Współpracy z Zagranicą, pani Dagmara Dębczak. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. To właśnie jeden z departamentów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w przyszłości Ministerstwa Nauki i Edukacji, będzie sprawował pieczę nad tą stroną koordynującą. Natomiast jeśli chodzi o monitoring, to właśnie ta ustawa wprowadza odpowiedzialność i obowiązek monitorowania, przekłada czy nakłada je na ministra właściwego, który określa te zasady wymagane przy zawodzie regulowanym. Także to wszystko dzieje się w tej przestrzeni, z którą mamy już do czynienia, a więc nie powołuje się tutaj zupełnie nowych bytów. Natomiast, tak jak tutaj powiedziano wcześniej, jak powiedział pan poseł Borys, na posłów, na senatorów, ale i na członków Rady Ministrów spadnie niejako regulaminowy obowiązek konsultowania i uzgadniania treści aktu prawnego z zasadą proporcjonalności, która zawiera się w tej właśnie nowelizacji, ona została dookreślona. Przede wszystkim pragnę na koniec, panie marszałku, Wysoka Izbo, podziękować wszystkim posłom pracującym w dwóch komisjach: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Gospodarki i Rozwoju. Rzeczywiście praca przy tej nowelizacji była przyjemnością. Dziękuję, panie ministrze. Rozumiem, że ustawa jest tak świetnie przygotowana, że pan zrobi nam przyjemność i już nie wejdzie. Proszę państwa, zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie działań podjętych przez rząd w związku z przygotowaniem do drugiej fali epidemii koronawirusa, a także planowanych działań i obostrzeń związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia oraz gospodarki w czasie epidemii, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut.

Stronnictwa Ludowego. Proszę bardzo. Z intelektem u pana marszałka, dowcipem i sprawnością w prowadzeniu nie ma problemu. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Dzisiaj bardzo ważna informacja rządu na temat sytuacji pandemicznej, niestety na temat zaniedbań, bo tak analizujemy to, co się wydarzyło, a bardziej to, co się nie wydarzyło w wakacje, kiedy nie dopełniliście waszych obowiązków, zajmowaliście się czymś innym. W rządzie dostrzegalny jest brak strategii, chaotyczne działania, które bardziej przypominają panikę. Kto na zebraniu głośniej się odezwie, ten wygrywa. Szpitale budowane są w panice, nie mamy strategii walki z epidemią. Dużo jest w działaniach rządu PR-u i propagandy. Nie można siać paniki, ale nie można też zaprzeczać rzeczywistości, bo rząd staje się niewiarygodny. Nie wiem, dlaczego nie potrafiliśmy poprawić funkcjonowania sanepidu przez tyle miesięcy. Obywatele zaczynają się przez to bać. Odmawiają przyjmowania skierowań na testowanie, bo za długo to trwa. Obawiają się kwarantanny. Stąd też jest mniej testów. Nie testujemy pacjentów bezobjawowych, więc nie wiemy jak rozległa jest pandemia. Żyjemy w fikcyjnym obrazie epidemii i fikcyjnie podejmujemy działania. Zanim zaczniecie mnie atakować, że przesadzam, że mówię za dużo, powiem, że to nie są nasze słowa. To są słowa posła klubu Prawo i Sprawiedliwość, członka Zjednoczonej Prawicy. To jest chyba najbardziej wiarygodna ocena, jaką z wnętrza możecie usłyszeć, bo jak opozycja, to możecie się zawsze oburzyć, że to jest spór polityczny. Tu nie ma sporu politycznego. Tu chodzi o zdrowie i życie obywateli, o ratowanie miejsc pracy, o przedsiębiorców, o polską gospodarkę, o naszą przyszłość i przyszłość naszych dzieci. Dlatego domagamy się rzetelnej informacji i skończenia z ciągłą propagandą, PR-em i lansowaniem się na koronawirusie. Jesteście skuteczni i sprawni w blokowaniu dodatkowych pieniędzy dla medyków, w przygotowywaniu dziurawych tarcz, w trzymaniu w zamrażarce ustaw, które mogą pomóc przedsiębiorcom, i zaniżaniu statystyk. Byliście niezwykle sprawni w kampanii Andrzeja Dudy. Członkowie Rady Ministrów wzięli udział minimum w 247 spotkaniach kampanii Andrzeja Dudy, to są ministrowie konstytucyjni, w tym wicepremier i wicepremierzy w 107. To są tysiące godzin, które poświęciliście na lansowanie Andrzeja Dudy, a nie na przygotowanie nas do pandemii. Nie analizowaliście naszych wniosków dotyczących otwarcia szkół. Bezkrytycznie otwarliście szkoły, bo byliście zakładnikami własnych słów, że wszystko wraca do normalności, że epidemia jest już w defensywie, że tak naprawdę ten koronawirus nie jest straszny. Przez pierwsze 2,5 tygodnia listopada zmarło w Polsce na COVID więcej osób niż przez 7 miesięcy pandemii, a pan minister zdrowia mówił dwa dni temu, że możemy się już delikatnie, troszeczkę uśmiechnąć. To jest kpina. Jeśli to mówi jeszcze minister zdrowia, to jest kpina z pacjentów, z lekarzy, pielęgniarek, ze wszystkich, którzy walczą z pandemią. Nie ma naszej zgody na takie podejście i takie traktowanie Polski i obywateli Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo! Domagamy się informacji na temat prawdy o liczbie zakażonych, bo dzisiaj jest za mało testów, testów, które są przeprowadzane, tak jak powiedział pan poseł Sośnierz. Czeka się nawet kilka dni, często mija okres kwarantanny, a wyniku jeszcze nie ma. Domagamy się odpowiedzi, czy stosujecie się do zaleceń komitetu powołanego przez Polską Akademię Nauk przy prezesie Polskiej Akademii Nauk dotyczących zmiany sposobu testowania, żeby testować tych, którzy mają kontakt zawodowy z dużą grupą osób. Co ze sprawami zaangażowania prywatnej ochrony zdrowia? Co z uruchomieniem przychodni i zakończeniem teleporad, które niestety nie zdają egzaminu? Co z informacją wyprzedzającą dla przedsiębiorców? Tak byli zaskoczeni producenci chryzantem, tak byli zaskoczeni właściciele galerii handlowych i sklepów, które się tam znajdują, czasem bardzo małe firmy. Nie prowadzicie dialogu z przedsiębiorcami, nie rozmawiacie, nie informujecie. Wykluczacie kolejne branże, dlatego wnosimy, żeby w kolejnej tarczy anty-COVID-owej, w szóstej tarczy anty-COVID-owej były wpisane nie branże PKD, ale uprawnienia do otrzymywania odszkodowania, by wsparcie było dla wszystkich firm, które po prostu straciły na pandemii. Czy otwarte będą sklepy, galerie? O to dzisiaj wnioskują przedsiębiorcy. Tych pytań dotyczących zdrowia, przedsiębiorczości jest bardzo dużo.

Tym obliczem są zachorowania kolejnych pacjentów, są tysiące osób, które nawet nie wiedzą, że są chore, bo nie mogą się dostać do lekarza ani nie mogą być przebadane. Najgorsze w tym wszystkim są te gigantyczne przyrosty zgonów z dnia na dzień. Wczoraj była czarna środa, dzisiaj jest niestety czarny czwartek. Zajmijcie się swoją pracą. Jesteście za to odpowiedzialni przed prawem, przed Wysoką Izbą, ale przede wszystkim przed rodakami, którzy powierzyli wam stery rządu. Nie zdajecie dzisiaj egzaminu z odpowiedzialności, nie zdajecie egzaminu z pracowitości, nie zdajecie egzaminu z przyzwoitości. To jest poważne oskarżenie, ale ono musi paść, żebyście się opamiętali. Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie pośle. Poproszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana ministra Waldemara Kraskę. Już wiemy więcej. Panie ministrze, proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Jestem senatorem, my troszeczkę dłużej zabieramy głos niż w Sejmie, ale postaram się chociaż w tych kilku minutach stwierdzić i państwu pokazać, w jakim momencie w tej chwili jesteśmy i co zrobiliśmy, bo pan przewodniczący zarzuca nam, że myśmy nic nie zrobili, co oczywiście jest wielką nieprawdą. Nasza strategia rzeczywiście jest inna niż strategia na wiosnę, ponieważ wiedzieliśmy, że nowych zakażeń będzie zdecydowanie więcej. Na wiosnę mieliśmy głównie bazę łóżkową opartą na szpitalach jednoimiennych i to wystarczyło, to się sprawdziło. Jednak wiedzieliśmy, że jesień. Pan jest także lekarzem i wie, że zakażeń jest zawsze więcej. Zwykłej grypy, zwykłych przeziębień, także i koronawirusa jest jesienią zdecydowanie więcej. Do tej strategii włączyliśmy praktycznie całą polską służbę zdrowia poprzez stworzenie bazy łóżkowej opartej na podziale szpitali na tzw. trzy poziomy, poziom pierwszy, drugi i trzeci. W tej chwili podmioty prywatne deklarują ponad 2 tys. miejsc w swoich szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Także organizujemy w tej chwili szpitale tymczasowe, bo wiemy, że epidemia jest nieprzewidywalna i miejsc może niestety nam brakować. Te szpitale są budowane przez wojewodów, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, MSWiA i spółki Skarbu Państwa. Mówił pan, że nasi pacjenci nie mają gdzie się leczyć.

Mamy w tej chwili bufor bezpieczeństwa, to jest ponad 11 tys. wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. Jeżeli chodzi o respiratory, to miesiąc temu mieliśmy ich dostępnych dla pacjentów z COVID 1131, obecnie mamy 2888. Mamy 808 wolnych respiratorów. Na poziomie drugim mamy ich 485, a na poziomie trzecim - 27.

To jest 101 obiektów, to jest ponad 11 tys. wolnych miejsc. To są wszystko miejsca, które czekają na polskich pacjentów. Mam nadzieję, że nie będą musiały być wszystkie wykorzystane. Wiemy, że w przypadku zakażenia koronawirusem tlen jest podstawowym lekiem, którego powinniśmy dostarczyć.

Mówi pan, panie przewodniczący, o testowaniu. Testy są zlecane przez lekarzy, lekarzy szpitalnego oddziału ratunkowego, lekarzy izby przyjęć, lekarzy POZ-u. Oprócz testów genetycznych, które w tej chwili są masowo używane, także dzisiaj jest rozdysponowanych po Polsce prawie 1 mln testów antygenowych. To są testy drugiej generacji, testy, które są porównywalne z testami genetycznymi. One będą dostępne i na izbach przyjęć, i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale także w karetkach pogotowia. Ale myśli pan, że jeszcze powinien mówić czy nie? Zdecydowanie uprości nam to w tej chwili. Mówimy o dostępności i szybkości testów.

Także i pielęgniarki. Także egzaminy lekarskie są w tej chwili przesunięte. Naprawdę robimy wszystko, aby w tej chwili polska służba zdrowia nie tylko posiadała łóżka i sprzęt, ale także miała personel medyczny, który by był dostępny i mógł naszych pacjentów leczyć. Dziękuję serdecznie. Umówiłem się z panem ministrem Niedużakiem, że będzie miał swoje 5 minut dosłownie i w przenośni, jak będziemy kończyli ten temat. Proszę państwa, zaczynamy pytania, ale. Pani poseł Barbara Bartuś, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Witam, pani poseł. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Pan przewodniczący, przedstawiając informację bieżącą, powiedział kilka bardzo ważnych tez. Pierwsze to, co było na końcu. Chodzi o zdrowie i życie, chodzi o przyszłość. Ale drugie, co pan ważnego powiedział, powiedział pan to troszkę wcześniej, że polityka propagandy ma bardzo złe skutki, dlatego odniosę się do tej pana informacji.

Ja wiem, co się dzieje chociażby w moim szpitalu, jak lekarze chorują. To nie tylko dotyka chorych na COVID, tych pacjentów. Przecież mamy też chorych, którzy byli chorzy, są chorzy i niestety często się tak zdarza, że będą chorzy, są wypadki samochodowe. A lekarzy, medyków, pomocy potrzeba. Szanowny Panie Ministrze! Pan przewodniczący zwracał się głównie o testy. Ale dochodzą do nas dobre informacje - informacje, które dają nadzieję.

Zwykle jednak badania nad szczepionkami trwają o wiele dłużej. Tutaj po roku, niespełna roku, dowiadujemy się, że jest szansa. I to byłaby duża szansa, nie tylko w kwestii zdrowotnej, ale też jeżeli chodzi o gospodarkę, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, chodzi o zdrowie, życie, ale i chodzi o przyszłość. Ten lockdown, który zastosowaliśmy na początku, w jakiejś mierze teraz dokucza wszystkim, i nie tylko w Polsce. A jeżeli za granicami też stosują ograniczenia, to przede wszystkim trzymają rynek dla swoich obywateli, bo każde państwo powinno o swoich dbać, więc to też nas dotknie. Dziękuję serdecznie. Oddaję prowadzenie panu marszałkowi Zgorzelskiemu. Popatrzę jeszcze przez chwilę, czy krzesło jest całe, bo mocno siadałem, czy się nie rozwaliło. Mam ostatnio taką sytuację. że rano dowiaduję się, że coś zrobiłem źle. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Szramkę, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Często mamy do czynienia z bałaganem informacyjnym. Na początku Ministerstwo Zdrowia twierdziło, że maseczki nie są potrzebne dla osób zdrowych. Jak widzimy na załączonym obrazku, jednak zmieniło zdanie. Pewnego czasu premier Morawiecki już odwoływał pandemię, mówił, że jest niegroźna, że jest w odwrocie. Jak widzimy, w tym również się mylił. Bywały też przypadki, że to, o czym mówił na konferencjach, trochę różniło się od tego, o czym mogliśmy przeczytać później w rozporządzeniach. Na tym posiedzeniu premier Kaczyński mówił, że opozycja ma krew na rękach, bo wyciąga ludzi na ulice. Ale z Ministerstwa Zdrowia słyszymy, że protesty nie wywołały większej fali zakażeń. Kiedy zadbacie, panie ministrze, o rzetelną i spójną politykę informacyjną? Bardzo często narzekacie na fake newsy, a jak widzimy, to chyba wy najwięcej ich tworzycie. Dziękuję bardzo. Proszę teraz panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, Koalicja Obywatelska, o zabranie głosu.

Chciałam zapytać o dwa obszary, chociaż tych obszarów zaniedbanych, nieprzygotowanych jest naprawdę bardzo wiele, m.in. o szpitalnictwo i inspekcję sanitarną. Przez fakt, że nie przygotowaliście na czas szpitali COVID-owych, polowych, jakkolwiek je nazwiemy, zmusiliście w pewnym momencie szpitale powiatowe do tworzenia, nagłej organizacji oddziałów zakaźnych. Przez to tak naprawdę porzuciły one realizację kalendarza planowanych przyjęć, a niektóre zostały praktycznie całkowicie zamienione w szpitale jednoimienne. Tak jest m.in. w Słupcy i w Środzie Wielkopolskiej w moim okręgu. I dzisiaj mieszkańcy protestują, nie godzą się na takie decyzje, bo boją się, że gdy dostaną zawału, udaru czy zdarzy im się nagły wypadek, pomoc medyczna nie przyjdzie na czas. A więc pytanie: Kiedy szpitale powiatowe przestaną pracować w ramach tylko i wyłącznie ostrego dyżuru i kiedy przywrócicie tam realizację planowanego kalendarza przyjęć? Nie wyobrażam sobie, żeby ten kalendarz nie został przywrócony do wiosny, a tak długo może potrwać druga fala. Druga rzecz to pracownicy inspekcji sanitarnej, którzy zgłaszają niezwykle pilną potrzebę zwiększania liczby etatów, uzupełniania wakatów i zgłaszają, że mają ogromne zaległości zarówno w wykonywaniu wywiadów epidemiologicznych, jak i w zakresie wprowadzania danych do systemu. To sprawia, że te statystyki dotyczące epidemii mogą być kompletnie oderwane od rzeczywistości, co próbował już wam udowadniać młody maturzysta, licząc realnie dostępne statystyki, nie licząc tych, które do systemu nie zostały w ogóle wprowadzone. Kiedy w końcu poprawi się sytuacja w sanepidzie? To nieprzygotowanie rodzi niestety wewnętrzne konflikty, a zwalnianie kierowników oddziałów epidemiologicznych nie jest tutaj żadnym rozwiązaniem, panie ministrze, natomiast tylko i wyłącznie po ten mechanizm dzisiaj sięgacie. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jest też możliwość zadania pytania, nawet jak się jest wnioskodawcą, a tych pytań mamy po prostu bardzo dużo. Pan minister - z racji tego, że jest reprezentantem ministra zdrowia - odnosił się tylko do kwestii zdrowotnej. Nasze pytanie, nasza informacja rządu ma dwie części: zdrowie, ale też gospodarka. Liczymy na pana ministra w drugiej części, na konkretne odpowiedzi. Bo w tym pytaniu, które zadaliśmy, było dużo konkretnych kwestii. Dwa zdania podziękowania dla pani poseł Bartuś. Bardzo dziękuję za docenienie i za zgodzenie się ze mną, że zdrowie, życie, przyszłość są najważniejsze. Chcieliśmy współpracować. Teraz kilka słów o współpracy, jaką proponowaliśmy panu premierowi. Gdy wybuchła pandemia, chodziłem na wszystkie spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta Andrzeja Dudy.

Kolejny raz poszliśmy. Pomimo rozczarowania tym, co zrobił premier, co zrobiliście jako rządzący, poszliśmy na kolejne spotkanie. Zgłosiliśmy propozycję zaangażowania prywatnej ochrony zdrowia i płacenia nie z kieszeni pacjenta, ale z NFZ za leczenie chorób innych niż COVID-19 w ramach prywatnej, czystej, niebiorącej udziału w leczeniu COVID-19 służby zdrowia.

Nie ma odpowiedzi na to. Wysłaliśmy swoich ekspertów na spotkanie z panem premierem. Ani nie uzyskali odpowiedzi na wiele pytań, ani nie zostali zaangażowani. Wyciągaliśmy wielokrotnie rękę. Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią poseł Józefę Szczurek-Żelazko o zabranie głosu. Wysoka Izbo! Pandemia jest jedną z największych tragedii współczesnych czasów i wymaga od nas wspólnych działań. Te działania wspólne powinny być nakierowane na ratowanie życia i zdrowia mieszkańców naszego kraju. Dlatego ze zdziwieniem przyjmuję stanowisko pana przewodniczącego, który mówi, że nie zdajemy egzaminu z przyzwoitości. To państwo przez 8 lat nie zrobiliście nic, aby zwiększyć ilość kadr medycznych, których teraz brakuje. My w ciągu 5 lat potrafiliśmy o 20 tys. zwiększyć liczbę lekarzy, o 15 tys. - liczbę pielęgniarek. Potrafiliśmy zwiększyć wynagrodzenia. Dzięki temu pielęgniarki i lekarze nie opuszczają naszego kraju. Proszę więc państwa, abyście nie mówili, że brakuje nam przyzwoitości. Gdyby te działania były podejmowane wcześniej, dzisiaj sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy mimo tych wielkich problemów staramy się prowadzić nasz kraj lepiej niż wiele innych krajów, które borykają się z pandemią. Proszę spojrzeć na wskaźniki chociażby w Szwecji, w Belgii, w Holandii czy we Włoszech i w Hiszpanii. W krajach, które o wiele więcej środków przeznaczały na ochronę zdrowia, wskaźniki są o wiele gorsze niż w naszym kraju. Przez wakacje, panie pośle, przygotowaliśmy strategię. Przygotowaliśmy nową strategię walki z COVID, przygotowaliśmy nową strategię testowania, przygotowaliśmy nowe szpitale, które teraz w pełni zdają egzamin. To wszystko powoduje, że Polacy mogą liczyć na pomoc.

Ale te miejsca dla pacjentów są zabezpieczane. Każdy wojewoda w zależności od potrzeb [[Dzwonek]] wskazuje odpowiednią liczbę miejsc w szpitalach po to, aby każdy Polak mógł się czuć bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pani minister jeszcze nie pozbyła się tych cech. Prosiliśmy, żeby było mniej propagandy, naprawdę. Otóż, panie ministrze, dokładnie 21 kwietnia w lubelskiej Klinice Chorób Zakaźnych kierowanej - z sukcesem, dodajmy - przez pana prof. Tomasiewicza przeprowadzono pierwszą w Polsce osoczoterapię u pacjenta z ciężkimi objawami COVID-19.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które neutralizują i niszczą koronawirusa, a tym samym blokują dalsze namnażanie się wirusa. Efekty takiej terapii są błyskawiczne. Przypominam: to był kwiecień. Minęło ponad 6 miesięcy, waszych miesięcy, naszych miesięcy, polskich miesięcy. O możliwości nasilenia zachorowań na jesieni mówiono właśnie na wiosnę. A służba krwi dzisiaj czuje się zaskoczona. W związku z tym mam cały szereg pytań, panie ministrze. Oczywiście pewnie nie zdążę wszystkich zadać. Oby tylko pan zechciał odpowiedzieć, a najlepiej uczynić coś w tym zakresie. Czy został opracowany ogólnopolski plan wzmożonego poboru osocza od ozdrowieńców? Czy zostały opracowane jasne wytyczne dotyczące osoczoterapii, które zobowiązują lekarzy do włączenia lub wykluczenia pacjenta z tej terapii? Czy opracowane są jasne kryteria zaniechania pobierania osocza? Czy wydano wytyczne dotyczące przebadania dawców wielokrotnych na obecność przeciwciał anty-COVID-owskich? Czy zostały opracowane procedury przekwalifikowania osocza dawcy z donacji zwykłej na ozdrowieńczą? Czy jest odpowiednia liczba separatorów - bo słyszymy, że ich brakuje - w oddziałach terenowych, w centrach rejonowych? Czy została zakupiona odpowiednia liczba zestawów do inaktywacji osocza? Nie apelujcie do ozdrowieńców o oddawanie, tylko przygotujcie centra do pobierania. Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz głos zabierze pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak pani minister wcześniej z tej mównicy powiedziała, epidemia to wyjątkowy czas, wyjątkowy i niezwykle trudny. To ogromny sprawdzian dla całego społeczeństwa. Szanowni państwo, przypominam sobie, jak na początku poprzedniej kadencji płynęły słowa krytyki w stosunku do pana ministra Antoniego Macierewicza, z którego to inicjatywy powstały Wojska Obrony Terytorialnej.

Chciałabym spytać pana ministra, czy ma taką informację, ilu żołnierzy zostało w tym zakresie przeszkolonych. Kolejna rzecz, o którą chciałabym spytać, to kwestia przeszkolenia pań pielęgniarek w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Szanowni państwo, w Polsce na ponad 200 tys. pielęgniarek czynnych zawodowo - konkretniej mamy chyba 226 tys. pań pielęgniarek - 34 tys. posiada kwalifikacje w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Panie ministrze, czy prawdą jest, że jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie, czyli czy mamy najwięcej przeszkolonych pań w tym zakresie wśród wszystkich czynnych zawodowo pań pielęgniarek? Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Monikę Wielichowską, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Szukają ich przede wszystkim seniorzy. Szukam też ja, wchodząc, pytając, i co chwilę słyszę: Nie ma. Może będą. Były trzy.

W tym samym czasie dolnośląski wojewoda niszczy dobrze wypracowany proces pobierania wymazów w kierunku koronawirusa. Przykład powiatu kłodzkiego, panie ministrze. Zadania zostały przekazane Wojskom Obrony Terytorialnej. Czy pan, panie ministrze, wie, że dziś zdarza się, że pacjenci oczekują ponad 10 dni na pobranie wymazu? Kiedy robiła to karetka ZOZ-u w Kłodzku, nadzorowana przez starostę kłodzkiego, oczekiwali dzień, teraz - 10 dni. Wie pan, panie ministrze, co wtedy robią ci pacjenci?

W związku z tym chcę zapytać - myślę, że odpowie mi pan na piśmie, nie tutaj, bo to są dosyć szczegółowe dane - ile testów w kierunku koronawirusa wykonywanych jest dziennie na terenie powiatu kłodzkiego właśnie przez WOT i jaki jest czas oczekiwania na wymaz w przypadku mobilnej karetki. Na koniec chcę zapytać, kiedy lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności laboratoryjni i wszyscy ci, którzy na pierwszej linii frontu walczą z koronawirusem, [[Dzwonek]] otrzymają przegłosowane w parlamencie, podpisane przez prezydenta dodatki do pensji. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Na początku mała uwaga dotycząca wypowiedzi pani minister Szczurek-Żelazko. Wnioskuję po niej, że pani podziela opinię pana marszałka Terleckiego, który stwierdził, że polska służba zdrowia uchodzi za najlepszą w Europie. Skoro tak jest, to proponuję, żebyście podzielili się tą opinią z Polakami, szczególnie tymi z Tarnobrzega, którzy chcąc odebrać receptę, musieli uderzać kijem o parapet. Chętnie zapoznają się z waszą opinią.

Teleporady muszą zniknąć, nikt nie chce z nich korzystać. Ludzie rezygnują, idą do prywatnego gabinetu i tam oddają swoje ciężko zarobione pieniądze. Państwo powinno refundować taką wizytę. Kiedy nie mogę się dostać do publicznego systemu ochrony zdrowia, NFZ powinien mi zapłacić za tę wizytę. Wiem, że ministerstwo zrobiło pierwszy krok w przypadku pacjentów COVID-owych. Wystarczy zrobić drugi krok. Właśnie to jest pole, na którym możemy współpracować. Naprawdę Polacy się tego domagają. Druga sprawa: sanepid. Nie chce mi się wierzyć, że nie pracujecie państwo nad zmianami w sanepidzie. One są konieczne. Mam nadzieję, że dzisiaj pan minister przynajmniej dwa zdania na ten temat powie. To samo, jeżeli chodzi o wzmocnienie pozycji opiekunów medycznych. Ta grupa zawodowa najczęściej jest przy ludziach od samego początku, od przyjścia do szpitala do wyjścia ze szpitala. Niestety często także jest, że jako jedyni są do ostatnich chwil tego pacjenta. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku chciałam podziękować Ministerstwu Zdrowia i wszystkim ministrom, którzy pracowali, żeby zadbać o zdrowie Polek i Polaków i ratować gospodarkę. Na wiosnę obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, z którą zmaga się cały świat. Jest wiele bardzo cennych inicjatyw z Ministerstwa Zdrowia przeprowadzonych tak, aby po prostu Polacy nie ponosili konsekwencji zdrowotnych. Zostały przeprowadzone w sposób perfekcyjny. Ja bym apelowała do naszych przeciwników, aby używali mniej polityki, a więcej merytoryki. Sanepid w powiecie tarnogórskim został zlikwidowany. I teraz, kiedy były problemy, to pracownicy sanepidów pracowali praktycznie 24 godziny na dobę. Za to chciałam ministerstwu podziękować i prosić o przeanalizowanie, czy nie warto by było wrócić do tego, aby we wszystkich powiatach ziemskich były sanepidy. Teraz jest czas na weryfikację, na dyskusję.

Wiem, że można krytykować, ale, szanowni państwo, zdrowie nie ma barwy politycznej. Apeluję: opozycjo, proszę współpracować, nie przeszkadzać, nie organizować różnego rodzaju przemarszów, które tylko potęgują wzrost zachorowalności. To, co się działo na przestrzeni ostatnich 4 tygodni, to było niewybaczalne. Razem, szanowni państwo, Wysoka Izbo, zadbajmy o zdrowie wszystkich Polek i Polaków. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Mroczka, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Nasz kraj zmaga się z wielkim zagrożeniem w postaci pandemii koronawirusa. Dramatycznie wzrasta liczba zakażonych i ofiar śmiertelnych. Niestety system ochrony zdrowia nie został przygotowany na jesienną falę zakażeń. Występują coraz większe trudności w dostępie do leczenia szpitalnego. Chorzy niekiedy przez wiele godzin wożeni są od szpitala do szpitala w poszukiwaniu wolnego miejsca. Konieczne jest pilne zwiększenie liczby miejsc szpitalnych poprzez tworzenie szpitali tymczasowych. Niestety rząd karygodnie zaniedbał swoje obowiązki w tym zakresie. Do tworzenia szpitali tymczasowych przystąpiono dopiero w październiku w obliczu wielkiej fali zakażeń. Tymczasem w Polsce zaplanowana jest i utrzymywana baza szpitali tymczasowych, ponad 900 szpitali tymczasowych. Te plany są corocznie aktualizowane. Nie słyszałem, żeby któryś z tych szpitali został uruchomiony. To są tzw. zespoły zastępczych miejsc szpitalnych.

I jeszcze słowo na temat wojska.

Proszę teraz pana posła Andrzeja Grzyba, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panowie Ministrowie! Może najpierw zapytam o rzecz, o którą proszą przedsiębiorcy. Pytanie: Czy jest przewidziana renegocjacja obecnych warunków funkcjonowania poszczególnych branż i ewentualnie ich, że tak powiem, kwestii otwarcia czy minimalnego otwarcia, po to, żeby te branże po prostu nie umarły? Kieruję to akurat do pana wiceministra. Natomiast chciałbym podziękować panu ministrowi. Siłą rzeczy to jest skrótowa informacja, trudno jest odpowiedzieć. My nie twierdzimy, że wszystko jest złe, że wszystko, co się dokonało, jest złe, np. decyzja o tym, żeby włączyć POZ-y w tę działalność, to była najlepsza decyzja, jakiej mogliśmy oczekiwać, a w chwili obecnej oczekiwalibyśmy, żeby POZ-y. zrezygnowały w dużej mierze z porad telefonicznych, żeby się otwarły na pacjentów, bo pacjenci tego oczekują.

Coś z tym trzeba by było zrobić, bo szpitale po prostu nie wytrzymają tych stawek.

Czy korzystaliśmy z pieniędzy europejskich na zakup urządzeń do plazmaferezy, do separacji osacza, jako polskie centra krwiodawstwa, ponieważ taki kontrakt, takie zapytanie zostało rozpisane dla krajów członkowski Unii Europejskiej? Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pytanie ważne szczególnie w sytuacji epidemii koronawirusa, dlatego przychodząc na salę plenarną, miałam nadzieję, że będzie merytorycznie. No niestety, zawiodłam się po raz kolejny. Mimo wszystko, szanowni państwo, cieszy to, że po 8 miesiącach od wybuchu epidemii - myślę o tej pierwsze fali - posłowie opozycji wyrażają swoje zainteresowanie sprawami zabezpieczenia zdrowotnego, a także gospodarczymi, szczególnie jeżeli przy pierwszej fali epidemii głosowali przeciwko tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Słucham dzisiaj posłów opozycji, którzy mówią: Jak to, nie mamy jeszcze szczepionki na koronawirusa, a już pan premier dystrybuuje, już robi plany? No tak, proszę państwa, dlatego że na tym polega odpowiedzialna praca rządu i odpowiedzialna praca premiera, żeby pewne rzeczy czynić z wyprzedzeniem. Jeśli to robimy, to państwo mówicie, że za wcześnie, a z drugiej strony, jak przygotowujemy szpitale tymczasowe i łóżka COVID-owe dla pacjentów, to ja z kolei słyszę od posłów opozycji: No tak, ale one nie powinny stać puste. To się państwo zastanówcie, bo one właśnie powinny stać puste.

A państwo mówicie: No nie mogą stać puste. Cieszymy się, że są firmy, które mówią, że ich szczepionki mają 90%, a nawet ponad 94% skuteczności. I chcemy, rzeczywiście, aby jak najwięcej Polaków zdecydowało się na szczepienie. Ale mamy też grupę Polaków, która nie chce się szczepić, bo boi się tych szczepień, a wręcz boi się, że te szczepienia będą obowiązkowe, mimo że pan premier Morawiecki zapewniał, że Polacy nie będą zmuszani (Dzwonek), mimo że mówił o tym minister zdrowia. Bardzo proszę, panie ministrze, żeby pan jeszcze raz powiedział, jak to będzie wyglądało, jakie mamy zabezpieczenie i czy faktycznie Polacy mogą być spokojni, że nie będą to przymusowe szczepienia. Choć mam nadzieję, że jak najwięcej osób uda się do nich przekonać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od początku walki z pandemią koronawirusa mamy do czynienia z dramatyczną wręcz nieudolnością obecnego rządu i kompletnym brakiem strategii.

Miarą braku przygotowania rządu do walki z tą pandemią jest to, że wielu lekarzy i wiele szpitali prosi o wsparcie, takie jak batoniki, środki czystości. Pomagamy i Polacy pomagają, starają się być solidarni. Natomiast mam trzy konkretne pytania. W ogóle mamy bardzo gwałtowny, dramatyczny wzrost śmiertelności. To po pierwsze. Po drugie, czy macie zamiar wprowadzić jakąś strategię w celu zwiększenia liczby testów, bo wiecie przecież doskonale, że wykrywanych przypadków zakażenia koronawirusem jest dużo mniej niż realnych przypadków, bo przecież wiele osób choruje bezobjawowo? Gdybyśmy wiedzieli, że więcej osób przeszło zakażenie koronawirusem, moglibyśmy od tych osób też pobierać osocze, które jest szczególnie ważne. Trzecie pytanie. W Poznaniu pojawiła się informacja o bardzo trudnej sytuacji w szpitalu im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej, co wynika z dramatycznych braków kadrowych i jest charakterystyczne dla większości szpitali. Rozwiązać te problemy można dzięki m.in. takiej pomocy, jaka była zaproponowana w ustawie COVID-owej, [[Dzwonek]] jeśli chodzi o wsparcie dla medyków, która została także podpisana przez prezydenta, a jeszcze przez premiera nieopublikowana. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Zdrowie i gospodarka to tak naprawdę dwa najważniejsze tematy. I mam pytanie dotyczące właśnie gospodarki i przedsiębiorców. Wielu małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców skorzystało z pomocy kierowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale też przez urzędy marszałkowskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i były tam deklarowane etaty w przypadku tworzenia bądź rozwoju tych przedsiębiorstw. Te etaty trzeba utrzymywać odpowiednio 2 bądź 3 lata od wypłaty drugiej transzy, ostatniej transzy płatności.

z wielu powodów. Oczywiście, ministerstwo rolnictwa miało taki aneks przygotować. Czas biegnie, od lipca wzór aneksu się nie pojawił, urzędy marszałkowskie takiego wzoru nie otrzymały. Rozumiem, że karuzela się kręci, w ministerstwie rolnictwa jeden minister donosi na kolejnego, później zrzuca winę na poprzednika, ale przedsiębiorcy czekają na ten wzór i czekają na pieniądze, które za chwilę być może będą musieli zwracać, bo jeśli nie aneksują umowy, to za chwilę wasze służby będą ich z tego rozliczać. Więcej działania, mniej polityki.

Dziękujemy bardzo. Teraz proszę pana posła Krzysztofa Lipca, Prawo i Sprawiedliwość, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zdrowie i gospodarka - to na pewno łączy nas wszystkich w tej Izbie, ale to są tylko słowa.

Proszę szanowną opozycję, żeby zechciała to docenić. Dzisiaj w Polsce jest 40% wolnych łóżek dla chorych na COVID, dzisiaj w Polsce jest 28% wolnych respiratorów.

Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Macieja Laska, Koalicja Obywatelska, o zabranie głosu.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Potraficie wiele zdrożnych rzeczy, ale niestety nie potraficie zarządzać. Uwielbiacie słowo: narodowy, ale pierwsze, co wam przychodzi do głowy, to lockdown. Średniej wielkości firma czy organizacja pozarządowa buduje strategię swojego rozwoju i zarządza ryzykiem i kryzysem. Moglibyście się od takiej firmy wiele nauczyć, ale niestety tej lekcji nie odrobiliście. Zarządzanie przez was krajem to jak pilotowanie samolotu przez osobę, która nawet nie ma prawa jazdy kat. B. Niemal 60% Polaków źle ocenia przygotowanie rządu do walki z drugą falą koronawirusa. Dlaczego? Chaos i permanentne gaszenie pożarów. W szpitalach nie ma personelu, brakuje tlenu, karetki jeżdżą po całym województwie, nie mając komu przekazać pacjentów. W przepełnionych powiatowych szpitalach pacjenci całymi dniami czekają na SOR-ach na przyjęcie. W tym czasie szpital narodowy świeci pustkami. W związku z tym chciałbym zadać pytania: Czy rząd przygotował plan zarządzania ryzykiem związany z drugą falą koronawirusa, a jeżeli tak, to kiedy?

Co było przyczyną wstrzymania budowy szpitala kontenerowego przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie?

Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Paszyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie!

I to nie jest, panie pośle, lipiec, wkładanie kija w szprychy, tylko informacja, która powinna być dla was czerwoną lampką. Kilka pytań. Co planuje resort zdrowia, żeby zwiększyć system badania? Bo pan dobrze wie, jakie są dzisiaj konsekwencje. Ludzie, mając w perspektywie tygodniowe oczekiwanie na testy, po prostu ich nie robią, chorują, zarażają dalej.

Dlaczego dzisiaj są niedobory leku Remdesivir?

Proszę o statystykę, na ile łóżek dzisiaj na oddziałach COVID-owych przypada jeden lekarz. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Ewa Szymańska, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Aż się zepsujesz”

Nawet ci wszyscy antymaseczkowcy, którzy demonstrowali swoją postawę, że nie ma koronawirusa, też się już o tym przekonali.

Bezobjawowo zupełnie, ale musiałam być najpierw w kwarantannie, później w izolacji. Zrobiłam sobie późnej test na przeciwciała, których nie mam. Mam pytanie w związku z tym, bo trochę na ten temat czytałam: Jak to jest z tymi testami i wymazami w przypadku koronawirusa? W jakim stopniu one są pewne co do swoich wyników?

Dziękuję bardzo. Proszę panią poseł Monikę Rosę, Koalicja Obywatelska, o zabranie głosu.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po pierwsze, chciałabym zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby zgonów w Polsce.

Te 12 tys. zgonów to są zgony, ukryte ofiary epidemii. Stąd moje pytanie: Czy państwo dedykujecie seniorom specjalny program ochrony, tak żeby ułatwić im dostęp do lekarza w dobie koronawirusa? Te teleporady czy też dostęp przez nowoczesne środki komunikacji jest dla nich często utrudniony, bo nie mają telefonu, bo nie mają Internetu, nie korzystają, boją się wyjść z domu. Czy mają państwo jakiś specjalny program dedykowany DPS-om, gdzie jednak bardzo często dochodzi do stworzenia ognisk zachorowań? Państwo mówicie o dodatkowych wolnych łóżkach, natomiast te łóżka tworzone są kosztem łóżek w normalnych szpitalach powiatowych. Pacjenci narzekają na brak dostępności, karetki stoją w kolejkach, SOR-y są przepełnione. Epidemia nie jest czymś nowym.

To jest duży problem. Czy państwo monitorujecie te braki w szpitalach? Po raz kolejny, tak jak na początku pandemii, ludzie muszą się zbierać i do szpitali dostarczać rzeczy, które są im po prostu niezbędne. Kwestia szczepionek. Chciałabym spytać, czy jeśli już będzie ta nasza wymarzona szczepionka, jaki będzie system wsparcia, szczególnie grup medyków, osób starszych. Czy także osoby z niepełnosprawności mogą liczyć na pierwszą kolejność, jeśli chodzi o szczepienia? Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Jarosław Rzepa, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Pierwszy temat. Mówicie państwo, że tak bardzo wspieracie gospodarkę. To ja wam dam konkretny przykład. W tym miesiącu chcecie pozbawić pracy 201 stoczniowców w Świnoujściu. Proszę o interwencję. Oni mają 120 km każdego dnia dojeżdżać do pracy. Taka jest państwa propozycja. Taka jest propozycja Skarbu Państwa w dobie kryzysu i koniunktury na remonty statków. Państwo likwidujecie przemysł stoczniowy, mówiąc o tym, że będziecie go odbudowywać. Drugi temat. Szanowni państwo, przed nami grudzień, jeden z najważniejszych okresów dla handlu, dla biznesu. Oczekuję jasnej odpowiedzi od pana ministra zdrowia, jaką strategię ewentualnie będzie miało ministerstwo w momencie, kiedy będzie decyzja o tym, żeby to otworzyć zgodnie z projektem, jaki złożyła Koalicja Polska, jeśli chodzi o wszystkie niedziele. Szanowni Państwo!

Ci ludzie często mają po kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego miejsca, w którym mogą oddać krew.

Bardzo prosiłbym o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy powiaty oznaczone kolorem zielonym, żółtym, a gdzieniegdzie czerwonym. Dziś wydaje się, że mijamy szczytowy punkt drugiej fali koronawirusa, o czym może świadczyć niewielkie zahamowanie gwałtownego wzrostu zachorowań, choć mówię to z dużym zapasem ostrożności. Myślę, że na dzień dzisiejszy takie środki zaradcze jak zachowanie dystansu społecznego, samodyscypliny, noszenie maseczek i dezynfekcja są skutecznym środkiem w walce z pandemią. Ale nie brak też opinii, że przed nami, jeśli nie trzecia fala, to kolejne fale epidemii koronawirusa. Dlatego chciałbym zapytać, czy jest wiadomo, z jaką skalą zachorowań możemy mieć do czynienia w przyszłości i czy dotychczasowe metody zaradcze będą wystarczające. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz panią poseł Joannę Jaśkowiak, Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Miałam przygotowanych kilka pytań, ale myślę, że ograniczę się do jednego. Jesteśmy świadkami niesamowitej polityki pieniężnej w sektorze zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił, w jaki sposób będzie pokrywał koszty leczenia pacjenta chorego na COVID-19. Okazuje się, że różnice pomiędzy różnymi miejscami, do których trafi pacjent, mają przede wszystkim wymiar pieniężny i sięgają nawet kilkuset złotych w przypadku poszczególnych placówek. To jest jawne nadużycie. Jak inaczej można nazwać to, że tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym otrzyma refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości ponad 1000 zł za dobę pobytu jednego chorego, podczas gdy pacjent z tym samym schorzeniem leczony w stacjonarnej placówce wyceniony został tylko na 330 zł?

Jeszcze inaczej wyceniane jest leczenie w prywatnych szpitalach, gdzie narodowy fundusz zapłaci 500 zł. Trudno oprzeć się wrażeniu, jakoby szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym był wybitną placówką leczącą najciężej chorych, wymagających drogich leków i zastosowania specjalistycznych procedur.

W sytuacji tak wysokiej wyceny świadczenia, jak minister zdrowia wytłumaczy niedawne obniżenie tej wyceny z 530 zł do 330 zł w szpitalach stacjonarnych i czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zmniejszyć różnicę w wycenie tych samych świadczeń w różnych placówkach leczniczych? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Dziękuję bardzo. Czy jest na sali pani poseł Anna Paluch?

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Można to poprawić i myślałem, że taki będzie ton pana wypowiedzi. Powiem panu szczerze, że nawet nie dziwi mnie dzisiaj to, że pan powiedział, że MON buduje jeden szpital i że pan nie potrafi go wskazać.

Nie ma po prostu lekarzy.

Dyrektorzy pytają, dlaczego pielęgniarki z wykształceniem średnim z krajów spoza Unii Europejskiej nie mogą pracować w ich szpitalu. Wojewodowie otrzymują informacje od starostów, że mają budynki po szpitalach, które dzisiaj nie są czynne, że można z tej bazy skorzystać. Z ilu takich budynków, panie ministrze, skorzystaliście państwo, żeby można było tam prowadzić szpitale zastępcze COVID-owskie? Bardzo dziękuję. Szanowni państwo posłowie, chciałbym poinformować, że zbliżamy się do końca regulaminowego czasu przewidzianego na zadawanie pytań, ale aby umożliwić zadanie takich pytań wszystkim państwu, proponuję, aby skrócić czas pytania do 1,5 minuty, i wtedy wszyscy się zmieścimy. Zgadzamy się? Zatem proszę o zabranie głosu panią poseł Teresę Pamułę, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.

Dziękuję tym wszystkim, którzy cicho na salach sprzątają, wynoszą, myją, karmią, wszystkim paniom i panom, tym cichym i spokojnym, za tę posługę. Dwudziestego pierwszego mamy Dzień Pracownika Socjalnego. Chciałabym też podziękować wszystkim, którzy opiekują się w różnych miejscach różnymi osobami, w różnym stanie.

Chciałabym też powiedzieć, że nieprawdą jest, jak wybrzmiało na tej sali, że czekamy na testy 5 czy 6 dni. Na testy czekamy ewentualnie kilka godzin. Dziękujemy bardzo. Proszę teraz pana posła Grzegorza Rusieckiego, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W marcu w pewien sposób wszyscy błądzili we mgle, w związku z tym dawaliśmy dużą taryfę ulgową. Ale od tego czasu minęło 9 miesięcy i to, że pandemia uderzy ze zdwojoną siłą jesienią, myślę, że chyba dla wszystkich było jasne. W związku z tym chciałbym zapytać, jak rząd, poszczególne ministerstwa wykorzystały ten czas. Dlaczego nie wydano odpowiednich rozporządzeń, które w inny sposób regulowałyby np. kwestie obecności dzieci w szkołach? Dlaczego w ten sam sposób traktuje się szkoły wiejskie, w których uczy się 50 uczniów, a w oddziale jest po siedmioro, dziesięcioro dzieciaków, i szkoły wielkie, które mają po 1000 uczniów, a w oddziałach jest po 25? Jak przygotowano kadrowo służbę pracowników sanepidu, tych, którzy dzisiaj z ogromnym poświęceniem, ale też zmęczeniem wykonują swoje działania? Jak przygotowano służbę zdrowia nie tylko do opieki nad zarażonymi koronawirusem, ale również nad tymi pacjentami, którzy chorują na inne choroby, np. onkologiczne? Pytam o branżę gastronomiczną, turystyczną, hotelarską, kluby fitness. Pytam o kwestie związane z placówkami kultury, o teatry, kina, spółdzielnie mieszkaniowe, które prowadzą domy kultury. Jakie jest wsparcie, jaki jest sens (Dzwonek) tak dużych ograniczeń? Proszę państwa, tych pytań byłoby dużo, m.in. również o kwestie związane z godzinami dla seniora, czy ktoś w ogóle monitoruje, jaka jest efektywność tego. Natomiast oczekujemy rzeczywiście tej zapowiadanej tutaj ze stron rządowych strategii. Gdzie ona jest i w czym się przejawia? Bo jeśli w tym, że ogłaszamy, że zamykamy cmentarze, na dzień przed świętem Wszystkich Świętych, to wygląda to raczej kiepsko. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Krupka jest obecna na sali? Jeżeli nie, to proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława Suchonia. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście dzisiejsza debata była bardzo potrzebna, bo chyba nikt z nas nie spodziewał się, że ten rząd może być aż tak nieudolny, a co więcej - w niektórych elementach wręcz kontrskuteczny, i to wiedzieliśmy zarówno w obszarze gospodarki, jak i obszarze zdrowia. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to chyba nie da się tego określić inaczej niż wszechobecny chaos, decyzje podejmowane na ostatnią chwilę, całkowity brak logiki i konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Można choćby wspomnieć takie proste obszary działalności jak np. place zabaw dla dzieci - te w centrach handlowych mogą działać, a te, które są położone poza centrami handlowymi, nie mogły działać. Przedsiębiorcy, którzy inwestują majątek życia, nagle zupełnie bez podstaw są zamykani. Pomoc ograniczona w zasadzie do okresu przedwyborczego. I Koalicja Obywatelska, i nasza Nowoczesna mówią: uwolnijcie handel w niedziele, dajcie ludziom możliwość pracy. Druga rzecz - ochrona zdrowia. Na pierwszy rzut Agencja Rezerw Materiałowych. Prosty przykład: respiratory. Okazuje się, że przez kilka miesięcy, w czasie wakacji, kiedy był na to czas, agencja nawet nie sprawdziła, czy ma odpowiednie warunki uruchomienia tych respiratorów. Panie ministrze, kwestia osocza. Pytanie, bardzo proszę o odpowiedź na piśmie: Dlaczego w wielu województwach tylko w jednym mieście, w wojewódzkim, można oddać osocze? Drugie pytanie. Myślę, że to jest ważne: Kto upoważnił premiera Morawieckiego do ogłoszenia w miesiącu lipcu końca epidemii? Dziękuję bardzo. Proszę panią poseł Teresę Wargocką, Prawo i Sprawiedliwość, o zabranie głosu.

Dziękuję, panie marszałku. Temat oczywiście jest bardzo aktualny, ponieważ pandemia nas nie opuściła i nie opuści przez najbliższe miesiące, i na pewno zawsze warto jest ten temat podnosić, żeby szukać dobrych rozwiązań. Państwo z opozycji apelujecie o dialog, o przyjmowanie waszych rozwiązań, a z tej mównicy nic innego nie jest mówione, jak tylko: wszystko jest źle. Wszystko jest źle, nie tak trzeba było powstępować, złe decyzje podejmowaliście, jest tragedia. I to jest ta właśnie polityczna narracja powtarzana jak mantra, która nie pozwala na zbudowanie wzajemnego zaufania, żeby faktycznie porozmawiać na temat rozwiązań. Trwa to już dobre pół roku, taka jest państwa narracja i ja osobiście nie widzę otwartego pola do współpracy. Wnioskodawca dzisiejszej informacji powiedział, że błędem było wysłanie dzieci do szkół we wrześniu. Absolutnie się z tym nie zgadzam. 6 mln dzieci i młodzieży w szkołach poniosło ogromne straty z powodu zamknięcia szkół na wiosnę.

Dzisiaj dzieci są w szkołach, szkoły są przygotowane do zdalnego nauczania, wspieramy nauczycieli finansowo, wspieramy szkoły sprzętem komputerowym i już są propozycje, jak w tym roku szkolnym przeprowadzić egzaminy, żeby młodzież mogła je zdać z powodzeniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz pana posła Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska, o zabranie głosu. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie Ministrowie!

Szanowni Państwo! Z panem posłem Jońskim w poniedziałek złożyliśmy w Ministerstwie Zdrowia pismo w sprawie pilnych działań, które powinien podjąć minister w sprawie akcji oddawania osocza. Szanowni państwo, w ciągu ostatnich 2 tygodni mieliśmy 150 tys. nowych ozdrowieńców. Ale ta liczba ozdrowieńców w żaden sposób nie przekłada się na ilość oddawanego osocza. Dzisiaj jeden z tygodników, tygodnik „Wprost”, podał dane, że w regionalnym centrum krwiodawstwa w Warszawie do tej pory osocze ofiarowało 250 osób. To pokazuje, jak małe są moce przerobowe w tej służbie. Panie ministrze, potrzebna jest pilna nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi, tak, żeby stworzyć również zachęty poprzez. bon dla ozdrowieńców, tak aby osoby, które mają trudności z dojazdem do regionalnych centrów, mogły otrzymać zwrot kosztów podróży.

Konsultanci wojewódzcy apelują do ministra Niedzielskiego, m.in. konsultant [[Dzwonek]] wojewódzka z Mazowsza, żeby pozwolił na zakup tego leku przez szpitale, które są włączane do walki z COVID-em. I ostatnia sprawa, panie ministrze, to jest czas, żeby pan tutaj przyszedł i wytłumaczył się, dlaczego przez 7 miesięcy nie egzekwowaliście 70 mln zł od handlarza bronią, od którego chcieliście kupić respiratory. Po 7 miesiącach skierowaliście sprawę do prokuratorii generalnej.

Proszę teraz pana posła Jana Mosińskiego, Prawo i Sprawiedliwość, o zabranie głosu. Wysoka Izbo!

Nasz polski rząd stara się stawiać czoła temu zjawisku, m.in. takim dobrym ruchem jest zwiększanie liczby łóżek i respiratorów.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie widzę na sali pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, zatem prosimy o wystąpienie w trybie zdalnym pana posła Tomasza Latosa.

Wysoka Izbo! W ostatnich tygodniach rozmawiałem z pracownikami i pracownicami poznańskiego sanepidu. Usłyszałem tam przerażające historie. Ludzie pracują od rana do nocy, są poddawani ogromnej presji, nie mają podstawowego sprzętu, brakuje dziesiątek etatów. Tam gdzie potrzebne byłoby 15 osób, w tej chwili pracują dwie. To warunki pracy niegodne tych, od których zależy bezpieczeństwo nas wszystkich. Ci ludzie są wycieńczeni. Jednego dnia na moich oczach karetki pogotowia przyjechały do dwóch osób, które zemdlały z nerwów i przepracowania. Rząd miał kilka miesięcy, żeby przygotować służby sanitarne do drugiej fali pandemii. Niestety nie zrobiono nic. Władza wolała zajmować się sama sobą, a nie bezpieczeństwem Polek i Polaków. W całej Polsce sanepidy mierzą się z problemami. Brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby. Pracownikom nie płaci się za nadgodziny, przez co w tak ważnym czasie muszą odbierać przymusowo wolne. Ten kryzys powoduje głębokie wewnętrzne konflikty. W Poznaniu cenioną epidemiolożkę panią Annę Pawłowską zwolniono z funkcji kierowniczej. Tak właśnie władza szuka kozła ofiarnego, by odwrócić uwagę od własnych błędów. To obrzydliwa podłość. W swoim imieniu z tej mównicy [[Dzwonek]] chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom i pracownicom sanepidu, którzy pracują w pocie czoła, poświęcając swoje życie osobiste, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Jesteście prawdziwymi bohaterami i bohaterkami. Ostatnie zdanie. Rząd proszę o przedstawienie szczegółowego planu działań w zakresie przygotowania służb sanitarnych do drugiej fali pandemii. Jeśli nie weźmiecie się do roboty, druga fala zmieni się w tsunami. Dziękuję bardzo panu posłowi. Tym samym pragnę poinformować, że lista osób zapisanych do głosu została wyczerpana. Zatem proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo proszę, panie prezesie.

Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję za debatę. Liczę jeszcze na odpowiedź pana ministra w sprawach gospodarczych. Trochę danych liczbowych dotyczących sytuacji, z jaką zastała nas pandemia, liczby łóżek szpitalnych. Najpierw liczba szpitali.

Czy pani poseł jest w stanie spokojnie wysłuchać wypowiedzi do końca? Czy to jest kulturalne przerywać komuś? Nikt państwu nie przeszkadzał, jak mówiliście. Słuchałem cierpliwie, czasem nawet różnych nieprawdziwych i głupich rzeczy. Liczba łóżek szpitalnych.

Co z oddziałami i z łóżkami na oddziałach chorób zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych? Rok 2015, kiedy oddajemy władzę - 3209 łóżek. I wy macie czelność mówić, że przygotowaliście nas do epidemii, że wszystko jest dobrze. Dane z wczorajszego dnia. To jest powód do satysfakcji i do tych głosów wdzięczności? Nie mówimy, że wszystko jest źle. Za wieloma rzeczami też głosowaliśmy. Dobry głos pana posła Latosa, to prawda, jemu się udaje prowadzić dialog. Ale też wiele naszych propozycji wniosków było odrzucanych z góry, bo to były wnioski opozycji. Czemu nie chcecie opublikować ustawy, która daje pieniądze medykom? Część z was za nią zagłosowała. Pięknie mówiła pani poseł Pamuła, i zgadzam się, o wdzięczności dla wszystkich pracowników, dla salowych, dla tych, którzy opiekują się, dla różnego rodzaju personelu, czasem nawet nienazwanego, asystentów osób starszych, dla wielu osób technicznych, którzy pracują w szpitalach, w miejscach pomocy. Ale wy im nie chcecie dać lepszego wynagrodzenia. Wczoraj ze szpitala w Morawicy za pośrednictwem pana posła Jarubasa dostałem informację o powołaniu związku zawodowego właśnie personelu pomocniczego. Oni nie są ujęci w podwyżkach, nie chcecie im dać im naszej premii dla bohatera.

Są tam też pracownicy socjalni, którzy są na pierwszej linii frontu. Słowa wdzięczności są ważne, słowa potrafią też uzdrowić, ale za słowami powinny pójść z waszej strony czyny. To wy wygraliście wybory. Możecie, a nie musicie z nich korzystać, ale wy ponosicie odpowiedzialność dzisiaj za rząd. Andrzej Duda tak często mówił o koronawirusie. Co prawda w drugą falę pandemii nie do końca wierzył 6 czerwca, wypowiadając się. Później w połowie września mówił, że epidemia jest pod kontrolą. Nie chciał może powiedzieć wszystkiego, ale dzisiaj już nie otwiera linii z płynem do dezynfekcji rąk. Nie ma Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma spotkań z ministrami, nie ma odpraw, nie ma inicjatyw prezydenckich. Wygrał wybory, tak jest, ale za zwycięstwem wyborczym powinno iść też działanie, a nie tylko mówienie. To niestety pokazuje, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Największe magazyny, czasopisma medyczne, m.in. „The Lancet”, podają, że właśnie szkoły stały się miejscem rozprzestrzeniania się wirusa. To jest smutne. Ja też bym chciał, żeby szkoły były otwarte, ale żeby były otwarte, muszą być bezpieczne. Pan minister Niedzielski sam to przyznał, więc bardzo proszę, panie ministrze, swoich posłów poinformować o tym, żeby nie siali później fake newsów, bo się robi problem. Macie do nas pretensje, że zwracamy wam uwagę, że mówimy, że coś nie działa, że nie było planu pandemicznego, że działacie w chaosie. Wybudowaliście szpitale polowe w trakcie wakacji czy zajmowaliście się kampanią wyborcą? Przygotowaliście plan pandemiczny i pokazaliście, kiedy będą zamykane sklepy, kiedy będą zamykane inne branże gospodarki, przy jakiej liczbie zachorowań? Nie pokazaliście, mówiliście, że nie będzie drugiego lockdownu. On się stał pomimo waszych zaklęć. On wynikał nie z waszego działania, tylko niestety z braku działania. Jeszcze raz wam przytoczę słowa posła Sośnierza. To jest poseł PiS-u, to nie jest poseł opozycji. Do niego też macie pretensję, że wam zwraca uwagę? Szpitale budowane w panice, nie mamy strategii walki z epidemią. Dużo jest w działaniach rządu PR-u i propagandy. Chcę współpracy. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli normalnej współpracy rozmowy, dialogu i porozumienia, szczególnie w tak ważnej sprawie. I patrzcie, ile było z naszej strony zaufania, nawet poparcia pierwszych ustaw COVID-owych, poparcia wielu poprawek, które zgłaszaliście w pracach komisji w różnych momentach. Czy z drugiej strony jest rozpatrzenie naszych projektów? Gdzie jest ZUS, który powinien być dobrowolny dla wszystkich przedsiębiorców, szczególnie w tak trudnym czasie? Naszym obowiązkiem jest przedstawianie takich projektów, to jest nasz obowiązek. Jeżeli zachęcacie do współpracy i mówicie obłudnie, że nie mamy programu, to wam właśnie go pokazuję, to jest nasz program. Wy go nie chcecie realizować. Macie większość, macie do tego prawo, ale nie mówcie nieprawdy, że opozycja nie przedstawia projektów, że nie przedstawia własnych pomysłów, że jest tylko od krytykowania. Tak, jesteśmy od wskazywania błędów. To jest naturalna rola opozycji w państwach demokratycznych, że pokazuje, gdzie leży problem. Niektóre rzeczy do was po czasie trafiają, bo przynajmniej obostrzenia nie były nakładane z godziny na godzinę. Jeszcze jak do tego dojdzie dialog z przedsiębiorcami, Rada Dialogu Społecznego będzie działała efektywnie. Proszę mi nie wskazywać, że jest po czasie, bo każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości także może mówić po czasie. Tak, proszę pani.

Mówię spokojnie, pokazuję wam dane liczbowe, pokazuję wam fakty i pokazuję wam propozycje. Nie obrażajcie się na prawdę. Ona może boleć, ale nie można się na nią obrażać. Szanowni Państwo! Rada Dialogu Społecznego nie podjęła uchwały pomiędzy związkami a pracodawcami popierającej rozwiązania antykryzysowe. To są fakty. Nie było porozumienia i paktu społecznego. Jest potrzebny pakt społeczny, umowa społeczna i wyjście z tej trudnej sytuacji. Pomimo wszystko myślę, że słowa, które mogą nas połączyć na koniec, to są słowa wdzięczności skierowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników sklepów, pracowników komunikacji miejskiej, różnego rodzaju instytucji samorządowych. Do tych wszystkich, którzy od marca walczą na pierwszej linii frontu, na różnych stanowiskach, w różnych miejscach. Dziękuję też tym wszystkim, którzy ciężko pracują w rządzie. Tak. Nigdy w życiu od was takich słów nikt z nas nie usłyszał, ale tym się też różnimy. Bo jeżeli ktoś robi coś dobrze, to zawsze będziemy to doceniać. Na pewno nie mamy problemu z powiedzeniem słów „dziękuję”, „proszę” czy „przepraszam” Dziękuję wam też za tę debatę, chociaż nie zawsze się zgadzamy. Myślę, że to życzenie zdrowia jest skierowane do każdego, niezależnie od tego, czy siedzi po prawej stronie, czy po lewej stronie tej sali, czy bardziej się go lubi dzisiaj, czy trochę mniej. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Teraz proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pana Marka Niedużaka. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! One też siłą rzeczy były pewnie w trochę mniejszym stopniu poruszane niż zdrowotne.

W tym obszarze nie ma jednomyślności w Radzie Dialogu Społecznego, ale ten dialog tam się toczy. Dialog nie oznacza, że wszyscy się zawsze zgadzają.

Zapewne również z tego powodu Polska, jeśli się popatrzy na Unię Europejską, ma drugi najlepszy wynik, jeśli idzie o PKB w tym roku. Bezrobocie znacząco nie spadło.

Natomiast na pewno te środki pomocowe też miały tu swój udział. Było pytanie o to, co zrobimy dla tych branż, które najbardziej cierpią z powodu obecnej sytuacji. Powiem tak: państwo, panie i panowie posłowie, będziecie mieli za chwilę okazję głosować nad ustawą, która dla tych branż przewiduje m.in. zwolnienie z ZUS-u dla każdego pracownika, przewiduje dofinansowanie do etatów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2 tys. zł na miejsce pracy, przewiduje świadczenie postojowe, przewiduje małą dotację w wysokości 5 tys. zł, bezzwrotną dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Panie pośle, zdaję sobie sprawę, że pewnie nie wszystkie z tych wydarzeń trafiają na pierwsze strony gazet, ale one się dzieją. Korzystając jeszcze z minuty, która mi pozostała, powiem tak: ogólnie należy pamiętać, że sytuacja gospodarcza Polski jest w tym momencie naprawdę nie najgorsza. Tak jak mówiłem, mamy spadek w tym roku, ale on jest jednym z najniższych w Europie. Jeśli ona się spełni - ona jest niesamowicie optymistyczna, to jest ponad 6% - to myślę, że naprawdę wszyscy na tej sali będziemy z tego powodu bardzo zadowoleni.

Wydaje mi się, że naprawdę warto go dzisiaj poprzeć i tym kilkudziesięciu branżom objętym projektem pomóc. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Pomimo że tak naprawdę został wyczerpany czas na odpowiedź, oczywiście prosimy pana ministra Waldemara Kraskę o zabranie głosu. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Dużo polityki, może mało merytoryki. Dziękuję za tę debatę, bo myślę, że jest bardzo ważna.

Czas jest krótki, ale odpowiem na kilka pytań, które na pewno są dość ciekawe i dość często się pojawiały. Po pierwsze, kwestia osocza. To było wielokrotnie poruszane. Powiem państwu, że w październiku w Polsce ozdrowieńcy, bo tylko tacy mogą oddawać osocze - które jest bezcennym lekiem właściwie dla pacjentów w ciężkich stanach, jeżeli chodzi o zakażenie koronawirusem - oddali 2634 jednostki. W czasie jednej sesji można oddać trzy jednostki osocza. Ale już w pierwszym tygodniu, czyli w ciągu pierwszych 7 dni listopada, polscy ozdrowieńcy oddali prawie tyle samo, czyli 2600 jednostek osocza. Nasza służba krwi naprawdę, proszę państwa, jest jedną z lepszych nie tylko w Europie, ale myślę, że na świecie, i w tej chwili ilość oddawanego osocza, tego bardzo cennego leku z dnia na dzień zdecydowanie rośnie.

Przypomnę, że na jednego pacjenta potrzeba pięć dawek. Wielokrotnie państwo mówiliście o sanepidzie. Jest to bardzo ważny element walki z pandemią, ale to my zwiększyliśmy ilość etatów, my zwiększyliśmy wynagrodzenia i zwiększyliśmy cyfryzację tej służby.

Rzeczywiście szczepienia, które będą na koronawirusa, to szczepionki, które w tej chwili już firmy farmaceutyczne zapowiadają, mam nadzieję, że pojawią się dość niedługo, są właściwie jedyną metodą, abyśmy wygrali tę walkę z pandemią, żebyśmy przerwali ten łańcuch epidemiologiczny. I jeszcze raz chcę powtórzyć, że te szczepienia będą dobrowolne. Dobrowolne, bezpłatne, chcemy zabezpieczyć szczepionki dla wszystkich dorosłych Polaków w naszym kraju. Chcemy, aby ta szczepionka była szeroko dostępna, chcemy stworzyć taki system dystrybucji tych szczepionek, aby każdy Polak mógł się zaszczepić. Oczywiście wiem, że wielu Polaków jest sceptycznie nastawionych do szczepień w ogóle, dlatego zorganizujemy akcję medialną, aby przekonać Polaków, że ta szczepionka nie tylko jest skuteczna, ale także jest bezpieczna. Bo ta wartość, że nie będzie powikłań po tym szczepieniu, myślę, że jest bardzo ważna. Dlatego chcemy, aby jak największa ilość Polaków wyszczepiła się, bo jest to, jak powtarzam, jedyna metoda, abyśmy przerwali tę epidemię, którą jesteśmy już tak bardzo zmęczeni od tylu miesięcy. Dziękuję bardzo panu ministrowi, którego wypowiedź kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Ogłaszam 3 minuty przerwy.

Wznawiam obrady. Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Stwierdzam kworum. Minuta, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zanim przedstawię mój wniosek, odczytam fragment pewnego wywiadu: Klub Lewicy 2 dni temu próbował przeforsować w Sejmie swój projekt dotyczący imienników na mundurach policjantów oddziałów zwartych. Ten projekt przepadł jednym głosem. Ale po tym, co pokazał wczoraj marszałek Czarzasty, a wcześniej na Strajku Kobiet w Katowicach poseł Lewicy Kopiec, to ja mogę jedynie stwierdzić, że te imienniki to może posłowie Lewicy powinni sobie wprowadzić. To byłby sygnał dla policjantów, że mogą zostać zaatakowani, i to ze strony najmniej oczekiwanej, bo przez parlamentarzystów. Taki czytelny sygnał: uwaga, poseł Lewicy, może nastąpić na ciebie atak. To słowa, szanowni państwo, przewodniczącego związku zawodowego policjantów, nie wiem, czy osoby, która ma niezmierny wpływ na środowisko, nie wiem, czy inspirowane przez kierownictwo Policji, czy też przez resort. Pani Marszałek! Zwracam się do pani z uprzejmą prośbą.

Panie pośle, bardzo dziękuję. Pan o tym doskonale wie. Właściwa komisja przedłożyła opinię w sprawie kandydata na rzecznika praw obywatelskich, druk nr 725. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt dotyczący tej sprawy. Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów, przedłożyło projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj, druk nr 750. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 758. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj (druk nr 750) Proszę państwa posłów o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj 3 grudnia 2020 roku przypada 80. rocznica mianowania pierwszych przedstawicieli konspiracji politycznej w okupowanej Polsce na stanowiska stałych delegatów rządu na kraj. Stanowisko delegata rządu dla terenów Generalnego Gubernatorstwa objął Cyryl Ratajski - prawnik, były minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, zapamiętany przede wszystkim jako wieloletni prezydent Poznania. Delegatem rządu dla ziem wcielonych do Rzeszy Niemieckiej został Adolf Bniński - ziemianin, wieloletni wojewoda poznański, senator, dwukrotny kandydat na urząd prezydenta Polski. Obaj delegaci - stanowiąc ogniwo pośrednie pomiędzy rządem Polski na uchodźstwie a krajem - pracowali na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: koordynowali współpracę polskich stronnictw politycznych na okupowanych obszarach, podejmowali decyzje w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych oraz stali na straży apolityczności wojskowych struktur konspiracyjnych. Ich działalność stanowiła ważny element kształtowania Polskiego Państwa Podziemnego. Adolf Bniński został aresztowany przez Niemców w lipcu 1941 roku i osadzony w więzieniu w poznańskim Forcie VII. Cyryl Ratajski, z powodu złego stanu zdrowia, zmuszony był złożyć dymisję z zajmowanego stanowiska 5 sierpnia 1942 roku. Zmarł 19 października w tym samym roku i został pochowany pod przybranym nazwiskiem na cmentarzu Powązkowskim. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 80. rocznicę powołania Cyryla Ratajskiego i Adolfa Bnińskiego na stanowiska delegatów rządu na kraj składa im hołd i wyraża przekonanie, że dobrze przysłużyli się Polsce. Proszę o przyjęcie tej uchwały przez aklamację. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego: - Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) o punkty: - Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu głosowania w wyborach na Prezydenta RP w 2020 roku za granicą,

Zieloni o punkty: - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sytuacji finansowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ze wskazaniem wydatków poniesionych przez Grupę w 2020 r. w związku ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego wywołanego zamrożeniem gospodarki przez rząd, a także źródeł ich finansowania, - Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat planowanego przez Rząd wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie w tej sprawie nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu głosowania w wyborach na prezydenta RP w 2020 r. za granicą. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosownia nad wnioskiem dotyczącym informacji prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sytuacji finansowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ze wskazaniem wydatków poniesionych przez grupę w 2020 r. w związku ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego wywołanego zamrożeniem gospodarki przez rząd, a także źródeł ich finansowania.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosownia nad wnioskiem dotyczącym informacji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat planowanego przez rząd wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosownia nad wnioskiem dotyczącym informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 709-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Przypadło mi w udziale przedstawienie dodatkowego sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z druku nr 709-A o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druk nr 704. Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r., zgodnie z regulaminem Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 709 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. W drugim czytaniu zgłoszono 99 poprawek.

Dziękuję. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 709. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Informuję, że poprawki nr 35, 40, 49 i 64 zostały wycofane przez wnioskodawców.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wymienionych poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki przyjął. Poprawki od 2. do 82. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy zawierającego zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 3., zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 4., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 9., zechce nacisnąć przycisk.

W 10. poprawce wnioskodawcy proponują m.in. dodanie art. 15gj. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 10., zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 11., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 38., zechce nacisnąć przycisk.

przeciw?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił.

Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 66. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 65., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Poprawki 72., 73. i 75. stały się bezprzedmiotowe. Z poprawką tą łączy się poprawka 92. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 79. i 80. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 78., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 79., zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 80., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 82., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 84., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 85., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 87., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 89., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. W 90. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę terminu wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 90., zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy.